Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji: - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - godz. 9; - Finansów Publicznych wspólnie z Komisją Infrastruktury - godz. 9.30; - Gospodarki i Rozwoju wspólnie z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi - godz. 10; - Finansów Publicznych - godz. 11; - Rolnictwa i Rozwoju Wsi - godz. 12; Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach - godz. 13.30. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani posłanko. Miło tak siedzieć wspólnie w prezydium. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 29. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego (druk nr 1516) Proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Szymona Giżyńskiego o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Bardzo proszę, panie ministrze.

Z satysfakcją przedstawiam państwu projekt ustawy, która jest krótka, wyrazista, konkretna, w najwyższym stopniu oczywista i przez to niekontrowersyjna. Zajmujemy się w tej ustawie rolniczym handlem detalicznym w kierunku dostosowania ustawowych realiów do potrzeb rolników, do coraz wyższych standardów wymaganych na rynku, jak i zapewnienia producentom rolnym większych zysków, większej pewności i możliwości działania.

W pierwszym z nich, można tak powiedzieć, cały kraj, cała Polska jest dostępna dla każdego producenta funkcjonującego w ramach rolniczego handlu detalicznego. Wszędzie może poszukać swojego odbiorcy. I tutaj nie ma znaczenia, czy będzie sprzedawał bezpośrednio dla tzw. końcowego klienta, czy też będzie korzystał z pośrednictwa stołówek, sklepów czy restauracji. Obowiązywały do tej pory pewne konkretne limity, one zostały całkowicie cofnięte, jeżeli chodzi o sprzedaż do końcowego klienta. Tych limitów po prostu nie ma już w tej chwili. Natomiast utrzymane zostały, z pewnych oczywistych względów, limity przy zaopatrzeniu w produkty z RHD stołówek, sklepów czy restauracji. Informacji o tym, o jakie produkty chodzi, jakie to są limity, można oczywiście zaczerpnąć z rozporządzeń, które tutaj są integralną częścią ustawy. Na przykład dla pewnego skojarzenia i usytuowania w realiach można powiedzieć, że rocznie do jednej restauracji można sprzedawać mięso w ilości 2300 kg.

Chcę zakomunikować Wysokiej Izbie - ma to pewne konsekwencje, ponieważ w takich realiach w tym wypadku się obracaliśmy i obracamy - że projekt ustawy został notyfikowany Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej. Zgodnie z obowiązującą procedurą uwagi mogą spływać do 8 listopada 2021 r. Szanowni państwo, końcowa uwaga dotyczy takiej nadziei, że te warunki, które stwarzamy, tak myślę, przy poparciu Wysokiej Izby, ze względu na charakter ustawy, jej cele i bardzo jasne skomunikowanie tych przepisów z rzeczywistymi potrzebami rynku i rolników będą bardzo dobre. I to jest taki cel, że dojdziemy do sytuacji, w której rolnicy w ramach rolniczego handlu detalicznego będą konkurować między sobą. To jest oczywiście już w jakimś sensie faktem, bo w całej tej operacji też jest bardzo ważny aspekt jakościowy, że odbiorcy liczą na żywność najwyższej jakości. To się dzieje, ale w obszarze dystrybucji żywności najwyższej jakości będzie jeszcze lepiej, jeżeli między producentami już wystąpi zjawisko rzeczywistej konkurencji. Myślę, że idziemy razem z państwem, z Wysoką Izbą dokładnie w tym kierunku. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam ogromny zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, druk nr 1516. Procedowany projekt ustawy jest przede wszystkim realizacją zawartej w dokumencie rządowym Polski Ład inicjatywy nazwanej: uwolnienie rolniczego handlu detalicznego. Rząd Prawa i Sprawiedliwości robi zatem kolejny krok w kierunku jeszcze lepszego wykorzystania wprowadzonego w 2017 r. narzędzia dedykowanego rolnikom, narzędzia, które cieszy się wśród nich dużą popularnością, o czym świadczy fakt, iż obecnie w naszym kraju taką formę sprzedaży żywności prowadzi kilkanaście tysięcy rolników. W projekcie ustawy zaproponowane zostały zmiany przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które mają na celu, po pierwsze, powiększenie obszaru, na którym będą mogły być prowadzone dostawy żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. restauracje, stołówki, sklepy - do terytorium całego kraju. Obecnie obszar ten obejmuje województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach RHD, oraz powiaty lub miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa sąsiadujące z tym województwem, przy czym sprzedaż konsumentom finalnym w ramach tej działalności będzie mogła odbywać się tak jak dotychczas na terytorium całego kraju. Takie rozwiązanie umożliwi rolnikom rozszerzenie rynku zbytu wyprodukowanej żywności przy jednoczesnym spełnieniu wymogów z zakresu bezpieczeństwa żywności. Po drugie, w projekcie ustawy zaproponowano zniesienie maksymalnych limitów żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego konsumentom finalnym i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego. Takie rozwiązanie umożliwi rolnikom zwiększenie sprzedaży żywności konsumentom, zmniejszy obciążenia administracyjne związane z prowadzeniem dokumentacji, a ponadto pozwoli na lepsze wykorzystanie przez rolników możliwości zwolnień podatkowych wprowadzanych projektowaną ustawą. Po trzecie, projekt ustawy przewiduje dodatkowe zwolnienie producenta z podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. podwyższenie z 40 tys. do 100 tys. zł kwoty przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnej produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów zwolnionych z podatku dochodowego. Przyjęcie takiego rozwiązania ograniczy liczbę osób obowiązanych do składania pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy, a z drugiej strony umożliwi uzyskanie wyższych dochodów przez producentów rolnych uzyskujących przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych. Podsumowując, efektem proponowanych zmian powinno być zwiększenie możliwości rozwoju działalności rolniczego handlu detalicznego przez rolników poprzez rozszerzenie zakresu odbiorców żywności, np. sklepów, restauracji, stołówek i innych tego typu zakładów z terytorium całego kraju, oraz wprowadzenie nielimitowanej sprzedaży żywności konsumentom, a także powinno to przyczynić się do podwyższenia dochodów producentów rolnych. Przedmiotowy projekt ustawy podlega procedurze notyfikacji Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej, a więc ostatecznie zakres proponowanych zmian zależeć będzie również od opinii Komisji Europejskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej zgłoszonych w ramach tej procedury.

Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pragnę poinformować, że Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie wspierał rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw (Dzwonek) w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego w dalszym toku prac parlamentarnych. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zanim przejdę do oceny znowelizowanych przepisów dotyczących rolniczego handlu detalicznego, najpierw kilka sprostowań. Po pierwsze, wbrew temu, co napisano w uzasadnieniu ustawy, przepisy nie wynikają - cytuję - z dokumentu rządowego Polski Ład. O ile mi wiadomo, rząd Polskiego Ładu, czyli spisu haseł i ładnych obrazków - tak dla przypomnienia wygląda ten dokument - do dzisiaj oficjalnie nie przyjął jako swojego programu, czyli nie jest to program rządowy. A jeśli jest inaczej, to proszę o podanie daty posiedzenia Rady Ministrów, na którym program partyjny Polski Ład został przyjęty jako oficjalny program rządowy. Przestańcie wreszcie zaśmiecać pisma państwowych urzędników sformułowaniami typu: rządowy program Polski Ład. Po drugie, słuchając pana posła sprawozdawcy z Prawa i Sprawiedliwości, można odnieść wrażenie, że proponowane zmiany rozwiążą problemy polskiego rolnictwa, a wieś stanie się krainą mlekiem i miodem płynącą. Otóż tak się nie stanie. Z czego to wynika?

A ile mamy gospodarstw pobierających dopłaty w Polsce? Czyli z dobrodziejstwa rolniczego handlu detalicznego korzysta mniej niż 1% gospodarstw rolnych. Warto o tym pamiętać. Dzisiaj produkcja żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego o wartości do 40 tys. zł jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. W nowelizacji ustawy proponuje się podniesienie tej kwoty do 100 tys. zł. Czy są jakieś ekspertyzy, opinie, które potwierdzają, że ma być to kwota 100 tys. zł?

Wiadomo, że kwoty 40 tys. zł nie możecie utrzymać, bo planujecie zwolnić z płacenia podatku PIT wszystkich obywateli Polski osiągających dochody roczne do 30 tys. zł. Tak więc pozostawienie tych 40 tys. zł dla rolników w przypadku rolniczego handlu detalicznego byłoby groteską. Ten limit musicie podnieść - również z powodu galopującej inflacji.

Dlaczego tak mało? Naszym zdaniem odpowiedź jest prosta: bo rolnicy nie chcą się użerać z waszą biurokracją. Zróbcie coś z tym, a wtedy na pewno kwestie dotyczące rolniczego handlu detalicznego wystrzelą w górę. Przyznacie, że to kwota niewielka. Sam Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa więcej rocznie wydaje na premie i nagrody, trzynastki itd. Oto mamy prawdziwy cud - za niewiele ponad 15 mln zł rząd Prawa i Sprawiedliwości uzdrowi polskie rolnictwo. A dlaczego tak mówię? Bo w waszym Polskim Ładzie uwolnienie handlu detalicznego, czyli tę omawianą przez nas tu i teraz ustawę, wymieniacie jako jedną z trzech najważniejszych zmian, jakie nastąpią w polskim rolnictwie. Pierwsza proponowana to Kodeks rolny, druga to zwrot akcyzy, a trzecia to właśnie projekt ustawy o rolniczym handlu detalicznym. A my pytamy: Gdzie jest skuteczna strategia walki z ASF, gdzie opłacalność produkcji rolnej, gdzie odbudowa całego sektora trzody chlewnej, gdzie holding spożywczy, gdzie powszechne ubezpieczenia? Nie mówimy już o kwestiach związanych ze wzrostem wydatków na rolnictwo do 3% PKB. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska wnoszę o skierowanie niniejszego projektu ustawy do dalszych prac legislacyjnych.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu parlamentarnego Lewicy wobec rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, druk nr 1516. Wyjaśnię najpierw krótko, na czym polega rolniczy handel detaliczny, w skrócie RHD. Jest to specyficzna, funkcjonująca w Polsce od 2017 r., forma handlu detalicznego dedykowana rolnikom. Podstawowym warunkiem prowadzenia RHD jest to, że żywność musi w całości lub w części pochodzić z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Rolniczy handel detaliczny jest korzystny ze względu na zwolnienia podatkowe. Obecnie rolnicy są zwolnieni z opodatkowania przychodów do kwoty 40 tys. zł. W ramach rolniczego handlu detalicznego możliwa jest produkcja, w tym również przetwórstwo żywności na małą skalę, i jej zbywanie konsumentom finalnym, a także lokalnym zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego. W ramach rolniczego handlu detalicznego można sprzedawać surowce pochodzenia roślinnego, np. zboża, warzywa, owoce, zioła, i zwierzęcego, np. mleko, śmietanę, jaja, miód, ale również przetworzoną żywność, np. oleje, chleby, dżemy, soki, przetwory, a także możliwa jest sprzedaż i przygotowywanie posiłków, takich jak pierogi, kopytka, kluski śląskie, knedle itd., itd. Omawiany projekt ustawy zawiera kilka kluczowych zmian w funkcjonowaniu rolniczego handlu detalicznego. Po pierwsze, w projekcie ustawy proponuje się zupełne zniesienie maksymalnych limitów żywności w odniesieniu do sprzedaży konsumentom finalnym i pozostawienie tylko tych limitów, które odnoszą się do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny, np. do sklepów, restauracji czy stołówek. Druga zmiana polega na podwyższeniu limitu przychodów ze sprzedaży zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych: z 40 tys. do 100 tys. zł. Kolejna zmiana to zwiększenie obszaru, na którym mogą być prowadzone dostawy żywności do zakładów prowadzących handel detaliczny, takich jak sklepy, restauracje i stołówki, do terytorium całego kraju. Obecnie obszar ten jest ograniczony do województwa oraz powiatów lub miast sąsiadujących z województwem. Ostatnia zmiana polega na zmianie definicji pojęcia rolniczy handel detaliczny. Jeśli produkt składa się z jednego składnika, definicja pozostaje bez zmian. Zmiana następuje w przypadku żywności zawierającej więcej niż jeden składnik, np. przetworzone produkty mięsne, produkty mleczne, ale również gotowe posiłki. Tu proponowana jest zmiana polegająca na tym, że żywność powinna zawierać co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Co do zasady sama koncepcja uproszczenia sprzedaży płodów rolnych jest potrzebna. Powinniśmy dążyć do skrócenia łańcuchów dostaw i do tego, by rolnicy osiągali wyższe wynagrodzenie za swoją pracę, włożony kapitał i poniesione ryzyko. Ten kierunek jest zgodny z polityką Europejskiego Zielonego Ładu, od pola do stołu, choć trzeba zaznaczyć, że kraje unijne proponują różne rozwiązania. Zwracam jednak uwagę, że proponowane w ustawie zmiany wiążą się też z pewnymi ryzykami. Pierwsze dotyczy finansów państwa, np. zniesienie maksymalnych limitów żywności może rodzić ryzyko, że część żywności będzie sprzedawana w sposób nieuczciwy, bez podatku, nie tylko finalnym konsumentom, ale także sklepom, restauracjom i stołówkom. Zmiana definicji rolniczego handlu detalicznego wydaje się również zbyt daleko idąca. Co np. jeżeli w gotowym posiłku będą tylko polskie rzodkiewki, a reszta to ryż z Chin, soja z USA, mięso i pomidory z Hiszpanii? Według tej definicji ten posiłek będzie można sprzedawać bez podatku. Mam nadzieję, że ta ustawa nie była pisana pod kogoś. Chcę zakładać dobre intencje wnioskodawcy i liczę na poprawienie jej w procesie legislacyjnym. Równocześnie zwracam się do pana ministra z prośbą o przygotowanie rzetelnego porównania dotyczącego tego, jakie rozwiązania prawne funkcjonują w innych krajach Unii Europejskiej, abyśmy na posiedzeniu komisji mogli podjąć dobrą decyzję. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Mirosława Maliszewskiego z Klubu Parlamentarnego. No właśnie - Koalicja Polska. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Bo ono dotyczy tylko gospodarstw małych albo bardzo małych i gospodarstw specyficznie położonych, czyli np. w pobliżu dużych aglomeracji miejskich, a szczególnie w pobliżu ośrodków turystycznych. Taki model sprzedaży bezpośredniej rolniczego handlu detalicznego obserwujemy od kilkunastu lat czy nawet dłużej w krajach Europy Zachodniej.

Wyjaśnijmy jeszcze jedną rzecz. Rolniczy handel detaliczny powinien się odnosić - i ma uzasadnienie tylko w tym przypadku - do produktów przetwarzanych w warunkach domowych czy w warunkach gospodarstwa, bo sprzedaż produktów nieprzetworzonych jest dzisiaj możliwa z gospodarstwa bezpośrednio do wszystkich odbiorców, którzy są na rynku, niezależnie od ich wielkości, potencjału, siły ekonomicznej. I to nie jest obłożone podatkiem dochodowym czy obrotowym, tak jak w tym przypadku. To dotyczy więc tylko możliwości przerabiania produktów na poziomie gospodarstwa. Dlaczego jest takie małe zainteresowanie tym? Z tych powodów, o których mówiłem wcześniej. Żadne gospodarstwo średnie albo duże nie jest w stanie swojej produkcji zagospodarować w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Bo gdzie? Nie ma takiego odbiorcy, który taki specyficzny produkt w takiej ilości byłby w stanie kupić. Teraz o ułatwieniach, które w tej ustawie się pojawiają. Dziwi mnie też, że w dokumencie, który ma być strategicznym dokumentem odnoszącym się do polskiej wsi, działanie kierowane do mniej niż 1% gospodarstw jest wymieniane jako priorytetowe. To są działania o marginalnym znaczeniu dla polskiego rolnictwa. Dzisiaj czas wymaga tego, aby podejmować bardziej radykalne działania niż takie drobne. Rzeczywiście podniesienie limitu zwolnienia z podatku z 40 tys. do 100 tys. dla wielu może być szansą.

To jak gdyby uwiarygadnia te słowa, które przed chwilą wypowiedziałem. Natomiast gdybyśmy połączyli to rzeczywiście z możliwością sprzedaży poza województwem, na terenie którego znajduje się gospodarstwo, i może przeprowadzili też inne działania ustawowe, które by zmuszały dużych odbiorców produktów do tego, aby sięgali po produkt lokalny, produkt pochodzenia lokalnego - takie rozwiązania są w niektórych krajach Unii Europejskiej, np. we Francji - to moglibyśmy spowodować większe zainteresowanie konsumentów, ale także np. sieci handlowych produktami wytwarzanymi w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Oczywiście będziemy zgłaszali propozycje zmian w najbliższym czasie, również w formie projektów ustaw, bo np. warto w ramach rolniczego handlu detalicznego zająć się produkcją nalewek, destylatów i innych produktów na bazie alkoholu, na bazie owoców.

Dziękuję za ten głos panu posłowi z PSL-u. Pan poseł Michał Urbaniak, koło Konfederacja. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Sprzedaż bezpośrednia wśród rolników jest pewną odpowiedzią na wiele problemów małych gospodarstw rolnych, które tym sposobem mogą sprzedawać produkowaną przez siebie żywność na tę niewielką skalę. Wyeliminowanie pośredników przyniesie korzyści zarówno dla samego producenta, jak i dla konsumenta, który jest w stanie ominąć ten cały łańcuch dostaw, kupować produkty dobrej jakości i w szerokiej gamie. Najważniejszym elementem zazwyczaj jest kwestia preferencyjnych i uproszczonych form opodatkowania. To się tutaj pojawia, że ta forma i wysokość przychodu mogą zachęcać rolników do korzystania z niej.

Pamiętamy też, że to jest kropla w morzu potrzeb. To na plus. Nasze wątpliwości natomiast wzbudza zapis, który mówi, że ustawa zmienia nadzór nad produkcją i zbywaniem żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego na kontrolę urzędową tutaj prowadzoną przez sanepid i Inspekcję Weterynaryjną.

Naturalne jest to, że każdy rolnik, który produkuje coś, który przetwarza pewne produkty, chce dać produkt dobrej jakości, bo to jest wtedy jego marka, on to sygnuje swoim nazwiskiem. My ten projekt zasadniczo poprzemy, oczywiście z tymi uwagami, które też będziemy zgłaszać, choć, tak jak mówiłem na początku, to pewnie nie przyniesie radykalnej zmiany, ale zawsze jest coś na plus. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Koła Parlamentarnego Polska 2050 stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. Deklarowanym przez rząd celem projektu ustawy są ułatwienia w zakresie rolniczego handlu detalicznego. W projekcie proponuje się szereg zmian. Po pierwsze, chodzi o zmianę definicji pojęcia „rolniczy handel detaliczny” w celu doprecyzowania pochodzenia składników wykorzystywanych do produkcji w tej formie działalności. Projekt prowadzi także do rozszerzenia obszaru, na którym mogą być prowadzone dostawy żywności. Od momentu przyjęcia tego projektu będzie można to robić na terytorium całej Polski. Ustawa zmierza także do doprecyzowania kwestii pochodzenia składników wykorzystywanych do produkcji żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, a kolejna zmiana to modyfikacja upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia dotyczącego posiadania maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego, co ma skutkować zniesieniem limitów produktów dostarczanych w ramach tej formy działalności. W projektowanej ustawie zaproponowano także podwyższenie z 40 tys. zł do 100 tys. zł kwoty przychodów ze sprzedaży, które są zwolnione z podatku dochodowego. Oczywiście są to generalnie zmiany idące w dobrym kierunku, jednak nie mogę się oprzeć takiemu wrażeniu, że przed chwilą pan minister opowiadał o tym projekcie tak, jakby to był Święty Graal rolnictwa. Tymczasem z rolniczego handlu detalicznego skorzystało zaledwie 12 876 gospodarstw, czyli stosunkowo niewielka grupa rolników. Koszt tych zmian, które proponuje rząd, to zaledwie 15,5 mln zł, choć sam tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości, zakładam, wydaje prawdopodobnie miliony złotych na catering w swojej administracji. Po drugie, nasuwają się wątpliwości, czy tak szerokie ujęcie definicji nie doprowadzi do sytuacji, w której bez podatku będą sprzedawane także produkty pochodzące zza naszej granicy. I to jest dosyć duża wątpliwość. Po trzecie - myślę, że to najważniejsza rzecz - wbrew temu, co, wydaje się, wynikało ze słów pana ministra, ten projekt wcale nie uleczy problemów polskiego rolnictwa. Szalejąca drożyzna, wysoka inflacja, ale także brak odważnych działań w sprawach dotyczących rolnictwa to są rzeczy, za które odpowiada rząd, a które wykańczają dzisiaj polskich rolników. Tych problemów projekt nie rozwiązuje. Ale, tak jak powiedziałem, te rozwiązania, choć wąskie, idą w dobrym kierunku (Dzwonek), więc w imieniu Koła Parlamentarnego Polska 2050 wnoszę o przekazanie projektu do komisji celem dalszych prac. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Właśnie widzę. Niech pan uważa na siebie. Wysoka Izbo! W imieniu koła Kukiz’15 - Demokracja Bezpośrednia mam zaszczyt przedstawić stanowisko koła w stosunku do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. Na wstępie - bardzo się cieszę, że już rozpoczęliśmy procedowanie ustaw, które zostały przygotowane w ramach Polskiego Ładu dla rolnictwa. Zmiany w tej ustawie są bardzo pożądane przez rolników, ponieważ obecnie działające rozwiązania, tak jak słyszeliśmy, są niewystarczające, bo rolnicy na razie masowo się do tego nie garną. Przypomnę również, że już w ubiegłej kadencji Klub Parlamentarny Kukiz’15 przygotował ustawę o sprzedaży bezpośredniej, i dodam, że tu kilka elementów znowu się pojawiło się w tej ustawie. Szkoda, że tak późno, aczkolwiek dobrze, że one są. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze tę ustawę modyfikowali. Ale, co ważniejsze, ta ustawa jest komplementarna z kolejną ustawą, którą będziemy procedowali na kolejnym posiedzeniu Sejmu, czyli ustawą otwierającą miasta właśnie na rolniczy handel detaliczny, tak żeby rolnicy mieli dobre miejsce do sprzedaży swoich produktów, a konsumenci dostęp do smacznych, zdrowych produktów rolniczych.

To jest jeden z elementów, ale to bardzo ważny element dywersyfikujący dochody rolników.

Myślę, że te liczby, które były podawane, niewielkie liczby co do tych rolników, którzy dotychczas skorzystali z możliwości prowadzenia rolniczego handlu detalicznego, w tej chwili przy całym pakiecie tych rozwiązań znacznie się zwiększą, a konsumenci będą powszechnie korzystali z możliwości bezpośredniego kupowania żywności od rolników, bo jest to żywność nieprzetworzona, żywność z produktów najwyższej jakości. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do pytań. Ustalam limit czasu na pytanie - 1 minuta. Mirosław Suchoń, poseł Polski 2050, jak zwykle pierwszy. Bardzo proszę, panie pośle.

Warto pamiętać o tym, że potrzebujemy takiego silnego wsparcia dla rolników, także dlatego że jest to żywność zdrowa, jest to żywność zazwyczaj taka, która dobrze wpływa na funkcjonowanie organizmu. Te zmiany, tak jak powiedziałem w wystąpieniu klubowym, idą w dobrym kierunku, jednakże dosyć niewielka w gruncie rzeczy grupa gospodarstw wykorzystuje tę możliwość. Jakie jeszcze działania rząd zamierza podjąć, żeby jednak stało się to bardziej powszechne, ta bezpośrednia sprzedaż konsumentom? Dziękuję bardzo. Pani poseł Iwona Maria Kozłowska, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Zapraszam. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jeśli stan gospodarki rolnej nie ulegnie poprawie, w polskim rolnictwie pracować będzie za chwilę od 1 do 3% ludności. Dlatego każda zmiana, która może pomóc w wyprowadzeniu z kryzysu polskiej wsi, jest warta uwagi, ale niestety nie takie propozycje. Rozmawiałam na temat tego projektu z rolnikiem, który potwierdził to, co rzeczywiście widzimy, że produkcją żywności na wsi zajmują się przede wszystkim pasjonaci. Są to nieliczni rolnicy z małych gospodarstw, którzy chcą nie tylko utrzymać swoje gospodarstwo, swój majątek, ale mają przede wszystkim wiedzę, pomysł na innowacyjność i na zmianę profilu swojej działalności. Omawiany projekt m.in. doprecyzowuje przepis, iż rolniczy handel detaliczny pozwala na produkcję żywności zawierającej co najmniej jeden składnik pochodzący z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Mój rozmówca pyta, czy nie można po prostu pozwolić rolnikom na produkcję żywności w całości pochodzącej (Dzwonek) ze składników z innych, sąsiednich gospodarstw. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Piotr Borys, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Proszę, Piotrze. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chodzi o to, jak zwiększyć handel detaliczny rolników, aby nie 12 tys. polskich rolników z 1100 tys. gospodarstw, ale setki tysięcy polskich rolników były w stanie produkować żywność i w tym tak naprawdę bardzo krótkim łańcuchu zasilać polskich obywateli, szczególnie obywateli mieszkających w miastach.

Szukajmy takich właśnie rozwiązań, a nie rozwiązań błahych czy niecałościowych. Dziękuję. Panie Ministrze! Rolniczy handel detaliczny to forma sprzedaży, która funkcjonuje od 2017 r. Została wprowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość. W tej formule, pani poseł. Dziś po kilku latach obserwacji ten pierwotny model podlega modyfikacji, m.in. właśnie poprzez poszerzenie, rozszerzenie możliwego rynku zbytu na obszar całego kraju. Dotychczasowe ograniczenie sprzedaży do obszaru województwa było jedną z barier dla rolnika. I moje pytanie: Gdzie ministerstwo rolnictwa widzi inne bariery? Chodzi przede wszystkim o te bariery pozaprawne, których brak mógłby spowodować, że rolnicy chętniej korzystaliby z możliwości, jaką daje rolniczy handel detaliczny. Dziękuję serdecznie. Pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Pan poseł Waldy Dzikowski, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Nie ma.

Koalicja Polska, panie marszałku. Jakaś blokada mózgu, ale sobie zaraz odblokuję. Proszę bardzo. Ale to, o co zapytam, być może panu marszałkowi trochę poprawi humor i poprawi dzień. Pytałem w wystąpieniu klubowym o możliwość produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznego destylatów, nalewek i cydru.

I drugie pytanie, dotyczące produktu, który jest dzisiaj w Polsce wytwarzany czy był wytwarzany, z którym polscy sadownicy wiązali ogromne nadzieje, mianowicie: cydr. Jest to stary polski napój alkoholowy, zwany kiedyś, przed wojną jabłecznikiem, wytwarzany z jabłek, który był wielką nadzieją na zagospodarowanie nawet 100 tys. t jabłek rocznie. W produkcję tego napoju zainwestowało kilkaset gospodarstw w Polsce, które dzisiaj upadają (Dzwonek), jeżeli chodzi o tę produkcję, z tego powodu, że podatek akcyzowy zabił produkcję cydru w Polsce, zabił jego konsumpcję.

Dziękuję serdecznie, panie pośle z Koalicji Polskiej. Bardzo proszę, pani posłanka Dorota Niedziela, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo mówicie, że otwieracie, i bardzo dobrze, przestrzeń, otwieracie możliwości, zwiększacie limity, ale podstawowa rzecz, o której mówimy, to nałożenie na rolników kagańca pod nazwą: kontrola.

Na pewno nie. Panie pośle, proszę to zmienić, będziemy składać taką poprawkę. Ten zapis nie ma sensu, jeśli nałoży się na rolników kontrolę.

W tej ustawie nakładacie na rolników jeszcze jedną kontrolę. Do tej pory (Dzwonek) rolniczy handel detaliczny, czyli sprzedaż bezpośrednia, był nadzorowany. Dziękuję bardzo. Pan poseł Kazimierz Plocke, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Powiem troszeczkę w kontekście tego, co powiedziała pani poseł Niedziela. W uzasadnieniu do projektu ustawy napisaliście państwo, że celem tych nowelizowanych przepisów ma być ułatwienie prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. Natomiast z drugiej strony z tych przepisów, które proponujecie państwo, wynika, że nakładacie dodatkowe obowiązki na producenta żywności poprzez kontrolę inspekcji sanitarnej i inspekcji weterynaryjnej.

Czym innym jest kontrola, czym innym jest nadzór. Dziękuję serdecznie. Zacznę od: dziękuję, pan wie, za co. Szanowna Izbo!

Ta ustawa będzie zachęcała.

Pan poseł Jan Szopiński, klub parlamentarny Lewica. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Powiedzieliście tutaj państwo, że tą ustawą rozpoczynamy Polski Ład dla rolnictwa. A ja chciałbym zapytać, czy nie jest tak, że mówicie o pewnych mechanizmach pozwalających rolnikom na prowadzenie działalności pozarolniczej, licząc na to, że rolnicy zajmą się działalnością gospodarczą, co odwróci ich uwagę od faktycznych problemów polskiego rolnictwa. Chciałbym zapytać, czy przydrożne stragany, na które rząd wysyła rolników, będą musiały posiadać kasy z łącznością on-line. I drugie: Czy rolnik będzie zwolniony z obowiązków sanitarnych, którym podlegają inni producenci? Szanowny Panie Ministrze! Dziękuję bardzo. Panie Ministrze!

Dlaczego nałożono urzędową kontrolę do nadzoru nad rolniczym handlem detalicznym zamiast nadzoru? W czym ten nadzór był gorszy?

Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przedłużył pan o pół minuty, panie pośle. No właśnie. Bardzo proszę. Pani poseł Teresa Pamuła. Pan poseł Krzysztof Grabczuk, Koalicja Obywatelska. No właśnie. Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rolniczy handel detaliczny wciąż osiąga bardzo niski poziom. Chociaż dotyczy niewielkiej grupy rolników, to warto o tym rozmawiać, warto wspierać tego typu rozwiązania.

Drugi element: absolutnie powinniśmy dążyć do tego, by wspierać zdrowe produkty ekologiczne. Z uporem maniaka będę przypominał, że wciąż powinniśmy nad tym pracować, tworzyć warunki, żeby w Polsce powstawało coraz więcej gospodarstw ekologicznych, ponieważ w tym zakresie jest przyszłość. Oczywiście ten limit, który był, czyli 40 tys., jest zbyt niski.

Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. W związku z tym jesteście absolutnie usprawiedliwione, w nagrodę dopisujemy was na koniec.

Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. Pytania moje do pana ministra.

Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Janusz Kowalski, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Grzegorz Wojciechowski, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dwie najważniejsze cechy gospodarstw rodzinnych, które są najczęściej wymieniane, to zbywanie produktów na lokalnym rynku oraz wrażliwość na kontrolę środków produkcji.

Nie został on wprowadzony.

Pan poseł Paweł Rychlik, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Widzę to na przykładzie rolników z powiatów wieluńskiego, pajęczańskiego, wieruszowskiego.

Czy ta nowelizacja ustawy przewiduje możliwość handlu na terenie całego kraju? Dziękuję bardzo. Pani poseł Anna Dąbrowska-Banaszak, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Wysoki Sejmie! Rolniczy handel detaliczny w nowej odsłonie stwarza też nowe oczekiwania.

Dziękuję bardzo. Pani poseł Urszula Nowogórska, Klub Parlamentarny Koalicja Polska. Wydaje się, że jest to dobra ustawa, ale chciałam zadać kilka pytań. Mieszkam na terenie powiatu limanowskiego, w okolicy pięknych powiatów - gorlickiego, sądeckiego i Podhala. Tam w większości przypadków mamy do czynienia z rodzinnymi gospodarstwami, które są bardzo rozdrobnione.

To jest bardzo ważne. To poprawi zdrowie tych, którzy będą z tych produktów korzystać.

Pani poseł Anna Wojciechowska, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Oczywiście popieram wszystkie uwagi moich koleżanek i kolegów z Koalicji Obywatelskiej dotyczące tego projektu. Uważam, że likwidacja limitu jest dobrą inicjatywą, idzie w dobrym kierunku.

Bardzo wielu rolników indywidualnych posiada mnóstwo owoców czy przetworów, które są naprawdę fantastyczne, zdrowe, bez chemii, ale trudno jest znaleźć tych producentów. Czasami nawet nie wiemy, że coś takiego istnieje.

Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! Wysoki Sejmie!

Mam pytanie do pana ministra.

Pani poseł Teresa Pamuła, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Bardzo się cieszę, że ta ustawa jest poprawiona. To bardzo wzmocni rolników na rynku, który mocno się rozwija. Na Podkarpaciu prawie 80% to są małe i średnie gospodarstwa.

To są małe mleczarnie, to są małe serowarnie, to są małe piekarnie. Była taka niemoc, że nie można zrobić tego czy tamtego. Dopiero w 2017 r. mogliśmy wprowadzić rolniczy handel detaliczny, teraz go rozwijamy. Widzimy, że na małych rynkach, na różnych festynach są produkty przygotowane przez rolniczy handel detaliczny. Panie Ministrze! Czy możemy jeszcze liczyć na wsparcie tego rolniczego handlu detalicznego, żeby rolnicy mogli przygotować miejsca do produkcji zdrowej, świeżej i wspaniałej żywności dla Polaków? Dziękuję serdecznie. Odpowiedzi na pytanie, czy możemy jeszcze liczyć na wsparcie, udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan minister Szymon Giżyński. Zapraszam, panie ministrze, uprzejmie.

Dziękuję, szanowni państwo, za te wszystkie szczegółowe uwagi, pytania, ale także za oceny gremialne, bo i takich nie brakowało. Wszystkie są w jakimś sensie równo cenne, bo nawet te, które są niesprawiedliwe i postawione w sposób niemający wiele wspólnego z materią sprawy, też potwierdzają słuszność naszych zamierzeń, może w najwyższym stopniu. Te pytania i wątpliwości pojawiały się zarówno w wystąpieniach klubowych, jak i potem w serii pytań. Jednocześnie gwarantuję, że to, co będzie konieczne, oczywiście niezwłocznie uzupełnimy w formie odpowiedzi pisemnych.

Oczywiście krytykował i sam przesądzał, że ten związek jest uzurpacyjny, chodzi o rolniczy handel detaliczny i Polski Ład.

I to jest najzupełniej jasna i wystarczająca w tym przypadku odpowiedź. To akurat był być może wyjątek, te złośliwości pana posła Plocke, były nam tutaj zafundowane w nadmiarze, nawet jak na nasze przecież niewyszukane sejmowe w tym wypadku czy nie nadmierne wątpliwości, że muszę pozostawić pana posła z nimi sam na sam.

Taka troska, wątpliwość, uwaga, przytyk, że to jest mała skala, że rolnicy na to nie reagują tak, jak powinni, że te zachęty są niewystarczające i że coś nie jest tak.

Taką oczywistość, jeżeli chodzi o zamiary propagandowe, pewną oczywistość w tym względzie.

Na to trzeba czasu, cierpliwości i wiarygodności, i tę wiarygodność zapewniamy, skoro poprawiamy tak ważną ustawę.

Ale, szanowni państwo, te wzorce zachodnie, wzorce innych państw Unii Europejskiej i spoza niej pchają rolników w ramiona spółdzielczości, w ramiona innych form gospodarowania i różnie z tym wychodzi. Więc tutaj bądźmy cierpliwi i konsekwentni. A do pewnych szans, które się tutaj pojawiają, jeszcze za chwilę wrócę. Krótko odpowiem panu posłowi Mirosławowi Maliszewskiemu.

Teraz jest już znacznie, znacznie więcej i trzeba powiedzieć, że jeżeli ta tendencja się utrzyma, jeżeli te przedsięwzięcia, te gospodarstwa będą dochodowe i trwałe, to, proszę państwa, będzie to w moim odczuciu i w naszych zamiarach być może najistotniejsza strukturalna zmiana w naszym rolnictwie, bo ma to bezpośredni związek z bezpieczeństwem żywnościowym Polski.

To jest kwestia przyszłościowa polskiego bezpieczeństwa żywnościowego.

Nie mówimy tutaj, szanowni państwo, w kategoriach mistycznych, w kategoriach literackich, legendarnych, tylko mówimy w kategoriach bardzo realistycznego, bardzo przyszłościowego projektu, o którego powodzenie musimy wszyscy razem zabiegać, a także ta dyskusja i państwa deklaracje, myślę, są gwarancją tego, że będziemy dbać o RHD. Myślę, że jeszcze w niejednej inicjatywie ustawowej i w codziennej praktyce nieraz będziemy czynić to razem.

Mam je oczywiście ułożone w takim porządku, w jakim państwo zabierali głos. Już w serii pytań wystąpił również pan poseł Suchoń. Do jego pytania dołączam informację o ustawie o handlu w niedziele, która rozszerza możliwości działania RHD.

Pan poseł Piotr Borys również nie jest zwolennikiem małej skali czy też w nią nie wierzy. Szukajmy razem rozwiązań, a to, co powiedziałem w takiej wypowiedzi programowej, jest również odpowiedzią na wątpliwości pana posła Piotra Borysa.

Przecież nic z tych rzeczy. Jest tutaj pewna sytuacja, gdzie musieliśmy bardzo jasno odpowiedzieć na pewne żądania, wymagania Unii Europejskiej.

Nic więcej, nic ponad to. Istota ta sama, w istocie się nic nie zmienia, tylko obroniliśmy się tutaj pewną układnością semantyczną, czyli dostosowaniem naszego rozwiązania prawnego do języka wymaganego w Unii. Natomiast to, co do tej pory było, całkowicie pozostaje. Kontrola będzie nie prewencyjna, lecz tylko interwencyjna, kontrola przez nadzór, kontrola rzadka. Myślę, że to państwa powinno uspokoić, bo ta skala stosowania RHD jest już na tyle szeroka i jej powodzenie jest pod pewną kontrolą osądu społecznego, osądu samych rolników, że jasno widać, jak te kontrole funkcjonują.

więc chcę jasno zapewnić: Nic tutaj się nie zmieni. Jeżeli było dobrze i były tu kontrole pożyteczne, racjonalne, sensowne i w swoich wymiarach skuteczne, nic się tutaj pod tym względem nie zmieni.

Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, zawarty w druku nr 1516, do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 30. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1515) Proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych pana Macieja Małeckiego o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Zapraszam pana ministra. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić państwu projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. To największa od 20 lat reforma Kodeksu spółek handlowych, przygotowana przez działającą przy Ministerstwie Aktywów Państwowych Komisję ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego. Te prace były prowadzone przy szerokich konsultacjach i wielu dyskusjach. Pragnąc zachęcić państwa do wspólnej pracy nad przekształceniem tego projektu w część polskiego porządku prawnego, chciałbym przybliżyć powody, dla których ten projekt reformy Kodeksu spółek handlowych powstał. Przedstawię również sylwetki osób, które były zaangażowane w jego przygotowanie. Opowiem o szerokich konsultacjach, jakie towarzyszyły przygotowaniu projektu, który jest przedmiotem naszych dzisiejszych obrad. Przybliżę też państwu najważniejsze instrumenty, które znalazły się w projekcie. Zacznijmy jednak od tego, dlaczego Ministerstwo Aktywów Państwowych rozpoczęło prace nad kodeksem. Jest to bezpośredni efekt rozmów z przedsiębiorcami i sygnałów, że oczekują zmian. Zatem projekt, który przedstawiam, jest przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez polski biznes. Ale potrzeba zmian wynika również z sukcesu naszej gospodarki, tego, w jak dużym stopniu nasza gospodarka rozwinęła się w ciągu ostatnich lat. W miejsce 205 tys. spółek, które funkcjonowały w roku 2000, dziś mamy 460 tys. spółek, a podmioty, które w 2000 r. dopiero stawiały pierwsze kroki w biznesie, dziś niekiedy zarządzają dziesiątkami spółek zależnych i obracają miliardami złotych. Bardziej złożona gospodarka wymaga prawa dostosowanego do swoich potrzeb. Zresztą ten rozwój polskiej gospodarki, polskich spółek wciąż postępuje, z czego, mam nadzieję, jest dumna cała Wysoka Izba. Nasze państwo konkuruje też z innymi krajami coraz odważniej i dynamiczniej, więc potrzebuje do tego właściwych narzędzi. Dobre prawo gospodarcze jest sposobem, by Polska jak najczęściej tę rywalizację wygrywała. Takie warunki stwarza ten projekt, daje zaawansowane narzędzia do dobrej, konkurencyjnej walki na bardzo wymagających zagranicznych rynkach. Co istotne, konsekwencją wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej jest to, że nasze państwo konkuruje z innymi krajami jako miejsce lokowania działalności gospodarczej. Żeby Kodeks spółek handlowych spełnił postawione przed nim wymagania, zaprosiliśmy do współpracy uznanych ekspertów z dużym zakresem wiedzy praktycznej. Zespołami, które przygotowały projekt, jaki dziś przedkładamy Wysokiej Izbie, kierowali: prof. Andrzej Szumański z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który jest jednym z trzech autorów Kodeksu spółek handlowych, dr Radosław Kwaśnicki, uznany ekspert z obszaru ładu korporacyjnego, oraz prof. Piotr Pinior z Uniwersytetu Śląskiego, również czołowy ekspert z zakresu prawa handlowego. Chcę podkreślić też bardzo ważną rolę, ogromną pracę wykonaną przy tym projekcie przez obecnego tutaj dyrektora, doktora prawa Filipa Ostrowskiego, [[Oklaski]] kierującego Biurem Reformy Właścicielskiej w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

I wielką zaletą tego projektu jest to, że w jego przygotowywaniu od samego początku uczestniczyli nie tylko naukowcy, ale też przedsiębiorcy. Nie mamy tu więc do czynienia z projektem, który został tylko skonsultowany z biznesem, ale mamy do czynienia z takim projektem, którego biznes jest współautorem. Do przedstawienia stanowisk zaprosiliśmy ponad 200 podmiotów. Wydłużyliśmy do 45 dni czas konsultacji. Otrzymaliśmy ponad 800 stron uwag i te uwagi w wielu wypadkach uwzględniliśmy w projekcie, który dzisiaj przedkładamy Wysokiej Izbie. Przez pierwszą część prac nad projektem, także tych organizacyjnych, w Ministerstwie Aktywów Państwowych odpowiadał za ten obszar pan minister Janusz Kowalski, [[Oklaski]] któremu dzisiaj bardzo dziękuję z tego miejsca. Na czele Komisji ds. Reformy Właścicielskiej stoi wicepremier, minister aktywów pan Jacek Sasin. Flagową częścią projektu jest regulacja grup spółek, która ma dać spółkom dominującym możliwość efektywnego zarządzania spółkami zależnymi przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów innych uczestników życia gospodarczego. Obecnie obowiązujące przepisy art. 7 Kodeksu spółek handlowych nie spełniają żadnego z tych celów. Niekiedy w doktrynie można spotkać się z poglądem, że problemy w tym zakresie rozwiąże sądownictwo, ale polski system prawny nie należy do systemów krajów prawa zwyczajowego. Odpowiedzialność za stanowienie prawa i mandat społeczny do tego, by to robić, należą właśnie do Wysokiej Izby. Po wejściu w życie nowych przepisów spółki dominujące uzyskają prawo wydawania spółkom zależnym wiążących poleceń. Otrzymają możliwość uzyskiwania ze spółek zależnych informacji na szczególnych zasadach. Uzyskają również możliwość wykupu wspólników mniejszościowych. Z dodatkowymi uprawnieniami spółki dominującej koresponduje jej dodatkowa odpowiedzialność wobec wierzycieli i wspólników mniejszościowych. Interesy tych dwóch grup zostały zabezpieczone formalizmem, jaki ma towarzyszyć wydawaniu poleceń wiążących. Odpowiednikiem przysługującego spółce dominującej prawa wykupu jest natomiast przyznane wspólnikom mniejszościowym prawo odkupu. Rozwiązania z zakresu poprawy efektywności rady nadzorczej to jest odpowiedź na sygnalizowane problemy, że wielokrotnie po tym, gdy w jakiejś spółce dochodziło do nieprawidłowości, pojawiały się później problemy. Gdzie była rada nadzorcza? Dlatego proponowane zmiany dotykają kwestii fundamentalnych dla ładu korporacyjnego, tego, jak zadbać o to, by rada nadzorcza miała informację o tym, co się dzieje w spółce i żeby była w stanie tę informację przetworzyć. Po wejściu proponowanych przez nas przepisów w życie tak właśnie będzie. W pozostałym zakresie w projekcie znalazły się przepisy doprecyzowujące fundamentalne obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych: obowiązek zachowania tajemnicy, obowiązek lojalności. Znalazła się także skodyfikowana już w wielu państwach europejskich zasada biznesowej oceny sytuacji. Jeden z ojców polskiego prawa handlowego Aleksander Doliński pisał: Prawnik daje tylko formę, treści dostarcza nam ekonomista. Tak właśnie w nawiązaniu do najlepszych tradycji polskiego prawa gospodarczego powstawał ten ambitny projekt. Treści dostarczył biznes. Wybitni prawnicy dali formę. I teraz pozostaje nam tylko zwrócić się do Wysokiej Izby o rzeczową i merytoryczną pracę nad tym projektem. Tradycja legislacji w obszarze prawa handlowego polega na tym, że nawet tam, gdzie ludzi dzieliły różnice polityczne, a te dzielą nas także dzisiaj, można współtworzyć dobre prawo dla polskiej gospodarki, bo przecież różnice dzieliły autorów kodeksu handlowego z 1934 r. i dzieliły tę Wysoką Izbę, która w 2000 r. uchwalała Kodeks spółek handlowych. Ale w obu przypadkach udało się wspólnie pracować ponad podziałami w celu jakże ważnym i nakierowanym ku pożytkowi publicznemu. Do takiej właśnie współpracy zachęcam i zapraszam koleżanki i kolegów z Wysokiej Izby. Dziękuję serdecznie. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Bardzo proszę pana posła Janusza Kowalskiego, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny Panie Ministrze! Mam wielki zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość odnośnie do przedłożonego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych i innych ustaw. Oczywiście jest to stanowisko pozytywne i wnioskujemy o przesłanie projektu do dalszych prac. Komisja ta, ponad 60 jej ekspertów, przygotowała ten projekt ustawy, przerywając kilkunastoletni spór na temat prawa holdingowego, prawa koncernowego, ponieważ rzeczywiście można powiedzieć i trzeba powiedzieć, że to jest największa reforma Kodeksu spółek handlowych od 20 lat, ponieważ ten dział IV, który proponujemy, Prawo grup spółek jest fundamentalną nowością w polskim porządku prawnym. Innymi słowy, odpowiadamy na potrzeby polskiego biznesu, szczególnie tego, który chce się rozwijać za granicą, który chce realizować transformację energetyczną, który chce realizować ekspansję i zarządzać w ramach realizacji interesu spółek grupami spółek w sposób absolutnie profesjonalny. Odpowiadamy takim kompromisowym rozwiązaniem - kompromisowym, dlatego że wysłuchaliśmy i biznesu, i praktyków.

Pierwszy, tak jak powiedziałem, to oczywiście prawo grup spółek.

Takie rozwiązania funkcjonują m.in. w Niemczech, na Słowenii, w Czechach czy w Portugalii. Jestem w stanie bronić poglądu, że jeżeli Wysoka Izba zaakceptuje to rozwiązanie, będzie to najnowocześniejsze prawo holdingowe w Europie, ponieważ patrzyliśmy również na błędy popełnione w innych państwach i staraliśmy się wyciągnąć z nich wnioski. Likwidujemy asymetrię informacyjną między zarządem a radą nadzorczą. Rada nadzorcza zgodnie z tym projektem stanie się realnym partnerem w zarządzaniu czy w kontroli nad spółką. Mieliśmy niedawno do czynienia z dyskusją dotyczącą tego, gdzie była rada nadzorcza spółki GetBack, której członkowie mówili, że o niczym nie wiedzieli, mówili: O niczym nie wiedzieliśmy, ponieważ zarząd nie informował o sytuacji spółki. Ten projekt jest właśnie odpowiedzią m.in. na takie sprawy, jak sprawa spółki GetBack. W końcu rada nadzorcza będzie mogła badać potencjalne nieprawidłowości czy dokonywać procesów rekrutacyjnych już poza decyzjami zarządu, będzie miała możliwość zatrudnienia doradcy rady nadzorczej. Taka formuła funkcjonuje w innych państwach. Przerywamy ją. Prawo musi być jasne, dlatego proponujemy określone rozwiązania, które w sposób bezsprzeczny przerwą tę kilkunastoletnią dyskusję. Najważniejsze, że doprecyzowujemy zasady dla członków rad nadzorczych i zarządów w kontekście lojalności, w kontekście poufności, w kontekście dbałości o interesy spółki również po wygaśnięciu kadencji. Szanowni Państwo!

Szukajmy najlepszych rozwiązań dla polskiego biznesu.

W czasie pandemii (Dzwonek) odblokowaliśmy zasadę działania spółek, ponieważ zdecydowaliśmy o elektronicznym podejmowaniu decyzji przez organy nadzorcze i przez zarządy. Druga kwestia dotyczy restrukturyzacji i upadłości; uratowaliśmy wiele polskich firm. Zachęcam państwa do merytorycznej dyskusji. Pani poseł Barbara Dolniak, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kodeks powinna cechować stabilność. Jego zmiana powinna następować tak rzadko, jak to możliwe. Decyzja o zmianie musi wynikać z potrzeby obrotu prawnego. Każda zmiana ma bowiem swoich adresatów. Pytanie brzmi: Czy są to beneficjenci zmiany, czy jej ofiary? O beneficjentach piszą w ramach ukazywania nepotyzmu w spółkach Skarbu Państwa Onet, Wyborcza i Radio ZET. Zmiany w prawie nie mogą być podyktowane interesami politycznymi. Takie działania zmierzają bowiem do zaburzenia systemu prawa oraz stanowią fundament wielu wykroczeń przeciwko literze prawa. Pan minister Małecki wyjaśnia, że otrzyma narzędzie, które pozwoli łatwiej zarządzać grupami spółek. Twierdzi, że proponowane rozwiązania skrócą czas podejmowania decyzji, bo właściciel spółki będzie mógł przez jej organy doprowadzić do podjęcia oczekiwanej decyzji. Zapytany o konkret, odpowiada, że dzięki nowemu prawu holdingowemu spółki odzieżowe dotknięte lockdownem uzyskają możliwość sprawnego przejścia od handlu tradycyjnego do internetowego, a także wdrożenia wspólnych zakupów. Jednak przez ostatnie 30 lat biznes wypracował rozwiązania znane pn. kodeks grupy w ramach istniejącego Kodeksu spółek handlowych, a orzecznictwo zaakceptowało te rozwiązania. Teraz to wszystko wyrzuca się do kosza. Kolejna zmiana to wzmocnienie nadzoru w spółkach kapitałowych. Minister przekonuje, że dzięki wprowadzonej zmianie zarządy w końcu będą obowiązane informować rady nadzorcze o sytuacji spółek, a rada nadzorcza uzyska uprawnienie do żądania od zarządu i pracowników informacji na temat tego, co dzieje się w spółce. Co więcej, minister podkreśla, że członkowie rad nadzorczych będą mogli korzystać z usług niezależnych doradców odpowiedzialnych przed radą nadzorczą. Jak te rozwiązania mają się do struktury spółek kapitałowych w Polsce, gdzie blisko 90 spółek z o.o. to spółki jednoosobowe, ok. 360 tys., a tylko ok. 800 spółek akcyjnych ma masowy akcjonariat, z czego ok. 70 ma wiodącego akcjonariusza? Jaki będzie koszt takiej zmiany dla codziennego funkcjonowania spółek, w tym tych najmniejszych? Uzasadnienie projektu milczy o tym. Co jest rzeczywistym celem tych zmian, skoro merytorycznie nie ma uzasadnienia dla takich zmian? Projekt legalizuje zjawisko instrumentalnego wykorzystywania spółek Skarbu Państwa w celach politycznych i fiskalnych. Prawo holdingowe ma to ułatwić, zadekretować, skoro projekt wskazuje, że spółka ma swój własny interes, niezależny od interesu udziałowców. Wiążące wydawanie poleceń spółkom zależnym przez zarząd spółki matki ma ułatwić zadekretowanie nepotyzmu. Niestety nie będzie jak w powiedzeniu: przykład idzie z góry. W tej sytuacji to rozkaz idzie z góry. Z kolei prawo odmowy wykonania tych poleceń ma zabezpieczać interesy poszczególnych frakcji. Co do rzekomego wzmocnienia rad nadzorczych, w istocie chodzi o rozmycie odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych z nadania politycznego poszczególnych frakcji. Celem jest, by nie można było ustalić osoby odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji o traktowaniu spółek z udziałem Skarbu Państwa jak świnek-skarbonek. Zmiany, które mają rzekomo wzmocnić nadzór nad spółkami, wprowadza wicepremier Sasin. Zbiega się to w czasie z publikacją wyników śledztwa dziennikarskiego o porażającej skali korupcji personalnej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. To jak wpuścić lisa do kurnika, aby strzegł kury przed lisem. Nie damy się nabrać. Intencje są znane, boicie się odpowiedzialności karnej za nepotyzm i szykujecie zmiany w Kodeksie spółek handlowych, aby przemycić legalizację nepotyzmu. Projekt ignoruje strukturę właścicielską spółek kapitałowych w Polsce, dorobek polskiego i zagranicznego orzecznictwa oraz doktryny, a także zasadę ekonomicznej analizy prawa i techniki prawodawczej nakazującą wykazanie, że korzyści ze zmian będą istotnie wyższe od kosztów ich wprowadzenia. Te zarzuty można mnożyć, co wskazuje, że projekt tej treści nie powinien być w ogóle procedowany. Dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo. Proszę, panie pośle, bardzo uprzejmie. Dziękuję. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu klubu Lewicy przedstawić stanowisko dotyczące projektu ustawy, który rzeczywiście jest istotny z punktu widzenia funkcjonowania spółek, grup kapitałowych i wprowadza kilka dobrych rozwiązań. Rzeczywiście zmieniają się realia gospodarcze. Od 20 lat Kodeks spółek handlowych nie był modyfikowany. Ale zwracamy uwagę na jedną rzecz, że ta modyfikacja musi służyć wszystkim.

Kadra zarządzająca w każdej spółce jest najistotniejszym elementem, jeżeli chodzi o uczciwość biznesową i rozwój tychże spółek. Pewnie ta zmiana Kodeksu spółek handlowych to jest odpowiedź na konflikty, które są dzisiaj w spółkach Skarbu Państwa, bo jeden prezes chce wyrzucić wiceprezesa, drugi prezes chce wyrzucić prezesa spółki zależnej, więc trzeba komuś dać do jednej ręki władzę. To mniej więcej w tę stronę idzie. Co do samej intencji wprowadzenia prawa holdingowego rzeczywiście to trzeba uporządkować.

Czy wyobrażacie sobie taką sytuację, że oto prezes Orlenu będzie ustnie wydawał polecenia wiążące prezesowi swojej spółki zależnej?

Mówicie o kwestii dostępu do informacji.

Te kompetencje są absolutnie niejasne, nieostre, w związku z czym to niewątpliwie powinno ulec zmianie. Rzecz druga to jest kwestia dostępu do informacji.

Kolejna rzecz to jest też wprowadzanie, myślę, dużego konfliktu. Mianowicie to jest kwestia wyboru doradców przez rady nadzorcze, poza zarządem. Będzie to polegało na tym, że rada nadzorcza, która akurat, bo tak się dzieje w spółkach Skarbu Państwa, będzie chciała wymienić jednego prezesa kolesia na innego prezesa kolesia, będzie zamawiać opinie prawne poza zarządem - nie wiadomo, za jaką cenę, w jakiej wysokości - żeby udowodnić, że ten zarząd źle funkcjonuje. Tak nie powinno się to dziać, bo to niestety jest zaburzenie porządku gospodarczego i finansowego w każdej z tych spółek. Wprowadzacie jakieś komitety rady nadzorczej.

A więc generalnie tych uwag jest naprawdę bardzo dużo, łącznie z tym, jak te rady nadzorcze są zwoływane - niestety dajecie możliwość taką, żeby bez udziału 100% (Dzwonek) członków rady nadzorczej zmieniać porządek obrad i podejmować inne decyzje. A więc my stoimy na stanowisku takim - sprawa jest bardzo poważna, zobaczymy, czy rzeczywiście intencje wasze są takie, żeby uporządkować sytuację, jeżeli chodzi o holdingi, w Kodeksie spółek handlowych. Będziemy składali poprawki, które będą te wszystkie nieścisłości wyjaśniały, i od tego uzależniamy nasze ostateczne stanowisko. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Mieczysław Kasprzak, Koalicja Polska. Zapraszam. Panie Marszałku!

Natomiast w projekcie jest szereg niejasnych, nieprecyzyjnych zapisów. Naprawdę one budzą wątpliwości tych, którzy wgłębiają się w materię tego projektu.

Tak jak tutaj poprzednik powiedział, ten projekt wymaga wielu zmian - zmian, które spowodują, że będzie to projekt jasny i czytelny. Mamy przykre doświadczenia z zarządzaniem spółkami Skarbu Państwa - właśnie Skarbu Państwa.

To potęguje jeszcze bardziej nasze obawy.

Znamy sprawy niewyjaśnione do tej pory. I to jest bardzo zastanawiające. Bo dyskutujemy o tym w tej chwili i to te próby zdejmowania odpowiedzialności za lekkomyślne wydatkowanie środków finansowych, narażanie na straty Polaków, obywateli polskich spowodowały to, że trudno mieć zaufanie do tych, którzy proponują takie rozwiązania. Pan minister powiedział, że akurat prawo gospodarcze w tej chwili mamy bardzo dobre, że ono się rozwija.

Nie będziemy popierać wniosku o odrzucenie, natomiast oczekujemy, że szereg spraw będzie wyjaśnionych.

Szereg niejasności zostało zgłoszonych również przez zainteresowane strony. Trzeba pracować. Trzeba szukać dobrych rozwiązań, ale to nie może służyć, jak ktoś z przedmówców już powiedział, sprawom politycznym. Zmieni się opcja rządząca, zmienią się politycy, a gospodarka musi się rozwijać, gospodarka musi zachować ciągłość. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Krzysztof Bosak, koło Konfederacji.

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Dobrze, że wreszcie po 20 latach Sejm zajął się nowelizacją prawa regulującego podstawy życia gospodarczego, czyli Kodeksem spółek handlowych. Ta ustawa zasługiwałaby na radykalne uproszczenie, na co zwracają uwagę przedsiębiorcy.

To jest głos ze środowiska przedsiębiorców, który dotarł do nas, do Konfederacji. Niemniej jednak jest kilka zmian, które warto dostrzec i które sprawiają, że te przepisy, które znamy jeszcze z lat 90., być może zaczną nadążać za rozwojem życia gospodarczego, które bardzo poszło do przodu. Pierwsza zmiana, chyba najbardziej probiznesowa, to ograniczenie tej zasady, że można kogoś sądzić i skazywać za działanie na szkodę własnej spółki. Wiemy, że wielokrotnie wobec przedsiębiorców ta zasada była nadużywana. Wiemy, że granica pomiędzy okradaniem własnej spółki a działaniem poprzez podejmowanie ryzyka gospodarczego i poniesieniem strat niekiedy w realiach życia gospodarczego bywa płynna i jest kwestią oceny. Te sprawy ostatecznie oceniane są przed sądem. Wprowadzenie do prawa zasady biznesowej oceny sytuacji polegającej na tym, że sąd, widzi, iż straty zostały poniesione przez spółkę, jest to bezsporne, natomiast wie też, że wynikało to z podjęcia ryzyka gospodarczego, a nie z próby wyprowadzenia pieniędzy z tej spółki.

Kolejna rzecz, która wydaje się rozsądna, to zakaz sprawowania funkcji we władzach spółek przez osoby skazane za łapownictwo, płatną protekcję, nie mówiąc już o nadużywaniu uprawnień funkcjonariusza publicznego. To, co też wydaje się ciekawe, to sytuacja wzmocnienia pozycji mniejszościowych akcjonariuszy poprzez sprawienie, że rady nadzorcze zostaną wzmocnione.

Jeżeli ktoś twierdzi, że w tej chwili w obecnym stanie prawnym jest to wyłącznie kwestia kompetencji, to znaczy, że niestety nie do końca wie, o czym mówi. Wprowadzenie także prawa holdingowego odbieram jako zatwierdzenie pewnego stanu faktycznego, który mamy w tej chwili w gospodarce, gdzie metodami dyskrecjonalnymi zarządza się grupami kapitałowymi poprzez swego rodzaju unie personalne. Natomiast aktualne prawo aktualizuje rzeczywistą sytuację gospodarczą w ramach porządku prawnego. Na minus: sporo niejasności, późne złożenie tego projektu i krótkie vacatio legis. To są jednak daleko idące zmiany. Być może warto rozważyć vacatio legis roczne, a nie zaledwie 6-miesięczne. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050.

Panie Ministrze! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050 w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Szanowni Państwo! Deklarowanym przez rząd celem ustawy jest wprowadzenie regulacji prawnej prawa holdingowego, jak również wyposażenie rad nadzorczych w nowe uprawnienia, a także wyeliminowanie wątpliwości podnoszonych w praktyce gospodarczej. Przeanalizowaliśmy bardzo dokładnie proponowane zmiany, zasięgnęliśmy opinii praktyków, wychodząc z założenia, że po ewentualnym przyjęciu projektowane przepisy mają służyć przede wszystkim gospodarce. Celowo rezygnuję z omawiania poszczególnych aspektów prawnych na rzecz sygnalnego omówienia tych zmian, które widzimy jako zmiany problemowe. Bo to właśnie ze strony rynku pojawia się najwięcej pytań i wątpliwości dotyczących proponowanych zmian. Pierwsza grupa to są zmiany dotyczące prawa holdingowego i trudno nie oprzeć się wrażeniu, co zresztą było już słychać, że będą one dotyczyły głównie spółek Skarbu Państwa.

Te jednak są wyłączone z uwagi na inne regulacje, bardziej restrykcyjne. Wydaje się, że jedyną grupą, dla której te zmiany mogą mieć znaczenie, są spółki Skarbu Państwa, a te zmiany spowodowałyby wzmocnienie politycznego nadzoru. Zresztą symptomatyczne jest to, że autorem nowelizacji jest MAP, a nie np. ministerstwo rozwoju. Warto zauważyć, że mimo zwiększenia tych zapisów o odpowiedzialności finansowej i karnej w praktyce przyjęte uregulowania mogłyby zapewnić bezkarność zarządom spółek w ramach grup firm, a przecież nie o to ma w tym projekcie chodzić. Znowu wracamy do traktowania spółek Skarbu Państwa jako łupu politycznego i stąd problemy decyzyjne, panie ministrze, bo każdy traktuje taką spółkę jak swoją synekurę i jak dojną krowę. Jest na to lekarstwo prostsze niż nowelizacja kodeksu: skończyć z nepotyzmem, skończyć z kolesiostwem. Właśnie teraz Polska 2050 przedstawia założenia do projektu ustawy, który właśnie ma z tym skończyć. Zachęcam do tego, aby skorzystać. Kolejna grupa to zapisy dotyczące rad nadzorczych. Amerykanie mówią, że jeżeli coś nie jest zepsute, to nie warto tego naprawiać. Tymczasem projekt bardzo mocno ingeruje w dotychczasowe uprawnienia rad nadzorczych i niestety skutkiem zmian będzie m.in. możliwość podejmowania zaskakujących decyzji pod nieobecność części członków czy możliwość wykonywania przez członków rady spółki dominującej zadań nadzoru nad spółkami podporządkowanymi. W efekcie trudno tak naprawdę mówić o odpowiedzialności rad nadzorczych spółek podporządkowanych (Dzwonek) i czytelności nadzoru korporacyjnego. W projekcie rezygnuje się także z zasady kolegialności, dając wszystkim członkom prawo do indywidualnego działania bez konieczności delegowania przez radę.

Umożliwia się także radzie zatrudnienie na koszt spółki dodatkowych doradców.

Powiem wprost: to jest kolejna autostrada do wyprowadzenia środków ze spółek Skarbu Państwa. Projekt wprowadza co prawda finansową i karną odpowiedzialność zarządu. za brak właściwej współpracy, ale nie wyjaśnia pomiędzy którą radą. Wspomniałem tylko o części tych problemów. W związku z tym tylko dlatego nie złożę wniosku o odrzucenie, ale oczekujemy bardzo pogłębionej dyskusji nad projektem w komisji. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rzeczywistość gospodarcza Polski ulega ciągłym przeobrażeniom i jak to często bywa, wyprzedza obowiązujące regulacje prawne, które nie sprzyjają zwiększeniu efektywności zarządzania przedsiębiorstwem. Procedowana ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw jako cel zasadniczy stawia wprowadzenie do polskiego prawa regulacji prawnej prawa holdingowego. Proponowane zapisy regulują relacje między spółką dominującą a jej spółkami zależnymi i wyposażają rady nadzorcze w narzędzia pozwalające na bardziej efektywny nadzór korporacyjny. Wprowadzona w 2000 r. regulacja prawa holdingowego uchylająca art. 7 Kodeksu spółek handlowych nie uwzględniła unormowania kwestii prawnych holdingów faktycznych, czyli spółek, między którymi powstał stosunek dominacji i zależności. Nowy dział pt. „Grupa spółek” dotyczy holdingów faktycznych i wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez przedsiębiorców. Środowiska gospodarcze są podzielone na zwolenników i przeciwników przyznania szerokich kompetencji organom spółki dominującej wobec spółek należących do grupy spółek. Utworzenie struktury holdingowej nie oznacza wyłączenia obowiązywania prawa podatkowego, które nakłada sankcje z tytułu transferu zysków, a szczególnie z tytułu naruszenia zasady zawierania umów między spółkami powiązanymi kapitałowo według cen rynkowych na takich samych warunkach jak między podmiotami niezależnymi. Elementem definiującym grupę spółek jest przyjęcie przez spółki uczestniczące w grupie wspólnej strategii gospodarczej, która wskazuje, że spółka dominująca sprawuje jednolite kierownictwo nad spółkami zależnymi. Jest to równoznaczne z przyjęciem kryterium funkcjonalnego. Jako koło Kukiz’15 - Demokracja Bezpośrednia uznajemy proponowane regulacje za potrzebne dla sprawnego zarządzania przedsiębiorstwami. Dlatego opowiadamy się za dalszym procedowaniem i liczymy na szybkie uchwalenie ustawy. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do pytań.

Zapraszam, panie pośle. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Rzeczywiście gospodarka ruszyła trochę do przodu, mamy już kilka lat po wejściu pierwszego kodeksu i kilku ostatnich zmian, ale też trzeba powiedzieć, że nastąpiły również ogromne zmiany w stosunku do obsady zarządów, rad nadzorczych, właśnie te, które obserwujemy dzisiaj w mediach społecznościowych. To partie polityczne nagle zaczęły zawłaszczać te organy. A wy co robicie? W tej ustawie mówicie tak: doradcy rad nadzorczych, dominujące rady nadzorcze, komitety rad nadzorczych. To kolejne synekury dla watażków partyjnych, dla ludzi z legitymacją jednej partii. My chcemy kodeksu, który ma być konstytucją przedsiębiorców, opartego na niezależności partyjnej. A że rzeczywiście macie takich, a nie innych członków rad nadzorczych, słabych, tylko z legitymacją partyjną, nie z kompetencjami, to trzeba ich obudować kolejną armią ludzi. Panie Ministrze!

Panie Ministrze! Chciałem zapytać o dwie sprawy, panie ministrze. Pierwsza rzecz to możliwość wydawania tych poleceń wiążących. Uregulowania powodują, że te polecenia mogą być wydawane w formie ustnej.

Drugie pytanie dotyczy procesu podejmowania decyzji przez rady nadzorcze. Zaproponowali państwo, aby rady nadzorcze mogły dokonywać przewrotów, bo tak należy odczytywać sytuację, w której pod nieobecność członków rady nagle na posiedzeniu pojawia się jakiś dodatkowy punkt i w ramach tego punktu mogą głosować tylko ci (Dzwonek), którzy są obecni.

Panie Marszałku! Już drugi raz się pomyliłem. Mało jest czasu, ale chciałem na początku wyrazić swoje zaskoczenie tym, że tutaj ten proces konsultacji i ukuwania tej ustawy jest negowany.

Bardzo prosiłbym. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Jan Szopiński, Klub Parlamentarny Lewicy. Wysoka Izbo! Po pierwsze, panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję, że określił pan, że nad tą ustawą nadzór sprawował pan minister Sasin. Ustawodawca bardzo precyzyjnie określił procentowy udział własności w ustawie zwanej antykorupcyjnej. W sytuacji występujących dużo częściej i na większą skalę problem ten jest jednak pominięty. Kto i na jakiej podstawie będzie określał, czy spółka jest spółką powiązaną czy zależną? Jaki jest maksymalny pakiet udziałów, który można objąć, aby urząd nie uznał spółki za zależną? Chodzi o propozycję OPZZ, aby udział pracowników w radach nadzorczych powyżej 50 osób był obowiązkowy. Uprzejmie proszę pana ministra o odpowiedzi na piśmie. Dziękuję bardzo. Pan poseł Dariusz Olszewski, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jak państwo wiecie, bliska mojemu sercu jest tematyka sportowa. Nasi przedsiębiorcy, a zwłaszcza czempioni naszej gospodarki, to podmioty, które odgrywają istotną rolę w finansowaniu sportu zawodowego. Za sukcesami naszych sportowych mistrzów takich jak Iga Świątek, Robert Kubica, Anita Włodarczyk czy Maria Andrejczyk stoi oczywiście wielki talent, stoi tytaniczna praca, ale potrzebne jest również zapewnienie im zaplecza finansowego. Zaplecze to zapewniają nierzadko spółki działające z wykorzystaniem grup kapitałowych. Dlatego chciałbym zapytać, czy projektodawca widzi potencjał, by wejście w życie prawa grup spółek przyczyniło się do lepszego, bardziej skoordynowanego finansowania sportu zawodowego czy również sportu amatorskiego w naszym kraju przez spółki działające jako grupy kapitałowe? Dziękuję serdecznie. Pan poseł Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Chodzi wam o to, żeby nie było prawa holdingowego, które odpowiada na najważniejszą rzecz? Bo dzisiaj kancelarie prawnicze łupią m.in. spółki Skarbu Państwa, bo prawo jest niejasne. Czy chodzi wam, Platformo Obywatelska, jednak o to, żeby nie wzmocnić rad nadzorczych, żeby był skuteczny nadzór nad spółkami Skarbu Państwa i nad 440 tys. spółek kapitałowych w Polsce? Jeżeli macie uwagi, zgłoście te uwagi. A dzisiaj stajecie dokładnie przeciw polskiemu biznesowi, który potrzebuje jasnych i czytelnych zasad. To jest nowoczesne prawo gospodarcze prywatne, nie macie żadnych merytorycznych argumentów i chcecie odrzucić projekt ustawy, który jest adresowany przede wszystkim do prywatnego biznesu. Dziękuję serdecznie. Pani poseł Maria Małgorzata Janyska, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Świat fikcji, swojego wąskiego podwórka i świat rzeczywisty. Ten świat rzeczywisty to są właśnie ci prywatni przedsiębiorcy, którzy twierdzą, że nie było należytej zapowiadanej pracy merytorycznej. To są autorytety, eksperci naukowi, ale także praktycy, którzy mówili, że była obietnica przygotowania dobrej pracy merytorycznej w oparciu o konferencje naukowe, także międzynarodowe. Niestety to się nie odbyło. 45 dni na konsultacje, i to jeszcze w okresie wakacyjnym. Czy można to nazwać prawidłowymi konsultacjami? Czy skierowanie wniosków to są konsultacje? Moim zdaniem nie. Pan minister zasłaniał się także dobrym prawem gospodarczym. Tymczasem za rządów Prawa i Sprawiedliwości mamy do czynienia z inflacją prawa na niespotykaną skalę. Jeśli chcemy stanowić dobre prawo gospodarcze (Dzwonek), to powinniśmy zacząć od tego - i to jest nasza propozycja - żeby uchwalić w tej Izbie wreszcie normalne, porządne i dobre zasady stanowienia prawa, które przede wszystkim będą się kierowały oceną skutków w działalności przedsiębiorców.

Pan poseł Andrzej Szewiński, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Tak jak powiedziała moja przedmówczyni, dobre prawo to proste prawo i egzekwowane prawo. A my, posłowie, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby z tej Izby wychodziły po konsultacjach społecznych, po konsultacjach z opozycją dobre ustawy. W przedmiotowym projekcie jest wiele też dobrych zapisów, natomiast diabeł tkwi w szczegółach. Pytanie, czy wprowadzenie nowelizacji ustawy wpłynie na zwiększenie kosztów prowadzenia spółek oraz ograniczenie decyzyjności i niezależności organów spółek podległych, których dotyczy projekt. Dziękuję bardzo. Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Czytając projekt ustawy, należy zacząć od uzasadnienia, bo uzasadnienie powinno przedstawiać, informować, dlaczego i w jakim zakresie jest zmieniane prawo. Tymczasem uzasadnienie już na samym wstępie jest niezgodne ze stanem faktycznym. Bo proszę państwa, czy to jest prawda, że inwestorzy zagraniczni korzystają ze sprzyjających warunków biznesowych w Polsce, czy też wybierają Polskę ze względu na atrakcyjność krajowego systemu prawnego?

Wskaźniki atrakcyjności biznesowej w Polsce się pogarszają, wszystkie wskaźniki światowe to potwierdzają, a PiS dzisiaj twierdzi (Dzwonek), że mamy najlepsze wskaźniki. Dziękuję bardzo. Pan poseł Rafał Adamczyk, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! W ramach konsultacji OPZZ postuluje o wprowadzenie do projektu ustawy przepisów, które zagwarantują udział pracowników w radach nadzorczych i zarządach spółek sektora prywatnego zatrudniających powyżej 50 pracowników. Co ważne, partycypacja we władzach spółek prywatnych powinna uwzględniać obowiązujące uprawnienia pracowników wynikające z ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Bardzo bym prosił o odniesienie się do tego postulatu i pisemną odpowiedź. Dziękuję bardzo. Pan poseł Grzegorz Lorek, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Główna nowelizacja albo, powiedzielibyśmy, kodeks, nad którym pracujemy, to rok 2004. Już dawno temu powinniśmy się tym kodeksem zająć.

Chciałbym powiedzieć, że dzisiaj zarząd spółki mówi radzie nadzorczej tyle, ile chce zarząd. I to umocnienie jest dobrym postulatem.

To jest ciekawy postulat także w przypadku NABE. Dziękuję bardzo. Pani poseł Barbara Dolniak, Koalicja Obywatelska. Dziękuję, panie marszałku.

Jest niejasna definicja grupy spółek i tym samym nie wiadomo, czy ona powstaje automatycznie czy dobrowolnie.

Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jako wieloletni samorządowiec z Podkarpacia, z ziemi sanockiej pragnę podkreślić, że w naszej gospodarce można wyróżnić ze względu na charakterystykę właściciela trzy typy spółek, tj. spółki prywatne, spółki Skarbu Państwa i spółki komunalne. W wypowiedziach dotyczących projektu reformy Kodeksu spółek handlowych zaznacza się, że w toku prac nad ustawą reprezentowane były zarówno spółki prywatne, jak i spółki Skarbu Państwa. Chciałbym zapytać o spółki komunalne, które stanowią przecież ważną część naszej gospodarki. Na ile ich perspektywa i perspektywa jednostek samorządu terytorialnego wybrzmiewała w toku prac i na ile będą one w stanie skorzystać z dobrodziejstw tej największej od 20 lat nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, przygotowanej z inicjatywy i pod koordynacją posła Janusza Kowalskiego? Pani poseł Joanna Jaśkowiak, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pan minister mówił dużo o tworzeniu dobrego prawa, przedstawiając uzasadnienie, z którego jego zdaniem tworzenie dobrego prawa wynika. Ja chciałabym zwrócić uwagę na problem, z którym jako świeżo upieczony, a może już doświadczony, poseł spotykam się tutaj, a mianowicie z kiepskim stanowieniem prawa. Chciałabym zwrócić uwagę, że nowelizacja Kodeksu spółek handlowych jest kolejną, bo jeśli dobrze pamiętam, siódmą nowelizacją tego kodeksu w tym roku. Tych nowelizacji jest bez liku, są nieprzemyślane, niepowiązane. Chciałabym zapytać w związku z tym, nie negując oczywiście konieczności wprowadzania zmian w materii kodeksowej: Kiedy wreszcie poważnie, rzetelnie i bez pośpiechu strona rządząca zabierze się do uporządkowania spraw objętych materią kodeksową? Kiedy zaprzestanie dokonywania zmian ad hoc celem przyjęcia regulacji przewidzianych do rozwiązania doraźnych interesów partii rządzącej? Chciałabym zaapelować tym samym o przywrócenie działania Komisji Kodyfikacyjnej zlikwidowanej w 2015 r. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Jako profesor prawa w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej, doktor habilitowany mam kontakt z naukowcami i praktykami. Cała nowelizacja stanowi zniszczenie Kodeksu spółek handlowych. Projekt prawa handlowego jest sprzeczny z wieloletnią praktyką orzecznictwa polskich sądów, w tym Sądu Najwyższego, jest konfliktogenny dla struktur grup kapitałowych. Jest szkodliwy dla akcjonariuszy mniejszościowych. Ma na celu panowanie rządzących nad grupami kapitałowymi spółek Skarbu Państwa. Zmiany w unormowaniu rady nadzorczej to legislacyjny, logiczny koszmar.

Dziękuję serdecznie. Pan poseł Mariusz Gosek, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Wreszcie po 21 latach powstała największa reforma Kodeksu spółek handlowych. Kłamstwem jest to, co tutaj państwo zarzucacie, że nie było konsultacji. Przede wszystkim przy tej ustawie pracowało 60 ekspertów z różnych stron i różnie można ocenić, 60 wybitnych ekspertów. 20 podmiotów brało udział w tych konsultacjach.

Dziś oni, jeżeli ten procedowany projekt ustawy wejdzie w życie, nie będą już mogli zasiadać w spółkach prawa handlowego i doskonale o tym wiecie, nie będą mogli zasiadać w radach nadzorczych. A do pani poseł jedno zdanie, [[Dzwonek]] bowiem pani poseł wskazała, że rada nie wydaje wiążących poleceń.

Nie ma Tadeusza. Pan poseł Krzysztof Grabczuk, Koalicja Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Temat jest bardzo poważny, ponieważ de facto dotyczy gigantycznych pieniędzy i dotyczy łatwości prowadzenia działalności gospodarczej.

Jest tam wiele niejasnych zapisów, np. rola i pozycja spółki wiodącej, odpowiedzialność rad nadzorczych i członków zarządu. System prawny musi być trwały i stabilny.

To, co jest państwa wielką wadą, państwo za każdym razem rzucacie projekt ustawy. Konsultacje - jeśli myślimy o czymś, żeby coś było trwałego i stabilnego - powinny trwać naprawdę długo, dużo dłużej, po to żebyśmy nie musieli później naprędce poprawiać przepisów prawa. Bardzo proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych pana ministra Macieja Małeckiego.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Patrzę na panią poseł Barbarę Dolniak. Drugi pan poseł już chyba wyszedł z sali, choć zadaje pytania we wszystkich sprawach. Raczej liczę na to, że nieprawda, która padła z ust pani poseł, wynikała z tego, że pani tej ustawy nie przeczytała. Otóż pani poseł powiedziała, zarzuciła pani, że wprowadzamy do ustawy możliwość wydawania poleceń spółce zależnej przez spółkę dominującą nie w formie pisemnej. Spółka dominująca wydaje wiążące polecenie w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności, pani poseł. Co więcej, wskazujemy, określamy katalog wymogów, jakie to polecenie musi spełniać, żeby było wiążące. To jest oczekiwane przez spółkę dominującą zachowanie spółki zależnej w związku z wykonaniem wiążącego polecenia. Polecenie musi zawierać interes grupy spółek, który uzasadnia wykonanie przez spółkę zależną tego polecenia. Musi określać spodziewane korzyści lub szkody spółki zależnej, które będą następstwem wykonania polecenia spółki dominującej, o ile występują. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeśli mowa o przewidywanej szkodzie, to musi być określony sposób i termin naprawienia tej szkody wobec spółki zależnej przez spółkę dominującą w okresie nie dłuższym niż 2 lata. Państwo posłużyliście się nieprawdą. Z tej mównicy padło wiele ogólnych sformułowań, że coś się nie podoba. Informuję, że zmian przepisów art. 21.1 do 21.16 nie stosuje się do Skarbu Państwa.

Przykładowo PKP SA może być spółką dominującą wobec spółek zależnych, z wyłączeniem spółek, które są spółkami publicznymi w tej grupie. W przypadku PKP to akurat PKP Cargo, bo jest notowana na giełdzie od 2013 r. Proszę państwa. Pani poseł, mam prośbę, żeby pani najpierw przeczytała ustawę, bo pani naprawdę. Liczę, że pani powiedziała kłamstwo z tej mównicy, bo pani tego nie przeczytała, i że nie kłamała pani świadomie. Proszę państwa, padł zarzut ze strony opozycji, że będą jakieś dodatkowe ciała w formie komitetów rad nadzorczych. Podstawowa rzecz: rada nadzorcza może tworzyć komitety do pewnych obszarów działalności spółki. To trochę tak, już tłumacząc państwu tak bardzo, bardzo przystępnie, jak Wysoka Izba tworzy komisje.

Odpowiadając na pytanie dziennikarza, w jaki sposób spółki, grupa spółek, spółka dominująca. Podałem przykład z czasów pandemii. Przyjmijmy, że mamy grupę spółek z branży odzieżowej i następuje lockdown. Są zamykane sklepy, galerie handlowe, tak było. W ramach tej grupy spółek jedne spółki radzą sobie lepiej z wejściem do sprzedaży internetowej, inne - gorzej. Jedne sprawniej uzyskują rynek w sieci, inne - nie. Ten przykład, który podawałem, opisywał dokładnie taką sytuację: że w przypadku grupy spółek, spółki dominującej i spółek zależnych, mogą pójść bardzo szybkie decyzje biznesowe. Po co? Po to, żeby ratować te firmy, żeby dawać im lepsze narzędzia do działania na konkurencyjnym rynku. Może chcecie odrzucić ten projekt dlatego, że zaostrzamy przepisy wobec osób skazanych za łapownictwo czynne, bierne, za płatną protekcję. Takie osoby nie będą mogły zasiadać w organach spółek. To jest jeden z zapisów naszego projektu. Wyśmiewaliście to państwo. Na początku liczyłem naprawdę na to, że będziemy merytorycznie rozmawiali, że będą konkretne przykłady, konkretne propozycje zmian. Nadal liczę na to w czasie pracy w komisji, bo wierzę głęboko, że Wysoka Izba nie przyjmie wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Jestem zaskoczony też z takiego powodu, że tych uwag, które dzisiaj państwo wytropiliście, tak jak np. to niby polecenie wydawane wobec spółki zależnej, które nie musi mieć formy pisemnej, eksperci i prawnicy w całej Polsce nie dostrzegali. A państwo to dostrzegacie.

Proszę państwa, my w czasie pandemii otworzyliśmy możliwość zdalnego uczestniczenia, elektronicznego uczestniczenia w posiedzeniu rady nadzorczej, i to nadal obowiązuje. Nawet jeśli ktoś nie pojedzie na posiedzenie rady nadzorczej, ale z telefonu, z którym się dzisiaj nie rozstajemy, z takim posiedzeniem ma łączność, to też może brać w tym udział. Pan poseł Dariusz Olszewski - bardzo dziękuję.

Daje możliwość koordynacji. Daje efekt skali. Liczę, że będzie to korzystne nie tylko dla polskiego sportu, ale także dla polskiej kultury, dla innych działań CSR-owych.

Tak, chcemy wyposażyć rady nadzorcze w możliwość korzystania z doradców po to, żeby rady nadzorcze miały taką możliwość, żeby zaciągały informacje nie tylko od zarządu spółki, ale żeby miały możliwość weryfikowania tych informacji. I to, co dzisiaj wyśmiewacie - być może gdyby w GetBacku rada nadzorcza była obligowana i odpowiadała w sposób realny, jaki chcemy tu wprowadzić, za nadzór nad spółką, i miała możliwość korzystania z doradców, nie doszłoby do tych skandalicznych zaniedbań. Przypomnę, to Prawo i Sprawiedliwość przygotowało ustawę, która wprowadziła transparentność kosztów usług prawnych, konsultingowych, doradczych. Też byliście przeciwni tamtym rozwiązaniom. Szanowni Państwo!

Rozumiem, że państwa jako opozycję może to uwierać, ale będę to powtarzał, bo o tym trzeba pamiętać i o tym trzeba mówić, że PKN Orlen w czasie pandemii, w czasie największego kryzysu po II wojnie światowej osiągnął w 1 rok większy zysk niż za waszych czasów łącznie przez 8 lat.

To kiedy, kiedy.

Polskie Linie Lotnicze LOT w czasie najgorszego roku w historii lotnictwa, roku 2020, osiągnęły większy przychód niż w każdym z wybranych lat rządów Platformy i PSL. Skupmy się na ustawie. Jesteśmy otwarci na argumenty i wierzymy, że także poprawki zgłaszane przez państwa, przez opozycję mogą coś poprawić, mogą wprowadzić korzystne zmiany w projekcie, który przygotowaliśmy, bo na tym polega praca w Wysokiej Izbie, w sali plenarnej i w komisjach, i do takiej pracy państwa jeszcze raz zapraszam mimo tych złośliwości, półprawd i oczywistych nieprawd, które dzisiaj ze strony opozycji padły z tej mównicy. Bardzo dziękuję. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 31. porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1225) Proszę bardzo pana senatora Ryszarda Bobera o przedstawienie uzasadnienia projektu.

Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo! W imieniu Izby wyższej polskiego parlamentu mam przyjemność przedłożyć państwu projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Tak naprawdę dotyczy on zapisów związanych z działalnością komorniczą w ramach windykacji w polskich gospodarstwach. W związku z tym, że rzeczywiście dochodziło w tym obszarze do wielu nieprawidłowości, komornicy działali na podstawie rozporządzenia, które co prawda było rozporządzeniem ministra finansów, ale w uzgodnieniu z ministrem rolnictwa, tym niemniej był to akt niższego rzędu, Senat Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, abyśmy zapisali to w formie ustawy i by nie dochodziło do takich sytuacji, które mają i miały miejsce. Nie mówię, że w 100%, ale w części windykacje doprowadzały do tragedii w rodzinnych gospodarstwach, nie tylko kończących się zaprzestaniem działalności rolniczych, ale również do osobistych tragedii rolników. Chcę zapewnić Wysoką Izbę, że procedowanie nad projektem ustawy w Senacie było bardzo długim procesem, była ogłaszana przerwa po to, żeby doprecyzować pewne zapisy, żeby skonsultować je z różnymi organizacjami, które wniosły uwagi do przedłożonego projektu ustawy.

Wnoszę tutaj i proszę Wysoką Izbę, abyśmy ten artykuł, który mówi, że w momencie, kiedy windykacja dotyczy wszystkich składników gospodarstwa, ma ona pierwszeństwo przed wszystkimi pozostałymi punktami, które odnoszą się do poszczególnych składników, rzeczywiście nie był procedowany, panie ministrze, żebyśmy przyjęli.

Jeszcze raz dziękuję Wysokiej Izbie i panu marszałkowi za szybkie procedowanie nad tak ważną ustawą i proszę Wysoką Izbę o przyjęcie w przedłożeniu senackim projektu ustawy - Kodeks postepowania cywilnego. Dziękuję. Jeśli pan senator zechce zostać podczas procedowania nad tym punktem, to później będzie możliwość odniesienia się do wystąpień oraz do pytań. Dziękuję bardzo panu senatorowi. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Grzegorz Lorek, który przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Senatorze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić opinię w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, druk nr 1225. Projekt ustawy przewiduje przeniesienie rozwiązań zawartych w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Przedmiotowy projekt jest zainspirowany postulatem zawartym w indywidualnej petycji wniesionej do Senatu, w której zwrócono uwagę m.in. na okoliczność, że w świetle wymogów konstytucyjnych wszelkie wyłączenia spod egzekucji dotyczące zwierząt i rzeczy ruchomych potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego muszą być uregulowane na poziomie ustawowym. Obecnie natomiast na poziomie aktu wykonawczego uregulowane są kwestie, które rzutują zarówno na prawo do sądów - w tym jego aspekcie, który wiąże się z gwarancją wykonywania prawomocnego orzeczenia - jak i na ochronę praw majątkowych wierzyciela, który decyduje się na wszczęcie egzekucji sądowej przeciwko rolnikowi prowadzącemu gospodarstwo rolne. Ponadto część postanowień rozporządzenia z dnia 5 lipca 2017 r. wykracza poza delegację z art. 830 Kodeksu postępowania cywilnego.

Celem jest także zwiększenie koherentności systemu prawa, albowiem w przypadku postępowania egzekucyjnego w administracji ustawodawca już na poziomie ustawowym określił te zwierzęta i rzeczy ruchome, które są wyłączone spod egzekucji w razie skierowania jej przeciwko rolnikowi prowadzącemu gospodarstwo rolne. Pozytywnie należy ocenić koncepcję ustawowego uregulowania zagadnień przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, jak też zasad postępowania w tej materii przez właściwe organy. Bez wątpienia przyczyni się to do zwiększenia ochrony prawnej dłużników będących rolnikami.

W konkluzji należy stwierdzić, że przyjęcie projektu w jego aktualnym kształcie skutkować będzie obniżeniem zdolności kredytowej rolników. Wadą dotychczasowego § 5 rozporządzenia jest konieczność równoczesnego kierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości, w sytuacji gdy egzekucja z jednej nieruchomości pozwalałaby na zaspokojenie wierzyciela. Tym samym należałoby zmierzać w kierunku poszerzenia możliwości prowadzenia egzekucji z nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego w sytuacji, gdy wierzyciel dysponuje hipoteką ustanowioną na jego rzecz przez samego dłużnika, względnie gdy tylko egzekucja z nieruchomości pozwoli na zaspokojenie wierzyciela.

Rozwiązania takie pozwoliłyby na zrównoważenie interesu wierzycieli i dłużników bez jednoczesnego stwarzania ryzyka dla rolników indywidualnych korzystających z pożyczek lub kredytów bankowych. Wysoka Izbo! Z uwzględnieniem przedstawionych zastrzeżeń klub Prawo i Sprawiedliwość pozytywnie opiniuje przedłożony projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, druk nr 1225, i wnosi o dalsze prace nad nim. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu posłowi. Teraz proszę panią poseł Joannę Jaśkowiak o przedstawienie stanowiska Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Panie Senatorze! Chciałabym przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska dotyczące senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, zawartego w druku nr 1225.

Zdaniem wnoszącego określenie zwierząt i przedmiotów należących do rolnika, który prowadzi gospodarstwo, a które nie podlegają egzekucji, stanowi materię ustawową. Do tej pory problematyka wyłączenia spod egzekucji określonych rzeczy była normowana przepisami rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Należy zgodzić się z poglądem, że w świetle wymogów konstytucyjnych wszelkie wyłączenia spod egzekucji, zarówno dotyczące zwierząt, jak i rzeczy ruchomych potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego, muszą zostać uregulowane na poziomie ustawowym. Nie ulega zatem wątpliwości, że rozporządzenie jest aktem normatywnym niższego rzędu, który może służyć jedynie wykonaniu ustawy, a nie może jej zastępować, uzupełniać, czy nie może modyfikować przyjętych rozwiązań. Dlatego w następstwie przyjęcia projektowanej zmiany regulacje dotyczące zwierząt i przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, które nie podlegają egzekucji, uzyskają walor konstytucyjności. Treść proponowanych zmian niemal wiernie odzwierciedla postanowienia wynikające z cytowanego rozporządzenia ministra sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o korekty, dotyczą one raczej zmian redakcyjnych lub dotyczących konieczności dostosowania odesłań czy terminologii. Ten projekt zakłada również uchylenie dotychczasowego art. 830 Kodeksu postępowania cywilnego ze względu na to, że wszystkie uregulowania zostaną unormowane w ustawie - te, które były unormowane w rozporządzeniu - i stanie się on po prostu zbędny. Ważne jest również wprowadzenie przepisów intertemporalnych, gdyż do spraw wszczętych pod rządami poprzednich przepisów będą stosowane dotychczasowe przepisy.

Bardzo dziękuję, pani poseł. Proszę teraz pana posła Romualda Ajchlera o przedstawienie stanowiska klubu parlamentarnego Lewica. Wysoka Izbo! W imieniu klubu Lewicy przedkładam stanowisko w sprawie uchwały Senatu o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Nowelizacja przedstawiona przez Senat jest stosunkowo nieobszerna, ale jest bardzo istotna z punktu widzenia rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, kiedy to z różnych powodów stał się dłużnikiem.

Dotyczy to takich gatunków zwierząt jak bydło mleczne, mięsne, konie, świnie, owce, drób, zwierzęta futerkowe i inne, łącznie z narzędziami potrzebnymi do prawidłowego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wysoka Izbo!

Nie było tu żadnej złośliwości ze strony rolnika, tylko zwykła niemożliwość spłaty zobowiązań, które przed nim stały. Wysoka Izbo! Przykład z Wielkopolski, niedaleko mojego biura poselskiego. Rolnik wziął kredyt na zakup maszyn rolniczych.

Tych wszystkich spraw możemy uniknąć, szybko debatując nad projektem ustawy. Dziękuję bardzo panu posłowi. Na sali obecny jest współautor tego projektu ustawy pan senator Bober, który z pewnością odniesie się do wszystkich zagadnień. A teraz pan poseł Zbigniew Ziejewski przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panie Senatorze! Mam przyjemność i zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, druk nr 1225. Procedowany projekt dotyczy określenia zwierząt oraz przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji - do tej pory było to unormowane przepisami rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji - oraz uchylenia art. 830 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, jako że przepis ten stał się zbędny. Trzeba zgodzić się z poglądem, iż w świetle wymogów konstytucyjnych wszelkie wyłączenia spod egzekucji dotyczące zwierząt i rzeczy ruchomych potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego muszą być uregulowane na poziomie ustawowym. Obecnie są one unormowane w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Rozporządzenie jest aktem normatywnym, który może służyć jedynie wykonaniu ustawy. Stąd też proponowane zmiany są uzasadnione. Bogate orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego jasno precyzuje relacje między ustawą a rozporządzeniem. Słusznie zauważono, że art. 92 ust. 1 konstytucji przesądza, że upoważnienie do wydania rozporządzenia ma określać organ właściwy. Stopień precyzji wymagany przez ustawę zasadniczą wyklucza zatem tzw. upoważnienia blankietowe tudzież niekompletne. Przepisy upoważniające obarczone tego typu wadą, zwłaszcza naruszające wymóg szczegółowości pod względem przedmiotowym lub treściowym, nie czynią zadość wyżej przywołanemu wzorcowi konstytucyjnemu. Stosownie do przywołanego art. 830 Kodeksu postępowania cywilnego minister sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem rolnictwa oraz ministrem finansów jest obowiązany określić w rozporządzeniu, jakie przedmioty należące do rolnika prowadzącego gospodarstwo nie podlegają egzekucji. To upoważnienie nie dość, że nie zawiera żadnych wytycznych co do treści aktu wykonawczego, to przekazuje do uregulowania na poziomie podustawowym kwestie, które rzutują zarówno na prawo do sądu w tym jego aspekcie, który wiąże się z gwarancją wykonania prawomocnego orzeczenia, jak i na ochronę praw majątkowych wierzyciela, który decyduje się na wszczęcie egzekucji sądowej przeciwko rolnikowi prowadzącemu gospodarstwo rolne. Istotny jest również zauważony przez autorów projektu fakt, że część postanowień rozporządzenia z dnia 5 lipca 2017 r. wykracza poza przytoczoną delegację. Reasumując, przeniesienie do ustawy rozwiązań, które do tej pory były zawarte w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, o treści, która niemal odzwierciedla postanowienia zawarte w rozporządzeniu, poza korektami terminologicznymi lub redakcyjnymi, uznajemy za zasadne i konieczne, mając na uwadze potrzebę zapewnienia przejrzystości i prawidłowości usytuowania norm prawnych w tym zakresie.

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Wysoka Izbo!

Istotą regulacji jest przeniesienie katalogu przedmiotów niepodlegających egzekucji komorniczej, jeśli są to przedmioty rolnika prowadzącego gospodarstwo. Tu następuje przeniesienie z rozporządzenia ministra sprawiedliwości do aktu rangi ustawowej, czyli do Kodeksu postępowania cywilnego. Jest to bardzo istotne ze względu na hierarchię aktów prawnych, ze względu porządek konstytucyjny. Rozporządzenie powinno je tylko doprecyzowywać czy dodatkowo klarować, a nie stanowić.

Te chronione dobra to zwierzęta i przedmioty szczególnie istotne dla funkcjonowania gospodarstwa rolnego. Nie mamy do czynienia z kolizją.

Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Pan poseł Tomasz Zimoch przedstawi stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050. Panie Marszałku! Panie Senatorze! Przedkładany projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego powstał w wyniku indywidualnej petycji wniesionej do Senatu. Autor petycji słusznie zaproponował zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, bo - przytoczę - określenie zwierząt oraz przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, stanowi materię ustawową. Wymaga tego konstytucja i aż dziwne, że w Ministerstwie Sprawiedliwości od 4 lat tego nie zauważono. Nawet najlepsze rozporządzenie ministra nie powinno, co więcej, nie może zastępować ustawy. Koło Parlamentarne Polska 2050 popiera rozwiązanie zawarte w druku nr 1225. Wskazane jest przeniesienie niemal dokładne, na zasadzie: kopiuj i wklej regulacji dotyczących zwierząt i przedmiotów rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, które nie podlegają egzekucji, z rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 2017 r. wprost do kodeksu, jednocześnie wykreślając jeden z jego artykułów. Ten projekt, moim zdaniem, winien być przyjęty na zasadzie mini-max, minimum słów, maksimum dobrego prawa. Doceniamy pracę Senatu, warto jednak podkreślić obywatelską siłę petycji. Zna on zagadnienie doskonale, bo z tego co wiem, jest komornikiem. W uzasadnieniu petycji podkreślił: w rozporządzeniu nie powinno się regulować stanów faktycznych, do których wymagane jest wydanie ustawy. Rozporządzenie winno być wydawane jedynie w celu wykonania ustawy, nie zaś jej zastąpienia. Problematyka wyłączeń od egzekucji przedmiotów należących do rolnika powinna być uregulowana w ustawie. Proponowana ustawa spełnia postulat regulowania praw i obowiązków w akcie prawnym rangi ustawowej oraz postulat spójności systemu prawnego. Brawa dla autora petycji. Sejmowe ukłony raz jeszcze dla pana Kamila i zapraszamy do współpracy. Bardzo dziękuję. Na tym lista posłów, którzy prezentowali stanowiska klubów i kół, została wyczerpana. Przystępujemy do zadawania pytań. Czy ktoś z państwa posłów chciałby jeszcze do tej listy się dopisać? Jeżeli nie, zamykam listę. Ustalam czas na zadanie pytania - 1 minuta plus. W związku z tym proszę pana posła Mirosława Suchonia. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na pewno w trakcie rozpatrywania tego projektu, rozpatrywania petycji zastanawiali się państwo i badali, jak duży zasięg może mieć ta legislacja, jak wielu przypadków może dotyczyć projekt, który państwo skierowali do Sejmu.

Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę pana posła Jana Szopińskiego. Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Senatorze reprezentujący Senat RP! Wysoka Izbo! Za słuszny i celowy należy uznać projekt przeniesienia zapisów rozporządzenia do ustawy i tym samym nadanie im rangi ustawowej. Problem dotyczy bardzo trudnej materii, gdyż mówimy tutaj o egzekucji dotyczącej żywych zwierząt. Zatem będziemy mieli ustawowy obowiązek odstąpienia od egzekucji zakontraktowanej części stada stanowiącego podstawowy przedmiot produkcji rolnej danego gospodarstwa, czyli stada podstawowego. Natomiast wydaje się, że do uregulowania pozostał problem zobowiązań płatniczych. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Mam pytanie do pana senatora.

Pan poseł Ziejewski przedstawił problem, który występuje na wsiach szczególnie u dłużników i u wierzycieli.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi.

Bardzo proszę, panie ministrze.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sprawa, o której dyskutujemy, i sposób, w jaki prowadzimy tę debatę, rzadkie są w naszym parlamencie w ostatnich latach. Senat składa przedłożenie legislacyjne, które w swojej istocie jest aprobatą dla działań, które od kilku lat podejmuje minister sprawiedliwości.

Te zmiany, które są proponowane, w związku z powyższym mają aprobatę rządu, bo jak inaczej rząd może odnieść się do sytuacji, w której to parlament chce przenieść do aktu wyższej rangi rozwiązania, które ten rząd zaproponował i stosuje. W drugiej kolejności chciałbym podkreślić, że zmiany, które były wprowadzone w systemie egzekucji sądowej, również w zakresie ochrony rolników, dzisiaj można jednoznacznie ocenić jako wielki sukces naszego państwa. Już nie ma patologii, które były wiele lat temu krytykowane przez opinię publiczną, gdy widzieliśmy dramatyczne sceny, kiedy komornicy odbierali podstawowe przedmioty rolnikom czy generalnie gospodarstwom domowym. Jednocześnie, co mogę z dumą powiedzieć, pomimo wyeliminowania patologii, ograniczenia ich występowania, znacząco poprawiły się wyniki egzekucji. W kolejnych latach od wprowadzenia reformy odnotowaliśmy bardzo duże wzrosty skuteczności egzekucji, jeśli chodzi o każdy jej czynnik.

Czyli mamy do czynienia z ucywilizowaniem procesu egzekucji sądowej w Polsce. Mam nadzieję, że przepisy, które od kilku lat skutecznie chronią polskich rolników, dzięki podniesieniu rangi tych przepisów, przeniesieniu ich do ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, w jeszcze dalej idący sposób pozwolą rolnikom w spokoju regulować zaległości, jeśli takie będą powstawać, i w ten sposób stabilność funkcjonowania ich gospodarstw rolnych pomimo napotkanych trudności będzie zachowana. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu ministrowi.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym zwrócić uwagę, że jest to jeden z etapów, bo nie uporządkujemy tej całej sytuacji, która jest w obszarze rolnictwa i działalności rolniczej. Myślę, że kolejnym etapem winno być stworzenie funduszu gwarancyjnego, który na takie nieprzewidziane sytuacje by reagował i wspomagał rolników znajdujących się w takich sytuacjach. Ktoś komuś nie zapłacił, są terminy, ktoś nawet ucieka się do różnych instytucji parabankowych, gdzie pierwsze miesiące są wolne od oprocentowania, natomiast przy takim łańcuchu, kiedy rolnik sprzeda swoje artykuły rolne i nie uzyska zapłaty, skutkuje to takimi sytuacjami, że dochodzi do egzekucji komorniczych. Było rzeczywiście zastrzeżenie ze strony jednego klubu parlamentarnego odnośnie do tych zapisów, rzeczywiście instytucje finansowe również lobbowały, żeby utrzymać ten zapis.

Izby rolnicze uznały, że ten termin jest właściwy i one są w stanie dokonać oceny, żeby dać odpowiedź, wydać opinię dla komornika. Ilu na tę chwilę to dotyczy? To jest pytanie pana posła Ajchlera. Nie potrafię powiedzieć, ale obawiam się, że tych problemów będzie coraz więcej, panie pośle. Przy tych galopujących cenach środków produkcji rolnej i innych zobowiązaniach, które są nakładane na gospodarstwa rolne, tych problemów może być coraz więcej.

Oczywiście były to różnego rodzaju ustawki.

Dziękuję, panie marszałku. Dziękuję bardzo. Senator Ryszard Bober, który w tej kwestii reprezentował Senat Rzeczypospolitej, zakończył swoje wystąpienie. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, na podstawie art. 87 ust. 2 w związku z art. 90 ust. 1 regulaminu Sejmu, kieruje senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, zawarty w druku nr 1225, do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 32. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1569)

Ta ustawa składa się, można powiedzieć, z trzech części. Pisaliśmy ją, opracowywaliśmy ją wspólnie z ministerstwem edukacji narodowej, nauki i szkolnictwa wyższego. To nowe rozwiązanie dla studentów chętnych rozpocząć kształcenie na kierunkach medycznych. Druga część tej ustawy to rozwiązania związane z umożliwieniem większej liczbie uczelni kształcenia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Trzecia część to rozwiązania z zakresu kredytów studenckich, nazwijmy to, standardowych.

Szanowni Państwo! Te rozwiązania, które państwu proponujemy do rozpatrzenia w zakresie kredytu studenckiego, mają swoje podłoże, założenia czy pewne przesłanki związane z obecną sytuacją. Z jednej strony jest to sytuacja, w której ciągle jest, chociaż znacznie mniejsza, chęć migracji młodych lekarzy, młodych absolwentów kierunków medycznych, a z drugiej strony jest pewna luka, którą mamy w zakresie niewypełnienia limitów przyjęć na kierunki studiów, na kierunki odpłatne. Widzimy, że na kierunkach bezpłatnych, na których sukcesywnie zwiększamy limity przyjęć, ta konkurencja jest bardzo duża. Często dostają się czy nie dostają się, bo są poniżej tego progu, absolwenci szkół średnich, którzy uzyskali naprawdę dużo punktów, ale jednak poniżej tego minimalnego poziomu. Widzimy taką lukę, bo kształcenie na studiach medycznych jest ogromnie drogie.

Jest pewnie nieco inaczej niż jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy mieliśmy do czynienia z tą największą migracją lekarzy. Rzeczywiście zdecydowaliśmy się w tej sytuacji pewnych braków kadrowych wśród lekarzy na podjęcie działań, które z jednej strony zapewnią dalsze możliwości zwiększania limitów przyjęć na studia, z drugiej strony wprowadzą pewne rozwiązania lojalnościowe, które systemowo zwiążą absolwentów kierunków studentów medycznych z późniejszą działalnością zawodową w Polsce. Jeżeli popatrzymy dzisiaj na tę sytuację związaną z pewnymi formami lojalnościowymi, to jest to już kolejna z takich form, którą chcemy w pewien sposób związać lekarzy, lekarzy specjalistów.

Podobne rozwiązanie proponujemy w tej ustawie dotyczącej instytucji kredytu na studia medyczne. Ten kredyt to kolejna forma, poza kredytami studenckimi, wsparcia finansowego dla studentów, ale nie jest to forma wsparcia materialnego jak stypendia socjalne czy zapomogi. To, co bardzo ważne i co jest podstawowym założeniem, to to, że kredyt na studia medyczne dla tych chętnych do wybrania formy płatnej studiów będzie dostępny zarówno dla studentów na nowo rozpoczynających kierunki medyczne, jak również dla tych, którzy kontynuują studia płatne w Polsce. Chyba najważniejszym założeniem tej ustawy jest to, że studenci, którzy podejmą lub odbywają dzisiaj studia na kierunku lekarskim w języku polskim na warunkach odpłatności, jeżeli zdecydują się na skorzystanie z tego kredytu, to uzyskają możliwość jego częściowego lub całkowitego umorzenia po spełnieniu pewnych warunków ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Po pierwsze, po odpracowaniu czy przepracowaniu w Polsce po ukończeniu studiów minimum 10 lat w podmiotach leczniczych, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie tylko w podmiotach publicznych, bo mówimy tu generalnie o tych, które udzielają świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Drugi warunek to obowiązek uzyskania specjalizacji, tytułu specjalisty w tym okresie w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego.

Tu przewidzieliśmy, od czego to jest uzależnione i jakie powinny nastąpić przesłanki. Co więcej? To już może pewne kwestie techniczne, ale projekt ustawy przewiduje, że kredyty będą obsługiwane przez Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Tak jak wcześniej mówiłem, środki w tym funduszu będą pochodziły przede wszystkim z dotacji celowych z budżetu państwa określanych corocznie w ustawie budżetowej. Myślę, że ta dyskusja dzisiaj może być szersza niż tylko dotycząca kwestii związanych z kredytem studenckim.

To jedna z cegiełek, jeden z kolejnych elementów, które realizujemy. My nadal planujemy zwiększanie limitów przyjęć na bezpłatne studia medyczne.

Duży komponent w zakresie wsparcia procesów kształcenia, nowoczesnego kształcenia, rozwoju bazy dydaktycznej, rozwoju bazy klinicznej znalazł odzwierciedlenie w Krajowym Planie Odbudowy. Ogromne środki w wysokości prawie 3 mld zł zostaną przeznaczone przede wszystkim na to, żeby zwiększyć potencjał dydaktyczno-kliniczny uczelni do kształcenia większej liczby studentów, studentów medycyny generalnie. Ta ustawa w zakresie kredytu medycznego dotyczy dzisiaj wyłącznie kierunku lekarskiego, natomiast wiele rozwiązań, które proponujemy, dotyczy również kierunków medycznych i innych zawodów medycznych. Szanowni Państwo! Po konsultacjach tej ustawy, po rzeczywiście długiej dyskusji ze środowiskiem ta ustawa w zakresie kredytów medycznych została dobrze przyjęta przez środowisko akademickie.

Jeżeli pan marszałek pozwoli, oddam głos ministrowi nauki w zakresie spraw dotyczących zwiększenia liczby uczelni.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szczególny stan pandemii objawił jedną bardzo ważną rzecz - albo wzmocnił ten przekaz - bo obserwowaliśmy, że łatwiej wybudować szpital i wyposażyć go, niż odpowiedzieć na pytanie o lekarzy.

Oczywiście nie ma mowy o jakichkolwiek liberalizacjach, jeśli chodzi o standardy kształcenia na kierunkach lekarskich. Nad tymi procesami czuwa Polska Komisja Akredytacyjna. Chciałbym poinformować, że jesteśmy w trakcie procesu i jest już zgoda - czekamy na dokumenty - na akredytację dla PKA, jeśli chodzi o stronę amerykańską.

W myśl przedstawionego projektu pozwolenie będzie mogła uzyskać uczelnia, która według stanu na dzień złożenia wniosku posiada kategorię naukową A+, A lub B+ w dyscyplinie nauki medyczne lub dyscyplinie nauki o zdrowiu albo prowadzi studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68, i posiada minimalnie kategorię naukową C w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu. To są główne założenia, jeśli chodzi o tę przestrzeń właśnie dania większych możliwości kształcenia na kierunkach lekarskich, ale z troską o jakość. W kontekście całego projektu jeszcze warto zwrócić uwagę, że pojawiają się też rozstrzygnięcia, w zasadzie korygujemy pewne zapisy, jeśli chodzi o łatwość i zmniejszenie biurokracji dla studentów starających się o stypendia.

Po konsultacjach z bankami, ze środowiskiem studentów wprowadzamy też taką możliwość, żeby w tym pewnym ograniczonym aspekcie, zakresie banki mogły korzystać z naszego systemu POL-on i po prostu już nie musiały męczyć studentów, bo sami są w stanie to sprawdzić. I tu jest parę rozwiązań takich wręcz technicznych, które nie zmieniają istoty, natomiast zmniejszają biurokrację i wprowadzają rozwiązania właśnie takie bardziej przyjazne. Dziękuję bardzo panu ministrowi. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję. Proszę pana posła Krzysztofa Szulowskiego o przedstawienie stanowiska Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Panie i Panowie Posłowie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Prawa i Sprawiedliwości w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1569. Deficyt kadry medycznej to od lat bolączka naszego systemu ochrony zdrowia. Zwiększenie dostępności tych kadr to jeden z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości, począwszy od 2015 r. Stąd chociażby zwiększanie limitów przyjęć na studia medyczne. Tendencja jest wyraźnie wzrostowa, niemniej jednak zwiększenie tych limitów i inne działania wciąż nie zaspokajają rosnącego zapotrzebowania pacjentów na świadczenia zdrowotne, a efekty są widoczne po latach. Jednocześnie Rzeczpospolita Polska nadal pozostaje krajem, który stanowi atrakcyjny rynek pozyskiwania wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego, jednocześnie na tym tracąc. Wyjazd wykwalifikowanego lekarza skutkuje ograniczeniem dostępu do usług medycznych w kraju. Nie jest to też oczywiście dobre dla pacjentów, którzy oczekują wysokich standardów opieki medycznej i dostępu do wysokiej klasy specjalistów. Projektowane rozwiązania mają stanowić element realizowanej polityki zdrowotnej, jak również odpowiedź na deficyt kadry medycznej. Ważną propozycją jest uelastycznienie warunków dotyczących uzyskania przez uczelnie pozwolenia na utworzenie studiów na kierunku lekarskim oraz kierunku lekarsko-dentystycznym, co przełoży się na zwiększenie zarówno liczby uczelni prowadzących studia na tych kierunkach, jak również liczby studentów oraz absolwentów, którzy po ukończeniu studiów i wyspecjalizowaniu się będą zasilać szeregi polskiej kadry medycznej. Priorytetem będzie oczywiście zapewnienie kształcenia na odpowiednio wysokim poziomie z zachowaniem warunków i jakości kształcenia, co deklarował pan minister. Kolejna propozycja to wsparcie ze środków budżetu państwa osób podejmujących i odbywających odpłatne studia w języku polskim na kierunku lekarskim z obowiązkiem ich późniejszego odpracowania w podmiotach, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. A więc to tzw. zobowiązanie lojalnościowe. Projektowane rozwiązanie oprócz wsparcia finansowego studentów podejmujących i odbywających te studia przyczyni się do ograniczenia zjawiska emigracji absolwentów polskich uczelni będących lekarzami oraz wzrostu liczby lekarzy specjalistów, w szczególności w dziedzinach medycyny uznanych za priorytetowe. Ponadto wprowadzenie przedmiotowego wsparcia będzie szansą na uzyskanie zawodu lekarza przez osoby uzdolnione, które pomimo uzyskania dobrych wyników na egzaminie dojrzałości nie dostały się na studia na kierunku lekarskim w trybie stacjonarnym, a które m.in. z powodu braku wystarczających środków finansowych nie mogły podjąć tych studiów odpłatnie. Przy skorzystaniu przez takich studentów z kredytu na studia medyczne na kierunku lekarskim będzie możliwe nawet całkowite umorzenie kredytu pod warunkiem spełnienia przez lekarza łącznie następujących warunków, o których również mówił pan minister: obowiązku odpracowania studiów po ich ukończeniu przez okres nie krótszy niż 10 lat w ciągu 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów i obowiązku uzyskania tytułu specjalisty w tym okresie w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego. Inne istotne zmiany w projekcie ustawy to zróżnicowanie okresu przysługiwania świadczeń dla studentów w zależności od czasu trwania studiów, a także doprecyzowanie sposobu ustalenia tego okresu, uatrakcyjnienie systemu kredytów studenckich dla kredytodawców, usprawnienie procesu weryfikacji statusu studenta i doktoranta podczas obsługi kredytu studenckiego i kredytu na studia medyczne w oparciu o system POL-on. Projektowane rozwiązania służące wsparciu finansowemu studentów, zwiększeniu liczby uczelni prowadzących studia na kierunku lekarskim oraz kierunku lekarsko-dentystycznym, a więc i liczby studentów, ograniczeniu zjawiska emigracji absolwentów polskich uczelni będących lekarzami oraz wzrostu liczby lekarzy specjalistów, w szczególności w dziedzinach medycyny uznanych za priorytetowe, uważamy za dobre, łagodzące w perspektywie bolączki naszego systemu ochrony zdrowia. Dlatego klub Prawa i Sprawiedliwości popiera przedstawiony projekt. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Poseł Jerzy Hardie-Douglas przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Panowie Ministrowie! Jedną z przyczyn tego stanu, jak wiemy, jest dramatyczny deficyt lekarzy.

Powodem jest po części emigracja medyków. Obecnie już co trzeci rezydent rozważa emigrację z Polski. Jak podają sami autorzy projektu ustawy, w trakcie rządów PiS-u, od 2015 r. do 2019 r., łączna liczba lekarzy wykształconych w naszym kraju, których kwalifikacje zawodowe uznano w Unii Europejskiej oraz Norwegii, zwiększyła się o ok. 63%. Po zdaniu LEP-u większość lekarzy otrzymuje propozycję pracy w krajach Unii, Wielkiej Brytanii lub Norwegii. Oferuje im się lepsze zarobki, łatwiejszy dostęp do specjalizacji, lepsze warunki socjalne, szacunek, ochronę. Są dobrze wykształceni, znają języki, więc wyjeżdżają. Mamy jeden z najniższych w Europie współczynników zatrudnienia w sektorze opieki zdrowotnej.

Załamuje się ratownictwo medyczne. Źle opłacani młodzi lekarze są obarczani bardzo licznymi dyżurami. Opieka zdrowotna powinna być w najbliższych latach absolutnym priorytetem w wydatkach budżetu państwa. Tak się nie dzieje. Ewolucyjne podnoszenie udziału PKB w wydatkach na opiekę zdrowotną jest zdecydowanie zbyt wolne. W skali świata wydatki na opiekę zdrowotną są zwiększane co roku o ok. 5%, co powoduje, że mimo nieco większych nakładów na zdrowie w Polsce kraje rozwinięte jeszcze bardziej nam uciekają. Autorzy ustawy chcą zwiększyć liczbę studentów medycyny, równocześnie próbując zatrzymać lekarzy w Polsce. Proponują: zwiększenie liczby uczelni, które mogłyby otwierać studia na kierunkach lekarskich i stomatologii; zachęcanie młodzieży do studiowania medycyny, czemu ma służyć nowy system stypendiów i pożyczek; powstrzymanie emigracji lekarzy, czemu ma służyć możliwość powiązania pożyczek i kredytów z obowiązkiem ich odpracowania w Polsce. Autorzy proponują zarówno modyfikację istniejących kredytów studenckich, co rzeczywiście powinno spowodować ich większą dostępność, choćby przez ustalenie stałej marży kredytów studenckich na maksymalnym poziomie 2%, jak i wsparcie ze środków budżetu państwa osób podejmujących odpłatnie studia na kierunku lekarskim przy zobowiązaniu ich do późniejszego odpracowania kredytów w podmiotach, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Taki kredyt będzie szansą na uzyskanie zawodu lekarza przez osoby, które nieźle zdały maturę, ale nie dostały się na studia na kierunku lekarskim w trybie stacjonarnym. Często te osoby z powodu braku wystarczających środków finansowych nie mogą podjąć studiów odpłatnie. Taki kredyt na studia medyczne rzeczywiście może spowodować zdecydowane zwiększenie liczby osób studiujących w trybie niestacjonarnym. Przecież co roku zostają wolne miejsca na studiach niestacjonarnych, a liczbę tych miejsc można jeszcze znacznie zwiększyć. Oczywiście należy zadać sobie pytanie, czy te środki w sposób znaczący zahamują odpływ młodych lekarzy. Bez zdecydowanej zmiany jakościowej w finansowaniu opieki zdrowotnej, bez podnoszenia płacy rezydentom, bez ułatwiania im uzyskiwania miejsc specjalizacyjnych oni i tak będą opuszczać Polskę. Mimo wszystko jesteśmy skłonni te pomysły popierać. Jednak w projekcie ustawy pojawił się też inny pomysł - pomysł poszerzenia liczby uczelni mogących kształcić na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym o uczelnie zawodowe. Ustawa ma dopuścić uczelnie zawodowe do kształcenia na kierunkach przypisanych dotychczas studiom o profilu ogólnoakademickim. Kształcić lekarzy mogłyby uczelnie zawodowe, które prowadzą już studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu medycznego, czyli np. zawodu pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty itd. Kształcenie lekarzy wymaga, jak wiemy, wielokierunkowej kadry akademickiej, zarówno wielobranżowych teoretyków, jak i klinicystów. Wymaga wielu pracowni, zakładów badawczych, laboratoriów, różnorakiego sprzętu, ale przede wszystkim - solidnego zaplecza klinicznego. Tego uczelnie zawodowe nie zapewnią. Ustawa doprowadzi do stworzenia produktu lekarzopodobnego. W 2016 r. ówczesny wiceminister zdrowia, zresztą z PiS-u, Jarosław Pinkas, odpowiadając w Sejmie na pytania posłów, też z PiS-u, o działania resortu w sprawie zwiększenia liczby specjalistów, stwierdził: Odchodzimy od felczeryzacji medycyny. Obecny pomysł niestety idzie właśnie w tym kierunku. Otwierajmy nowe uczelnie medyczne, pomagajmy już istniejącym się rozbudowywać - mówił o tym pan minister - zwiększajmy nabór na studia, zachęcajmy do studiowania medycyny i do pozostawania po ukończeniu studiów w Polsce, wspierajmy studia niestacjonarne, ale nie próbujmy (Dzwonek) iść na skróty. Bardzo dziękuję panu posłowi. Proszę teraz panią poseł Anitę Kucharską-Dziedzic o przedstawienie stanowiska klubu parlamentarnego Lewica. Wysoka Izbo! Rządowe przedłożenie ma być odpowiedzią na dramatyczny brak lekarzy w polskim systemie ochrony zdrowia, czyli na brak elementarnego bezpieczeństwa polskich pacjentów. Już wiemy, że ta sytuacja przekłada się na utratę zdrowia i życia obywateli. Mamy dane liczone zgonami i dramatami ludzkimi.

Pozostałe są wynikiem paraliżu systemu ochrony zdrowia spowodowanego COVID-em, ale w części pewnie także brakami kadrowymi.

Pielęgniarek mamy 5,1 na 1 tys. mieszkańców, co również klasyfikuje Polskę na szarym końcu, tylko przed Turcją, Kolumbią, Meksykiem, Łotwą i Izraelem. Według danych OECD Polska ma nieco ponad 90 tys. lekarzy, z kolei według danych Naczelnej Izby Lekarskiej mamy w Polsce ponad 140 tys. lekarzy wykonujących zawód, nie licząc dentystów. Gdyby przyjąć tę liczbę do przeliczeń, można by powiedzieć, że mamy ok. 3,7 lekarza na 1 tys. mieszkańców, czyli zasadniczo jest lepiej. Gdzie jest zatem poukrywane te 50 tys. lekarzy? Część to efekt braku rzetelnego raportowania do wojewodów przez placówki służby zdrowia. Ponadto Naczelna Izba Lekarska być może zawyża swoje dane, bo część lekarzy, np. emeryci, aktywnie zawodu już nie wykonuje. Czy planowana w Polskim Ładzie podwyżka składki zdrowotnej dla wielu przedsiębiorców rozwiąże ten problem? PKB wydawanych na ochronę zdrowia. Według Lewicy to za mało, a droga dochodzenia do tego poziomu jest zbyt długa. Problemu ludzkiego to nie rozwiąże. Czego potrzebujemy? którzy się u nas osiedlą i będą leczyć polskich pacjentów. I potrzebujemy natychmiast zatrzymać wyjazdy lekarzy za granicę. Lekarzy rezydentów i lekarzy, którzy nie mają możliwości poszerzania kwalifikacji, nie chcieliście państwo słuchać. Dane Komisji Europejskiej pokazują, że w okresie od 2005 r. do 2019 r. 9671 razy kwalifikacje zawodowe zdobyte w Rzeczypospolitej Polskiej uznano w krajach należących do UE oraz Norwegii, co stanowi w stosunku do 2015 r. ok. 63-procentowy wzrost. Średniorocznie to 886 wykształconych w Polsce absolwentów kierunku lekarskiego. 27,2% badanych lekarzy zadeklarowało, że aktualnie rozważa możliwość emigracji.

Ale chcecie państwo więcej kształcić.

Macie zamiar rozszerzyć krąg uczelni uprawnionych do wnioskowania o uzyskanie pozwolenia na utworzenie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Zwiększenie liczby uczelni, które będą mogły ubiegać się o pozwolenie na prowadzenie tych studiów po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego, jest według KKP Lewicy obarczone wysokim ryzykiem obniżenia jakości kształcenia. Nie przybędzie nam przecież nauczycieli akademickich z racji wprowadzenia tych ułatwień. Połączone Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Zdrowia powinny rzetelnie nad tym pomysłem pracować. Drugi państwa pomysł to ułatwienia kredytowe i zróżnicowanie okresu przysługiwania świadczeń dla studentów w zależności od czasu trwania studiów, a także doprecyzowanie sposobu ustalania tego okresu. Myślenie o ułatwieniach dla studentów i młodych lekarzy, którym umorzy się kredyty studenckie pod warunkiem świadczenia pracy w polskiej ochronie zdrowia, z punktu widzenia ekonomicznego i ludzkiego jest dobre. W lipcu złożyłam interpelację w tej sprawie. Nie otrzymałam słowa odpowiedzi, ale rozumiem, że ten projekt jest tą odpowiedzią. Uatrakcyjnienie systemu kredytów studenckich i zwiększenie dostępności tego produktu dla studentów i doktorantów - tak, obniżenie jakości kształcenia - nie. Analogiczne prace powinny się toczyć w przypadku pielęgniarek i pozostałych (Dzwonek) zawodów medycznych. Nie tylko lekarzami polski system ochrony zdrowia stoi. Dziękuję bardzo. Teraz pan poseł Dariusz Klimczak przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Proszę bardzo, panie pośle. Wysoka Izbo! Ta ustawa to klasyczny przykład indolencji PiS-u w sprawie naprawy systemu ochrony zdrowia. Nawet, jeżeli diagnoza jest słuszna, to leczenie fatalne. Podczas tegorocznego wiosennego naboru na specjalizacje lekarskie minister przewidział 11, 13 miejsc więcej w stosunku do okresu poprzedniego. Czy tak postępuje państwo w dobie kryzysu pandemicznego? Czy tak postępuje państwo w czasie, kiedy mamy ogromny niedobór lekarzy?

Podobnie jest przy naborach na studia medyczne.

Ale jest drugi problem. Szacuje się, że ok. 2 tys. miejsc w każdym roku akademickim nie jest obsadzonych, co jest spowodowane m.in. faktem, że część z tych studiów jest płatna. Obecna liczba uczelni medycznych w Polsce jest dosyć duża, ale ich potencjał jest niewykorzystany.

Przecież już teraz uczelnie niemedyczne mogą kształcić lekarzy, wymogi są zminimalizowane. Pytanie: Czy dalsze ich łagodzenie jest pożądane i czy idziemy w dobrym kierunku? Konsekwencje obniżania standardów kształcenia lekarzy poniosą przecież pacjenci. Poza tym dzisiaj nie jest problemem prawo, które uniemożliwia otwarcie nowego kierunku lekarskiego na studiach, lecz fakt, że piekielnie trudno jest to zrobić przez jakąkolwiek inną uczelnię niż wyspecjalizowany uniwersytet medyczny. Wspomniane wyżej problemy to np. podpisywanie umów ze szpitalami, w których działają kliniki na bazie oddziałów szpitalnych. Oczywiście nie mam nic przeciwko temu, aby więcej uczelni mogło kształcić lekarzy, ale konieczne jest utrzymanie wysokich standardów studiów medycznych.

Kredyty studenckie na studia medyczne. Powiem szczerze, że już dawno nie widziałem takiego potworka legislacyjnego. Obwarowania w celu uzyskania kredytu z możliwością jego umorzenia są zbyt skomplikowane i jest ich zbyt wiele, a pochopne podpisanie takiego kredytu może wiązać się z ogromnymi kłopotami w przyszłości. Owszem, kredyt może być pomocny ale w skrajnych przypadkach może zamienić się w niewolniczy kontrakt na kilkanaście lat. Uważam, że z powodu licznych błędów w proponowanym projekcie liczba zainteresowanych skorzystaniem z tej formy wsparcia będzie niewielka. Dzisiaj potrzeba nam prostego, przejrzystego, powszechnego systemu wsparcia dla każdego, kto wybiera się na studia medyczne, lecz go na to nie stać. Po drugie, nie wolno łączyć kwestii umorzenia kredytu z wyborem specjalizacji jeszcze przed rozpoczęciem studiów. Przeciwnie, powinien istnieć osoby system wsparcia lekarzy, którzy decydują się na określoną specjalizację.

Wykładnia prawna tego przepisu może doprowadzić do wniosku, że wymóg udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych odnosi się wyłącznie do podmiotu (Dzwonek) wykonującego działalność leczniczą i nie dotyczy praktyki zawodowej. Już kończę, panie marszałku, ostatnie zdanie. Szanowni Państwo! Emigrację lekarzy można ograniczyć, wprowadzając przede wszystkim rozwiązania poprawiające warunki pracy lekarzy, nie tylko w aspekcie finansowym, ale też organizacyjnym, oraz ułatwiające im podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy. Dziękuję bardzo panu posłowi. Pan poseł Robert Winnicki przedstawi stanowisko Koła Poselskiego Konfederacja. Wysoka Izbo! W sprawie tej ustawy i w ogóle w tego dylematu, jakim jest kształcenie lekarzy, zderzają się dwa systemowe problemy, z którymi jako Polska mierzymy się 30 lat, i niestety kolejne ekipy rządowe albo nie chcą, albo nie potrafią podołać temu wyzwaniu. Zarówno jeśli chodzi o kształcenie lekarzy, jak i o stan ochrony zdrowia sytuacja sięgnęła, można powiedzieć, dna. Oczywiście współwinny temu jest kryzys COVID-owy i polityka COVID-owa rządu, to jest jasne, ponieważ lockdown ochrony zdrowia dzisiaj paraliżuje ją w jeszcze większym stopniu, niż to miało miejsce przed COVID-em. Natomiast, szanowni państwo, ten problem systemowy, z jakim się mierzymy, jest oczywisty.

To znaczy mamy ogromne zastępy ludzi kończących studia wyższe, którzy nie mają żadnych szczególnych kompetencji do tego, żeby uprawiać w życiu jakiś konkretny zawód. Taka jest prawda. Masowość wykształcenia w Polsce zbiegła się z radykalnym obniżeniem jakości tego wykształcenia. Fakt, że nie postawiono przez te ostatnie 30 lat.

Z drugiej strony priorytetowe, potrzebne całemu narodowi dziedziny i działki jak właśnie szkolnictwo medyczne, jak kształcenie lekarzy, których tak dramatycznie dzisiaj brakuje, po prostu leży.

Niezdrowa jest sytuacja, w której zyski są prywatne, a koszty są publiczne. Szanowni Państwo! To nie jest problem tylko i wyłącznie zawodów medycznych. Co więcej - czas mi się niestety kończy - problemem jest przede wszystkim struktura systemu opieki zdrowotnej.

Bez likwidacji systemu NFZ-etowskiego, bez likwidacji tego niewydolnego, rachitycznego systemu, który wprowadziła lewica 20 lat temu, po prostu nie uzdrowimy systemu ochrony zdrowia, w tym nie zachęcimy lekarzy do tego, żeby oni w Polsce pozostawali, żeby w Polsce leczyli. To jest fundamentalne i od tego trzeba zacząć. Dziękuję. Pan poseł Wojciech Maksymowicz przedstawi stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050. Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Bardzo współczuję urzędnikom służby cywilnej Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki, zwłaszcza współczuję ministrowi Murdzkowi, który zastąpił mnie na stanowisku sekretarza stanu, bo musi firmować coś, co jest bardzo słabo przygotowane, utopijne, bzdurne. Lojalnie muszą to wykonywać, co zrobić. Nie wnikam w złożone zapisy dotyczące kredytu studenckiego, w tej sprawie pięciu członków kierownictwa Ministerstwa Zdrowia jako kształconych w ekonomii to z pewnością lepsi ode mnie eksperci, ufam im. Na pewno jeden z nich by się przydał w jakimkolwiek następnym rządzie. Mają duże doświadczenie w zakresie finansowania. Natomiast cała reszta niestety jest problemem. Tę część projektu ustawy zresztą normalnie poddano procedurze legislacyjnej, jednak dodana naprędce pierwsza część ustawy ma dwa fatalne błędy. Pierwszy to właśnie pogwałcenie zasad legislacji. To jest zbyt poważna sprawa. Rządowy projekt ustawowy przeszedł przez cały Komitet Rady Ministrów i Radę Ministrów zupełnie bez najmniejszej konsultacji z ciałami uprawnionymi do konsultowania, a dotyczy kluczowych spraw. To jest niebywałe. Nie wolno tak gwałcić sposobu tworzenia prawa. Nawet Rządowe Centrum Legislacji nie miało szansy się wypowiedzieć w tej sprawie. Drugi fatalny błąd to zupełnie absurdalne założenie gwałcące wypracowane w powszechnym konsensusie w dawnym rządzie Zjednoczonej Prawicy rozwiązania ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Mam tylko 3 minuty, nikt z rządu przecież nie będzie zainteresowany uwagami byłego dziekana wydziału kształcącego lekarzy, prorektora do spraw Collegium Medicum. Proszę państwa, co to może obchodzić ministra Niedzielskiego, który kurs wiedzy medycznej przeszedł w kilka miesięcy, i to eksternistycznie? Co to obchodzi ministra edukacji i nauki skupionego na osłabianiu autonomii uczelni? Postanowiono o uniwersytecie w każdym powiecie - ma być i już. Oto w każdej zawodowej szkole nieakademickiej w oderwaniu od rzetelnej nauki medycznej.

Proszę państwa, wystarczy jedynie zatrudnić ludzi, którzy wykazują jakąkolwiek pracę w naukach o zdrowiu. Jest jeszcze jeden aspekt, który czyni ten projekt utopią i powoduje, że w zasadzie nie będzie on realizowany.

Już przeprosiłem swojego rektora, że będę musiał to tutaj mówić, broniąc uczelni i akademickości. Otóż pominięto opiniowanie środowiska akademickiego w części dotyczącej organizacji kształcenia medycznego. Uważam, że w dniu inauguracji roku akademickiego dokonano czegoś niebywałego, bo zamiast szacunku dla środowiska obrażono polskich profesorów medycyny. Ja też czuję się urażony takim podejściem. To niebywała arogancja, ale dalej będziemy robić swoje, będziemy kształcić prawdziwych lekarzy, rozwijając prawdziwą naukę medyczną. Dziękuję bardzo panu posłowi. Teraz pani poseł Magdalena Sroka przedstawi stanowisko koła Porozumienie. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Dzisiaj rozmawiamy na temat proponowanych zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym. Pan minister Gadomski pokrótce zaprezentował założenia dotyczące kredytu studenckiego. Te założenia co do kierunków nie są najgorsze, jeżeli chociażby kilku studentów z tego będzie chciało skorzystać. Z brakami lekarskimi borykamy się od lat i wszyscy po kolei próbujemy podejmować działania, żeby zwiększyć liczbę lekarzy. Zwiększanie limitów na studiach to jest dobry kierunek, ale do tego trzeba zachęty dla studentów i ułatwień. Natomiast rozmawiamy dzisiaj także o zmianach, które mają dotyczyć kształcenia lekarzy. Ten projekt zakłada, że uczelnie zawodowe będą mogły kształcić na kierunku lekarskim czy lekarsko-dentystycznym. Czy naprawdę chcemy stworzyć szkoły zawodowe dla lekarzy? Pan minister Murdzek powiedział, że chęć zwiększenia ilości kadr medycznych to nie będzie obniżenie jakości. Przecież w tej chwili studia medyczne to są studia, które bez badań naukowych, bez badań klinicznych czy bez wykorzystania najnowszych technologii nie przyniosą zakładanych efektów. Ci ludzie w białym miasteczku codziennie siedzą przed kancelarią premiera. Czy naprawdę takie zmiany muszą być wprowadzane bez żadnych konsultacji z zainteresowanym środowiskiem? Przecież to są fundamentalne zmiany. Po prostu to się im należy, żeby takie konsultacje w tak ważnym temacie prowadzić w sposób bardzo szeroki. Tak że nie wydaje mi się, by chęć podniesienia ilości poszła w parze z jakością. Na tym lista posłów zapisanych do głosu w celu wygłoszenia stanowisk klubów i kół została wyczerpana. Do pytań zapisało się 21 spośród państwa posłów. Jeśli ktoś jeszcze chciałby się dopisać do listy, to bardzo proszę. Jeszcze nigdy tak się nie zdarzyło, żebym reglamentował czas. Natomiast ze względu na ilość i prośby, aby nie było tzw. obsuwy czasowej, ustalimy czas na 1 minutę, a jeśli będzie trzeba dłużej, to oczywiście tak. Jako pierwszy pytanie zada pan poseł Paweł Hreniak. Panie Ministrze!

A więc mamy zauważalną tendencję wzrostową, ale niestety nadal mimo pozytywnej zmiany nie zaspokaja to rosnącego w Polsce zapotrzebowania na biały personel medyczny. W związku z tym moje pytanie do pana ministra: Jak ministerstwo szacuje, o ile należałoby zwiększyć liczbę miejsc na uczelniach medycznych, tak aby w pełni zaspokoić nasze potrzeby w odniesieniu do opieki zdrowotnej? Pytanie zada pan poseł Rafał Adamczyk. Wysoka Izbo! Dzisiaj rozmawiamy o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw. Jak wielkie są braki w Polsce wśród kadry lekarskiej, doskonale wszyscy wiemy. Każda forma wsparcia w celu zwiększenia liczby lekarzy w naszej opiece zdrowotnej powinna być przede wszystkim skuteczna. Panie ministrze, czy ministerstwo obliczyło, jaka liczba studentów kierunków lekarskich skorzysta z propozycji dotyczącej kredytów studenckich, która została zaprezentowana w projekcie ustawy? Pytanie zada pan poseł Jan Szopiński. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Próby majstrowania przy szkolnictwie wyższym i tworzenia furtek prawnych w żaden sposób nie rozwiązują problemu braków w kadrze lekarskiej, przed którym stanęliśmy w wyniku wieloletnich zaniedbań. W niedługim odstępie czasu prezentujemy kolejną ustawę, tym razem mającą na celu wprowadzenie na uczelnie techniczne i zawodowe najpierw kierunków pedagogicznych, teraz kierunków lekarskich. Jednocześnie tworzy się przepisy zamykające drogę do kształcenia w podmiotach dla nauczycieli z 70-letnim doświadczeniem w danej dziedzinie. Nie wiem, czy sprzeczność tych przepisów wynika z działalności jakiegoś lobby, czy jedynie z braku wyobraźni urzędników tworzących kolejne regulacje prawne. Pytanie do pana ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi pisemnej: Jak należy rozumieć zablokowanie utworzenia w Bydgoszczy uczelni medycznej w oparciu o istniejące zaplecze do kształcenia lekarzy, zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym, w świetle tworzonych (Dzwonek) nowych przepisów otwierających taką drogę dla uczelni technicznych, które do tej pory miały niewiele wspólnego z kierunkiem kształcenia lekarskiego? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Pytanie zada pan poseł Zdzisław Wolski. Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Minister Gadomski mówił, że projekt był konsultowany z samorządem lekarskim, ale powiedział tylko część prawdy.

Jestem z Częstochowy.

Jest ogrom ludzi, pozytywne stanowisko prezydenta, rady miasta, dyrektorów szpitala i lokalnej izby lekarskiej. Mam nadzieję, że panowie ministrowie, szczególnie pan minister nauki, oczywiście również Państwowa Komisja Akredytacyjna, korzystając z tej ustawy, w trybie szybkim umożliwią otworzenie wydziału lekarskiego w Częstochowie, bo cały okręg częstochowski na to bardzo czeka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią poseł Joannę Fabisiak o zabranie głosu. Wysoka Izbo! Lekarze polscy wyjeżdżają i są rozrywani. A dlatego że są świetnie wykształceni, są po prostu dobrymi fachmanami.

Uczelnia, której specjalnością jest nauka o zdrowiu, a ma uczyć chirurgii - nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, że to są duże pieniądze, i nie mam czasu na rozwijanie tego wątku, ale trzeba się nad tym zastanowić. Sprawa druga to jest sprawa programu. Rozumiem, że za 2 lata, czyli w 2023 r., w październiku te uczelnie by ruszyły, prawda? A jeszcze nie było konsultacji. Najpierw konsultacje, potem programy, potem programy zaakceptowane przez ministerstwo - wiadomo, że to długo trwa - a potem wreszcie wyposażenie tych szpitali w stosowne. Pieniądze i czas - te dwie rzeczy, wydaje mi się, są ułomnie potraktowane w ustawie, a tym samym musi na tym w przyszłości cierpieć pacjent, ale i lekarz, bo lekarz też cierpi, jak nie może dobrze leczyć pacjenta. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze!

W związku z tym pytanie: Co na te 8 lat państwo przewidujecie? Czy państwo chcielibyście z tego skorzystać?

Czy tutaj nie należy dążyć do rozwoju innych zawodów medycznych, które miałyby pomóc czy też uzupełnić braki?

Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo! Po przeprowadzeniu konsultacji publicznych pomysłodawcy projektu dodali nowe, niezwykle istotne dla środowiska lekarzy i lekarzy dentystów, zapisy. Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich proponowane zapisy powinny zostać skonsultowane z samorządem lekarskim, ponieważ bardzo kontrowersyjne poprawki dotyczące rozszerzenia katalogu uczelni mogących kształcić lekarzy są zmianami istotnymi dla podmiotów, z którymi uprzedni tekst wcześniej konsultowano, a więc powinien on wrócić do konsultacji. Wynika to również z regulaminu pracy Rady Ministrów. Tak się nie stało. Jest to jaskrawe naruszenie zasad tworzenia aktów prawnych. Zwraca na to uwagę m.in. Rządowe Centrum Legislacji. Pytanie: Dlaczego państwo lekceważycie przepisy prawa jasno opisujące proces legislacyjny? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią poseł Katarzynę Lubnauer. Panie i Panowie Posłowie! Panie Marszałku! O tym, że brakuje lekarzy, wszyscy wiemy. Co więcej, kolejne rządy, zdając sobie z tego sprawę, zwiększały liczbę miejsc na studiach lekarskich.

Wiemy też, że w ten sposób bardzo szybko nie uzyskamy rezultatu, jakim są wykształceni lekarze. Dlatego być może na studiach w wyższych szkołach zawodowych należy zwiększyć kształcenie nie lekarzy, tylko np. asystentów medycznych, po to żebyśmy mieli ludzi, którzy chociaż częściowo odciążą lekarzy od niektórych czynności, nazwijmy je papierkowymi czy biurowymi. Problem polega na tym, że nie wykształcimy dobrego lekarza bez szerokiej bazy szpitalnej związanej z dużym ośrodkiem miejskim, bez uczelni, która prowadzi badania naukowe nie tylko w tej dziedzinie, w której kształci, ale również w pokrewnych. Możemy wykształcić - bo macie taką skłonność do tego, żeby dawać dodatkowe uprawnienia szkołom zawodowym - historyka, co do którego wiedzy nie mamy pełnego zaufania. Możemy wykształcić ekonomistę, który czasami będzie popełniał błędy, ale czy naprawdę chcemy mieć lekarzy, którzy będą mieli inny dyplom? Pytanie zada pani poseł Małgorzata Pępek. Wysoka Izbo! W procedowanej ustawie nie było mowy o zmianie, która zakłada, że nie tylko uczelnie akademickie, ale też wyższe szkoły zawodowe będą mogły starać się o pozwolenie na kształcenie medyków. Została ona wprowadzona na późniejszym etapie prac nad projektem nowelizacji. Czy tak ma wyglądać proces legislacyjny? Przedstawiciele izb lekarskich wprost komentują takie działania, posługując się wyrażeniem, że ręce opadają.

To jest niezwykle ważne. W jaki sposób rząd chce zagwarantować, że poziom kształcenia medyków nie ucierpi? W medycynie szczególnie powinno chodzić o jakość nauczania. W końcu to obywatele są potencjalnymi późniejszymi pacjentami takich medyków, w rękach których leży nasze zdrowie i życie. Bardzo dziękuję. Czy na sali jest pan poseł Waldy Dzikowski? Nie widzę. Proszę teraz pana posła Aleksandra Miszalskiego. Też nie ma. Pani poseł Magdalena Sroka. Zapraszamy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Również oni powinni mieć taką możliwość, co ułatwiłoby im przejście przez cały proces edukacyjny. Drugie pytanie: Czy planują państwo szerokie konsultacje w zakresie proponowanych zmian dotyczących sposobu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów? Czy tak przeprowadzony proces legislacyjny będzie spełniał podstawowe standardy? Dziękuję. Bardzo dziękuję.

Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Analizie poddano także chęć wyjazdu tych medyków, którzy pracują aktualnie w kraju.

Tak mówiła posłanka Prawa i Sprawiedliwości do lekarzy. Tak Prawo i Sprawiedliwość traktowało środowisko medyczne. Panie ministrze, kiedy wreszcie rzeczywiście te środki finansowe na wynagrodzenia środowiska medycznego będą odpowiadały wartości pracy tego środowiska? Pytanie zada pan poseł Marek Hok. Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! To dzięki tej zachęcie młodzi lekarze na zaproszenie „wyjeżdżajcie” wyjeżdżali i dalej wyjeżdżają. Myślę, że właśnie autorytet pani poseł, pani poseł z partii rządzącej spowodował, że uwierzyli w te słowa i wyjechali. Dzisiaj, proszę państwa, mamy ok. 140 tys. lekarzy, którzy pracują zawodowo, a w tej grupie jest ok. 30 tys. lekarzy emerytów. Jeżeli oni zrezygnują w ciągu jednego dnia z pracy, pada cały system ochrony zdrowia. Nie pomogą kredyty, nie pomogą bony lojalnościowe, lekarzy po prostu nie ma. Dlatego pytanie: Czy rzeczywiście nie należy sięgnąć do zmian w edukacji i w szkoleniu lekarzy?

Wysoka Izbo! Dziękuję panu ministrowi za przygotowanie tego projektu, bo nareszcie studenci od 1 października, czyli od dzisiaj, mogą uzyskać dofinansowanie do kosztów kształcenia na płatnych wydziałach lekarskich. Szanowni państwo, wszystkim nam zależy na tym, aby jakość kształcenia została utrzymana. Jak wiemy, zawód lekarza i kształcenie w zawodzie lekarza jest zawodem regulowanym przez Unię Europejską. W związku z powyższym mam pytanie do pana ministra: Czy otwarcie kształcenia na tych uczelniach, o których państwo mówicie, które mają doświadczenie w kształceniu np. fizjoterapeutów, diagnostów czy jeszcze innych zawodów medycznych, będzie odbywało się zgodnie ze standardami, które zostały przyjęte zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce?

Bardzo dziękuję. Pytanie zada pan poseł Dariusz Klimczak. Wysoka Izbo! Pierwsze pytanie, krótkie, dotyczy właśnie tych niewykorzystanych miejsc na studiach medycznych. Druga sprawa to jest kontynuacja tej myśli, którą wyrażał pan poseł Hok. Czy ministerstwo planuje, czy prowadzi prace w kierunku całkowitej reformy systemu kształcenia, szczególnie jeżeli chodzi o specjalizacje, ich tryb, liczbę, nabór? Czy wreszcie także chce połączyć to z niedawną zmianą legislacyjną dotyczącą map potrzeb zdrowotnych, planu transformacji? Czy państwo planują to połączyć? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Pytanie zada pan poseł Marek Rutka. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zacznę od zacytowania Mateusza Morawieckiego.

Koszt, jaki musi ponieść budżet państwa, czyli, mówiąc inaczej, każdy z nas, na wykształcenie lekarza, to ok. 1 mln zł. Aby uzmysłowić skalę tych wydatków - jest to kwota, za którą w każdym z województw można by wybudować przynajmniej po dwa nowoczesne szpitale. Zamiast opracować i wdrożyć atrakcyjne warunki wynagrodzeń i płacy, szczególnie dla absolwentów uniwersytetów medycznych, tak aby nie byli [[Dzwonek]] zmuszeni do emigracji, pogłębiając jednocześnie dramatyczną sytuację kadrową w polskim systemie ochrony zdrowia, rząd proponuje obniżenie standardów kształcenia. Jeszcze parę sekund. W projekcie zmiany ustawy czytamy, że na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów kształcących do zawodu lekarza i lekarza dentysty będą uprawnione uczelnie, które dziś przygotowują do wykonywania zawodu m.in. farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty, fizjoterapeuty. W praktyce to oznacza, że przyszli lekarze będą mogli być kształceni na akademiach wychowania fizycznego, czyli tam, gdzie dziś kształci się fizjoterapeutów - z całym szacunkiem oczywiście dla fizjoterapeutów.

Może od razu nazwijmy to programem felczer+ i wszystko będzie jasne. Dziękuję bardzo. Panią poseł Fabisiak prosilibyśmy o wyciszenie rozmowy lub przeniesienie się poza salę sejmową. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Myślę, że warto, aby z tej mównicy padło kilka ważnych informacji odnoszących się do wyjazdów i emigracji lekarzy, którzy kształcą się w Polsce. Otóż, proszę państwa, żebyście państwo mieli świadomość, że do Polski przyjeżdżają młodzi ludzie z Unii Europejskiej, kształcą się tutaj przez okres 6 lat i wracają do swojego kraju, po prostu biorą zaświadczenie o ukończeniu studiów i wracają do swojego kraju. W tej statystyce tzw. lekarzy wykształconych na polskich uczelniach jest ich ok. 1 tys. w skali roku. Chciałabym o to w pierwszej kolejności spytać.

Chcę zapewnić - z całą pewnością nie będzie tak, że każdy powiat będzie kształcił przyszłych lekarzy.

O to chciałam spytać.

Pytanie zada pani poseł Anna Dąbrowska-Banaszek. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie!

Każde działanie, którego celem jest zwiększenie kadry lekarskiej, jest ważne.

Jaka jest przewidywana większa ilość studentów, a w przyszłości lekarzy?

Bardzo dziękuję. Pytanie zada pan poseł Krzysztof Paszyk. Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Przedstawiciele PiS-u przed chwilą chwalili się, jak zwiększa się ilość miejsc na studiach o kierunku medycznym. To jest, panie i panowie posłowie, początek.

Mówię o dokumentacji, o niepotrzebnej biurokracji, którą mogą się zająć inni pracownicy.

Bardzo dziękuję. Pytanie zada poseł Wojciech Maksymowicz. Do tej pory nie dostałem oczywiście odpowiedzi. Za chwilę opozycja powie: jest za mało lekarzy, zobaczcie, to wszystko wasza robota.

Wiem, że tam jest trochę niżej. Efekt jest taki, że nie stosujemy działań, które mogą sprawić, że lekarzy będzie odpowiednio dużo tam, gdzie powinni być. To jest problem.

To jest problem. Dziękuję bardzo panu posłowi. Do wygłoszonych oświadczeń oraz zadanych pytań odniesie się podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pan minister Sławomir Gadomski. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję za te pytania. Bardzo cenne pytanie zadał pan poseł Hreniak. Odpowiedź pewnie nie jest taka oczywista. Jeżeli popatrzymy sobie na liczbę emerytów czy liczbę lekarzy wchodzących w wiek emerytalny, to żeby była w Polsce zastępowalność, powinniśmy kształcić, powiedzmy, między 6 a 8 tys. lekarzy.

Natomiast jeżeli patrzymy generalnie na potrzeby systemowe, na starzenie się społeczeństwa, na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne, to w oczywisty sposób nadal chcemy zwiększać tę liczbę lekarzy, bo dobrze też wiemy, że w systemie pracuje kilkadziesiąt tysięcy - tu padała liczba 30 tys., według moich szacunków to nawet więcej, ok. 40 tys. - lekarzy, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym.

Konkludując, nadal chcemy zwiększać limity przyjęć na studia, myślę, że do kilkunastu tysięcy rocznie na pewno.

Oczywiście dzisiaj opieramy się wyłącznie na pewnych szacunkach. Dzisiaj studentów studiujących na odpłatnych studiach w języku polskim jest łącznie 7 tys. Pod tym kątem przygotowaliśmy ocenę skutków regulacji, zakładając, że mogą skorzystać wszyscy.

Natomiast w oczywisty sposób bezpiecznego szacunku podać nie umiem. Chciałbym, żeby skorzystało z tego jak najwięcej osób. Co do niewykorzystanych miejsc, jak już jesteśmy przy tych liczbach miejsc. Nie wiem, panie pośle, skąd te dane.

Limity na studiach bezpłatnych zostały wypełnione praktycznie w całości. Pytał pan o rozwiązania.

Również w uzasadnieniu się znalazło, że zakładamy, że pewna część tych miejsc jest niepokryta właśnie dlatego, że studenci nie decydują się, bo nie stać ich na ten kredyt.

Jestem przekonany, że jeżeli tylko to zainteresowanie będzie wysokie, to w następnym roku te limity zwiększymy jeszcze bardziej.

W ostatnich 2 latach przede wszystkim zmniejszyliśmy liczbę limitów na studia anglojęzyczne, zwiększając jednocześnie przede wszystkim limity przyjęć na studia bezpłatne w języku polskim.

Bazujemy na pewnych uproszczeniach. Uproszczeniem są zaświadczenia pobierane przez absolwentów w izbie, uproszczeniem tak dużym, że wyciąganie z nich wniosków jest rzeczywiście daleko idącym uproszczeniem, bo po pierwsze, te zaświadczenia absolwenci mogą pobierać wielokrotnie, po drugie, to nie znaczy, że gdziekolwiek wyjechali, a po trzecie, faktycznie, jak słusznie pani poseł zauważyła, te zaświadczenia pobierają również studenci studiów anglojęzycznych, którzy, jak wiemy, niestety w większości wyjeżdżają z Polski. Ale tak jak mówiłem, my te limity zmniejszamy, zwiększając jednocześnie limity przyjęć na studia w języku polskim, aczkolwiek też nie zależy nam na takim drastycznym ograniczeniu tych limitów, bo nie traktujmy tych studentów jako studentów drugiej kategorii. Oni wnoszą umiędzynarodowienie uczelni, wnoszą pewne kontakty zagraniczne, umożliwiają wymianę z innymi krajami. A więc dalej chcemy to utrzymać, aczkolwiek nie musimy przyjmować ich tak dużo jak do tej pory. Pojawiły się również z tej mównicy postulaty dotyczące standardu kształcenia, pewnego skrócenia długości kształcenia.

Raczej opinia środowiska akademickiego jest dzisiaj taka, że wraz z nowymi formami kształcenia, wraz z rozwojem właśnie kształcenia w zakresie technik symulacji, wraz z rozwojem wieloprofilowych centrów symulacji - przy wszystkich uczelniach medycznych już dzisiaj powstały takie centra - ten program dzisiaj jest rozbudowywany, a nie skracany. Przypominam również, że Komisja Europejska wymaga, żeby kształcenie na studiach medycznych było co najmniej 5-letnie.

W naszej ocenie dzisiaj skrócenie cyklu czy studiów, czy kształcenia podyplomowego raczej nie idzie w parze z tym, o co sami państwo postulowaliście, czyli z najwyższymi standardami kształcenia, aczkolwiek pewnie - tu jestem w stanie się zgodzić - musimy zastanawiać się nad pewnym uelastycznieniem form kształcenia, nad pewnymi innymi możliwościami kształcenia doskonalącego. Sami zawarliśmy pewne postulaty i pewne zmiany w tym zakresie w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty w roku 2020, gdzie właśnie takie uelastyczniające formy zostały wprowadzone.

Pan minister nauki mówił, że musi wyjść, więc spróbuję wziąć ciężar odpowiedzialności za te pytania związane z rozszerzeniem liczby uczelni. Szanowni Państwo! Po pierwsze, nie możemy łączyć liczby uczelni, które będą mogły aspirować do tego, żeby kształcić lekarzy, z jednoznacznym obniżeniem standardu kształcenia. Dzisiaj stanowisko ministra zdrowia jest jednoznaczne: i standard kształcenia, i standard umożliwiający w ogóle rozpoczęcie kształcenia lekarzy pozostanie niezmienny.

Szanowni Państwo!

Nie będę wymieniał uczelni z nazwy. Natomiast są to postępowania, które toczą się od kilku lat. One spełniły wymóg formalny odnośnie do możliwości aspirowania do tego, żeby kształcić lekarzy, natomiast do dzisiaj nie przeszły procedury akredytacyjnej, bo jest ona tak skomplikowana. Pojawiły się pytania o pewne wymogi i wydatki inwestycyjne. Absolutnie tak, szanowni państwo, dzisiaj każda uczelnia, która zechce kształcić lekarzy, musi rozpocząć od pewnej analizy opłacalności.

To ogromny wydatek, to ogromne wyzwanie.

Ta ustawa dzisiaj w ogóle tego nie neguje. Te wymogi dalej będą musiały być spełnione. Porównałem to dzisiaj na posiedzeniu podkomisji i może jeszcze raz tego porównania użyję. To, że dzisiaj każdy z nas na tej sali może zostać pilotem, to jest fakt. Ale nie wiem, czy ktokolwiek z nas podjąłby się tego trudu.

Tę samą żmudną drogę będą musiały przejść uczelnie starające się o to, żeby kształcić lekarzy.

Tak że z punktu widzenia Ministerstwa Zdrowia dzisiaj absolutnie nie dopuszczamy myśli, że jakiekolwiek standardy kształcenia na takich uczelniach miałyby być inne niż na tych, które kształcą dzisiaj, że jakiekolwiek standardy wejścia do kształcenia, czyli spełnienia tych wymogów formalnych i merytorycznych, miałyby być inne, a już w szczególności niższe niż dzisiaj.

Jeżeli tylko znajdzie się kilka uczelni, które spełnią te wyśrubowane wymogi i będą w stanie kształcić lekarzy, to będzie to, jestem przekonany, wartość dodana dla całego systemu ochrony zdrowia. Tak jak mówię, wierzę w to głęboko, że ta jakość nie ucierpi.

Szanowni Państwo! Pan poseł mówił, że zmniejsza się liczba miejsc specjalizacyjnych. To nieprawda, ona się zwiększa, minimalnie się zwiększa. To na pewno trzeba odnotować. Natomiast ta liczba jest dostosowana do liczby absolwentów, którzy kończą uczelnie.

Na to również będziemy kierować dodatkowe nakłady w ochronie zdrowia. Myślę, że nikomu na tej sali, w szczególności ekspertom w ochronie zdrowia, nie zależy na tym, żebyśmy skupili się wyłącznie na zwiększeniu liczby miejsc specjalizacyjnych tam, gdzie dzisiaj jest ogromne zainteresowanie.

Jeżeli potrzebujemy onkologów, to rzeczywiście tam chcemy zwiększać tę aktywność. Szanowni Państwo! Konkludując, cieszę się z tej pozytywnej opinii co do kwestii związanych z kredytami medycznymi.

Oczywiście, panie ministrze. Właśnie chciałem panu podziękować za to, że pan dźwignął także pytania skierowane do pana ministra Wojciecha Murdzka, który opuszczając Wysoką Izbę, przez szacunek dla obecnych posłów mógł przynajmniej powiedzieć, że musi wyjść, albo w jakiś inny sposób zasygnalizować ten fakt.

Kończąc wątek, pan poseł Klimczak jeszcze tutaj wspomniał i chyba podniosła to też Naczelna Rada Lekarska. Panie pośle, nie zgadzam się z teorią, że zawieramy jakiś niewolniczy kontrakt. Kredyt medyczny jest fakultatywny. Przepraszam, racja. Uważam, że jest to pewien benefit, z którego ktoś albo zechce skorzystać, albo nie zechce. Co więcej, pokazujemy priorytetyzację kształcenia na kierunkach lekarskich, bo dzisiaj niestety, być może to się kiedyś zmieni, żaden informatyk nie może liczyć na to, że otrzyma kredyt na kształcenie na kierunku informatycznym. Jestem ekonomistą i niestety nie mogłem na to liczyć; dzisiaj żaden ekonomista na to liczyć nie może.

Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, zawarty w druku nr 1569, do Komisji Zdrowia oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 33. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1570) Proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów pana Piotra Patkowskiego o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić Wysokiej Izbie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

Dzięki proponowanym zmianom jednostki zyskają także możliwość korzystania z nowoczesnych narzędzi informatycznych, a użytkownicy sprawozdań będą mogli w szybki sposób pobierać, analizować i interpretować potrzebne im dane. Ponadto ta ustawa usprawnia, daje dodatkowe kompetencje Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Niedawno wprowadzona zmiana powodowała, że takie sprawozdania musiały być podpisywane elektronicznie przez wszystkich członków zarządu, co powodowało szereg problemów dla NGOs, także z mniejszych miejscowości, gdzie złożenie takiego podpisu elektronicznego i zebranie wszystkich przedstawicieli członków zarządu było problematyczne. Przedmiotowy projekt wprowadza tu zmianę.

Dzięki temu zarządy wieloosobowe będą mogły sprawniej podpisywać takie sprawozdania i nie będzie wymagany od wszystkich takich członków obowiązek posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Druga poważna zmiana, która jest dokonywana w przedmiotowym projekcie, to wprowadzenie obowiązku dla emitentów, którzy są zobowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych w jednolitym formacie elektronicznym standardowym dla państw członkowskich Unii Europejskiej i jest to tzw. format ESEF. Dla pozostałych jednostek stosujących międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej ustawa wprowadza obowiązek stosowania jednolitego formatu sprawozdawczego ESEF lub innego przeszukiwalnego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności.

Trzecia zmiana postulowana przez rynek, dość techniczna, ale ważna dla tych podmiotów, to zmiana dotycząca konsolidacji sprawozdań finansowych przez alternatywne spółki inwestycyjne. Biorąc pod uwagę charakter działalności ASI, obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez te jednostki nie zawsze jest uzasadniony. Nowelizacja ustawy o rachunkowości proponuje więc uproszczenia w tym zakresie. I ostatnia grupa zmian to zmiany, o których już wspominałem, czyli zmiany w działalności Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego w dużej mierze sprowadzające się do ucyfryzowienia działalności PANA. Po pierwsze, jest to doprecyzowanie przepisów ułatwiające odbywanie posiedzeń zdalnych oraz podejmowanie uchwał w trybie obiegowym przez radę agencji i organy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Po drugie, chodzi o umożliwienie przeprowadzania przez agencję kontroli zdalnych w firmach audytorskich w przypadku wszystkich kontroli oraz wprowadzenie kontroli zdalnych jako podstawowej formy działalności. I po trzecie, dotyczy to umożliwienia załatwiania spraw dotyczących obsługi listy firm audytorskich za pomocą systemu teleinformatycznego. Ponadto ułatwiamy komunikację pomiędzy agencją a firmami audytorskimi w trakcie kontroli, zmniejszamy pracochłonność w przygotowaniu dokumentów do kontroli poprzez korzystanie w znacznie większym stopniu z dokumentów w postaci elektronicznej zamiast papierowej, ograniczamy koszty kontroli po stronie zarówno firm audytorskich, jak i agencji oraz ograniczamy czasochłonność w załatwianiu spraw. Na koniec jeszcze raz podkreślę, że projekt był szeroko konsultowany. Odpowiada na postulaty naprawdę wielu podmiotów sprawozdawczych, szczególnie drobnych i niewielkich NGO-s. W związku z tym uprzejmie proszę Wysoką Izbę o przyjęcie projektu ustawy w wersji zaproponowanej przez rząd. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Szanowni Państwo! Celem projektu jest dostosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej oraz rewizji finansowej do nowych możliwości technologicznych. Wprowadzone zmiany mają m.in. ujednolicić format sprawozdań finansowych emitentów. Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych, z którym mamy obecnie do czynienia, wywiera istotny wpływ także na rachunkowość i pracę biegłych rewidentów. Możliwość korzystania z nowoczesnych narzędzi informatycznych sprawia, że jednostki łatwiej mogą wywiązywać się ze swoich obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Użytkownicy tych sprawozdań mogą natomiast w szybki sposób pobierać, analizować i interpretować potrzebne im dane. Dodatkowo cyfrowa transformacja życia gospodarczego została przyspieszona przez pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2. W tym kierunku podąża także prawo europejskie. Pragnę podkreślić, że projekt niniejszej ustawy jest zgodny z rozporządzeniem Unii Europejskiej, którego założeniem jest uporządkowanie elektronicznego formatu raportowania. Rozwiązanie stosowane na podstawie tego rozporządzenia ma poprawić dostępność i ułatwić porównywalność sprawozdań finansowych. Nowelizacja ustawy przewiduje także zmiany w zakresie podpisywania sprawozdań. Projektowane przepisy mają na celu wprowadzenie ułatwień dla kierowanych przez organ wieloosobowych jednostek, które ze względów organizacyjno-technicznych mają trudności z realizacją swoich ustawowych obowiązków. Jednocześnie przez wprowadzenie dobrowolności stosowania nowych rozwiązań projekt nie będzie miał negatywnego wpływu na jednostki, które posiadają wypracowaną i utrwaloną praktykę w zakresie zatwierdzania dokumentów finansowych. Omawiana zmiana przewiduje możliwość podpisania przez jednego z członków zarządu wieloosobowego sprawozdań finansowych oraz z działalności pod warunkiem uzyskania od pozostałych członków zarządu oświadczeń. Ponadto wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych usprawni pracę w zakresie sporządzania wyżej wymienionych sprawozdań i prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ich weryfikacji. Proponowane zmiany w ustawie o biegłych rewidentach związane z postępującą cyfryzacją życia gospodarczego przyczynią się do poprawy komunikacji między Polską Agencją Nadzoru Audytowego a firmami audytorskimi. Biorąc powyższe pod uwagę, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość deklaruję poparcie dla niniejszej ustawy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Zofia Czernow, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1570. Projektowana ustawa służy dostosowaniu obecnie obowiązujących przepisów w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz rewizji finansowej do aktualnej sytuacji prawnej i gospodarczej oraz do nowych możliwości technologicznych.

W projekcie ustawy wprowadza się zmiany w następujących aktach prawnych: ustawie o rachunkowości, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych wywiera istotny wpływ także na rachunkowość i rewizję finansową. Możliwość korzystania z nowoczesnych narzędzi informatycznych sprawia, że jednostki łatwiej mogą wywiązywać się ze swoich obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych.

W sytuacji gdy raport emitenta zawiera skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości, takie sprawozdanie wymaga specjalnego oznakowania. Rozwiązanie to ma na celu zwiększenie przejrzystości, dostępności i porównywalności sprawozdań finansowych sporządzanych przez spółki giełdowe oraz ułatwienie analizy tych sprawozdań. W projekcie wprowadza się także ułatwienia w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych, zwłaszcza dla jednostek kierowanych przez organ wieloosobowy. Odchodzi się od dotychczasowego obowiązku podpisywania sprawozdań przez wszystkich członków wieloosobowego organu na rzecz umożliwienia dokonania tej czynności przez co najmniej jednego członka. Zmiana w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadza możliwość składania do KRS elektronicznych kopii dokumentów - różnego rodzaju oświadczeń - które w oryginale zostały sporządzone w postaci papierowej, a następnie zeskanowane. Liczne zmiany wprowadzane się w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. W sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego biegły rewident wyraża opinię dotyczącą zgodności badanego sprawozdania z wymogami rozporządzenia 2019/815.

Proponowane zmiany wprowadzają do polskiego systemu prawnego regulacje prawa unijnego oraz inne regulacje, dotyczące zwłaszcza biegłych rewidentów, które wymagają zmiany bądź doprecyzowania. Reasumując, klub Koalicji Obywatelskiej rekomenduje skierowanie projektu ustawy do dalszych prac legislacyjnych. Dziękuję za uwagę. Bardzo proszę, pani poseł Anita Sowińska, Lewica. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu parlamentarnego Lewicy wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1570. Cyfrowa transformacja odbywa się w polskich przedsiębiorstwach i organizacjach społecznych już od wielu lat, a przez ostatni rok została przyśpieszona w wyniku pandemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Wiele przedsiębiorstw korzysta z nowoczesnych narzędzi informatycznych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Użytkownicy tych narzędzi mogą w szybki sposób pobierać, analizować i interpretować potrzebne dane. Przedsiębiorcy wdrażają też kolejne rozwiązania polegające na automatyzacji i robotyzacji usług finansowych i raportowania. Unia Europejska dostrzega olbrzymie znaczenie cyfryzacji i sztucznej inteligencji w sektorze finansowym, czemu daje wyraz w strategii Europejskiego Zielonego Ładu oraz w dyrektywach i rozporządzeniach wykonawczych. Jest ważne, aby Polska szybko wdrażała przepisy unijne ze względu na utrzymanie konkurencyjności polskich firm na rynku globalnym, np. w sektorze zewnętrznych usług finansowych. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Polska zajmuje pierwsze miejsce w Europie i trzecie miejsce na świecie, jeżeli chodzi o centra usług wspólnych. W całym kraju działalność prowadzi ponad 1050 centrów, w których jest zatrudnionych ponad 240 tys. pracowników, z czego najwięcej w usługach księgowych i informatycznych. W przedmiocie tej ustawy intencją Unii Europejskiej i rządu jest wprowadzenie przepisów mających na celu ułatwienie dostępności i porównywalności sprawozdań finansowych, tak aby raporty były sporządzane zgodnie z tymi samymi standardami technicznymi. To ma ułatwić nie tylko automatyzację procesów księgowych, ale również kontrolę sprawozdań finansowych. Swoje opinie i uwagi zgłosiły m.in.: Polska Izba Biegłych Rewidentów, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Konfederacja Lewiatan, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Giełda Papierów Wartościowych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich i inne. Ten projekt ustawy to krok w dobrą stronę. Lewica popiera dalsze prace nad tym projektem w Komisji Finansów Publicznych. Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Paszyk, Koalicja Polska. Bardzo dziękuję. Panie i Panowie Posłowie! Ponieważ już ze strony przedmówców dokonano całościowego omówienia projektu, nie będę tego powtarzał, natomiast zadeklaruję ze strony Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści, że tak jak zawsze można było liczyć na nasze wsparcie przy projektach, które usprawniają życie przedsiębiorców, które ułatwiają wszelkie formalności związane z tego typu działalnościami, tak samo w przypadku tego projektu można będzie na nas liczyć. Jesteśmy za tym, aby sprawnie procedować nad tym projektem i uchwalić te zmiany. Dominują właśnie rozwiązania usprawniające, a to, myślę, jest dzisiaj głównym zadaniem władz publicznych, aby takie usprawnienia z myślą o przedsiębiorcach, o biznesie wprowadzać. Dziękuję bardzo. I bardzo proszę, pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050 w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, ujętego w druku nr 1570. Szanowni Państwo! Przedmiotowy projekt ustawy dotyczy sfery cyfryzacji w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych. Z jednej strony wprowadzanie tego typu rozwiązań wymuszane jest przez postęp w dziedzinie cyfryzacji, z drugiej jednak strony dzięki informatyzacji organizacje mogą lepiej wywiązywać się z obowiązków nałożonych przepisami i raportować dane zainteresowanym stronom np. w postaci formatów przeszukiwalnych. Te przepisy, ten projekt wpisuje się właśnie w te postulaty. Myślę, że jedną z najważniejszych zmian w tym projekcie jest ujednolicenie przepisów o rachunkowości w zakresie stosowania jednego formatu elektronicznego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych przez emitentów.

Projektowane przepisy mają na celu wprowadzenie ułatwień dla jednostek kierowanych przez organ wieloosobowy, które ze względów organizacyjno-technicznych mają trudności z realizacją swoich ustawowych obowiązków. To jest bardzo techniczny język, natomiast to rozwiązanie, choć fakultatywne, z pewnością przyczyni się do tego, że te organy wieloosobowe będą łatwiej wypełniały swoje obowiązki.

W naszej ocenie ten projekt ustawy, który pozytywnie wpływa na możliwość wypełniania obowiązków, spełniania wymagań określonych przepisami, zasługuje na wsparcie i dalszą nad nim pracę. W związku z tym w imieniu Koła Parlamentarnego Polska 2050 wnoszę do Wysokiej Izby i pani marszałek o przekazanie projektu do dalszych prac w komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów posłów chce jeszcze zgłosić się do zadania pytania? Jeżeli nie, zamykam listę. Jako pierwsza głos zabierze pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. 1 minuta na zadanie pytania. Panie Ministrze!

To jest oczywiście bardzo istotna i ciekawa inicjatywa i chciałem od pana ministra usłyszeć informację, czy to będzie wiązało się z poniesieniem dodatkowych kosztów na te elementy cyfryzacyjne, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Proponowane zmiany zapisane w projekcie należy uznać za celowe. Mam jednak pytanie do pana ministra, które zadają też moi wyborcy. Dlaczego w Polsce istnieją instytucje obracające miliardami złotych, które albo nie prowadzą wcale sprawozdawczości, albo unikają publikacji wyników skonsolidowanych, co w praktyce uniemożliwia zapoznanie się z prawdziwymi danymi finansowymi tych jednostek? Dziękuję bardzo. Pani Zofia Czernow, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Z uwagą przeczytałam wyniki konsultacji społecznych i zaniepokoiło mnie stanowisko ministerstwa w sprawie uwagi wniesionej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Otóż Urząd Ochrony Danych Osobowych zauważa, że w ustawie jest zapis, który mówi, że sprawozdania finansowe podlegają przechowywaniu przez okres co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następnego itd.

Powinien być wskazany konkretny czas, jak długo przechowywane są sprawozdania finansowe. Wynika to z RODO, z zasady ograniczonego przechowywania, kiedy to przechowywanie nie jest potrzebne. Dlaczego ministerstwo nie chce zmienić tego przepisu? Dziękuję. Bardzo proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów pana ministra Piotra Patkowskiego o udzielenie odpowiedzi. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Odpowiadając najpierw na pytanie pana posła Suchonia, chciałbym wskazać, że ten projekt wręcz ogranicza koszty ponoszone przez budżet państwa, czyli należy do kategorii projektów najbardziej lubianych przez ministra finansów. Dokładnie o ile ogranicza, wskazuje pkt 6 w OSR i w pierwszym pełnym roku obowiązywania projektu będzie ponad 600 tys. zł oszczędności. Ta kwota będzie rosła do 700 tys., czyli w przeciągu 7 lat oszczędzimy na tym projekcie prawie 7 mln zł.

Szacujemy, że zmniejszenie wydatków o ok. 630 tys. zł rocznie wynika m.in. z tego, że agencja będzie prowadziła ok. 300 kontroli, w tym 250 kontroli planowanych i 50 kontroli doraźnych i tych tematycznych. Agencja zakłada, że 70% tych kontroli, czyli 210, będzie prowadzonych zdalnie, w związku z czym koszty będą niższe. Natomiast chciałbym tylko podkreślić, że każdy podmiot obowiązany do prowadzenia sprawozdań finansowych musi je złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej. Ten katalog podmiotowy jest bardzo ściśle określony, m.in. kryteriami kwotowymi.

Uwaga UODO dotyczyła tego, czemu to nie jest okres maksymalny. Odpowiedź jest taka i też podnosiliśmy to w konsultacjach, że nie możemy zakazać jednostkom trzymania danych analitycznych więcej niż 5 lat, m.in. dlatego, że, po pierwsze, to jest ich decyzja, po drugie, nie mając takich informacji, jednostki nie mogłyby przeprowadzać analiz czy być przygotowane na ewentualne toczące się sprawy sądowe. Tak że zapewniamy pewną dowolność podmiotom, natomiast to nie może w żaden sposób uchybiać innym przepisom UODO. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw zawarty w druku nr 1570 do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Ogłaszam 15 minut przerwy.

Proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury pana ministra Rafała Webera o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Polska jest dzisiaj bezpiecznym krajem, ale wciąż jest jeden wyjątek. To bezpieczeństwo na drogach. Nasze drogi są znaczone krzyżami, które oznaczają śmiertelne wypadki drogowe i tragedie tysięcy rodzin. Tymi słowami wygłoszonymi na tej sali, na tej mównicy podczas exposé pan premier Mateusz Morawiecki wskazał na problem, którego rozwiązanie w obecnej kadencji jest jednym z ważniejszych celów rządu i parlamentu. Znaczna poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym to nasz priorytet, a nawet szerzej - to zadanie, które stoi przed całą klasą polityczną. Polska od lat - można powiedzieć, że od dekad - jest na szarym końcu państw w Europie, jeżeli chodzi o liczbę wypadków i ofiar wypadków drogowych. Pomimo tego, że co roku w tym obszarze statystycznie mamy do czynienia ze spadkiem, to ten spadek jest za mało widoczny, za mało dynamiczny, a redukcja wypadków, ofiar i rannych wielce niewystarczająca. Tak jak w 2010 r. Polska była na 4. miejscu od końca wśród państw Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, tak i dziś, po ponad 10 latach, jesteśmy w tym samym miejscu, nadal w ogonie Unii Europejskiej. To musi się zmienić. Musimy podjąć takie kroki i takie działania, które doprowadzą do wyraźnej poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tego oczekują - można powiedzieć wręcz, że tego żądają - od nas kierowcy, pasażerowie, rowerzyści, piesi, tego oczekują od nas wszyscy ci, którzy na co dzień korzystają z polskiej infrastruktury drogowej, niezależnie od tego, czy to drogi krajowe, czy drogi zarządzane przez samorządowców.

Pierwsza to inwestycje drogowe. Druga to edukacja i wzmacnianie świadomości wszystkich uczestników ruchu drogowego. Trzecia sfera to zmiany w przepisach prawa. Dziś przedstawiam Wysokiej Izbie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zawarty w druku nr 1504. Proponowane zmiany mają zlikwidować dwie patologie, z którymi mamy do czynienia na polskich drogach. Pierwsza to piractwo - można powiedzieć, że bandyctwo - drogowe. Druga to pijani za kierownicą. Te dwie zmory muszą zostać wyeliminowane z drogowej rzeczywistości. Podnosząc stawki mandatowe piratom i pijanym za kółkiem, pokazujemy, że nie będziemy tego więcej tolerować, nie będziemy pobłażać tym, którzy radykalnie przekraczają dopuszczalną prędkość, a także tym, którzy siadają za kółkiem pod wpływem alkoholu. Tacy kierowcy są postrachem. Każdego dnia słyszymy o ludzkich tragediach, o zabranych życiach, o rozbitych rodzinach właśnie dlatego, że ktoś jechał za szybko, a inny znów jechał pijany. Musimy z tym skończyć.

Oczywiście w uzasadnionych przypadkach będzie można zastosować karę aresztu i o tym będzie decydował sąd.

W naszym zamierzeniu wzrost maksymalnej wysokości grzywny wystawionej w postępowaniu mandatowym do 5 tys. zł oraz do 30 tys. zł w postępowaniu sądowym jest jasnym sygnałem, że dla najcięższych wykroczeń drogowych nie będzie litości, nie będzie zmiłuj. Podkreślam słowo „najcięższych”, czyli takich, które w sposób bezpośredni zagrażają zdrowiu lub życiu. Tymi stawkami nie będą objęci ci, którzy popełniają drobne wykroczenia, np. niewłaściwe parkowanie. Mówię to, bowiem w ostatnich tygodniach, od momentu pokazania tego projektu ustawy, pojawiają się w przestrzeni medialnej różnego typu manipulacje, przekłamania i - można powiedzieć to językiem, który jest bardzo popularny w polityce - fake newsy.

Drobne wykroczenia nie będą podlegały zmianie przepisów tej ustawy. W dalszej kolejności wzmacniamy ochronę pieszych na przejściach dla pieszych poprzez zwiększenie minimalnej kary za nieprawidłowe zachowanie względem pieszego. Dane statystyczne jasno pokazują, że blisko 90% wypadków na przejściach dla pieszych powodują kierowcy. Stąd nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie lub omijanie innych pojazdów na przejściu dla pieszych będzie karane surowiej, bo mandatem minimum 1500 zł, a w przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego sąd będzie mógł orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Z innych kwestii projekt zakłada podniesienie stawki minimalnej także za: jazdę bez uprawnień, za objeżdżanie opuszczonych zapór i niedozwolone przyjeżdżanie na przejazd kolejowy, za utrudnianie lub tamowanie ruchu, za łamanie zakazu wyprzedzania, za niestosowanie się do sygnałów dźwiękowych. Poza podniesieniem punktowym, podniesieniem minimalnych mandatów proponujemy jeszcze zmiany w systemie naliczania punktów karnych. Punkty będą anulowane po 2 latach od ich otrzymania, ale pod warunkiem opłaty mandatu za dane wykroczenie drogowe. Podnosimy także do 15 pkt maksymalny wymiar za najgroźniejsze wykroczenia. Inne ważne zmiany dotyczą sfery ułatwiania możliwości otrzymania renty przez bliskich ofiar wypadków drogowych. Rodziny ofiar wypadków drogowych - chodzi o traumę, szok - nie radzą sobie z całą prawną procedurą uzyskania renty. Będą mogły otrzymać od struktur państwa wsparcie. Nie możemy takich osób w tak trudnych sytuacjach pozostawiać samych sobie. Dlatego projekt przewiduje uproszczenie postępowania w sprawie renty, która będzie wypłacana przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym osobom najbliższym dla ofiary wypadku drogowego, mającej na utrzymaniu osoby, które w efekcie straciły żywiciela. Świadczenie to będzie zwolnione od podatku dochodowego i niewliczane jako dochód przy obliczaniu świadczeń rodzinnych. Kolejną istotną propozycją jest uzależnienie wysokości składki ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych od liczby punktów karnych i historii popełnianych najcięższych wykroczeń. Projekt ustawy przewiduje udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i umożliwi dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. Po zakończeniu oceny ryzyka zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek niezwłocznie usunąć dane o punktach karnych kierowcy. Mamy nadzieję, że ten przepis pozwoli w odpowiedni sposób nagradzać, preferować tych, którzy jeżdżą bezpiecznie, tych, którzy nie łamią najpoważniejszych zasad ruchu drogowego. Oni będą płacili niższe składki OC, a ci, którzy dopuszczają się w ruchu drogowym łamania przepisów ruchu drogowego - cały czas mówię tylko i wyłącznie o najcięższych wykroczeniach, które są określone w tym projekcie ustawy - będą siłą rzeczy zobowiązani do opłaty wyższej składki ubezpieczeniowej. Proponujemy więc cały pakiet zmian prawnych. Jestem przekonany, że w pozytywny sposób wpłyną one na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zależy nam na tym, aby uratować, ocalić jak najwięcej żyć, ale też zależy nam na zmniejszeniu kosztów finansowych wypadków drogowych, które są liczone w dziesiątkach miliardów złotych rocznie. W roku 2019 to rekordowe 56 mld zł, a więc im mniej wypadków, im mniej ofiar, tym mniejsze koszty dla nas wszystkich. Trudno mi przeliczać życie na pieniądze. Używam tego argumentu, aby pokazać, że w tej dyskusji również i ten kontekst ma miejsce, i ten kontekst jest ważny, i na ten kontekst w różnego rodzaju dyskusjach, choćby w dyskusji o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w poszczególnych latach, państwo parlamentarzyści zwracają uwagę. Konkluzja mojego wystąpienia: celem zmian jest wyeliminowanie pijanych za kierownicą. Dość powiedzieć, że tylko wczoraj policja zatrzymała blisko 200 nietrzeźwych, natomiast w skali roku takich zatrzymań jest nawet ponad 100 tys. W roku 2019 ponad 100 tys. pijanych kierowców zostało zatrzymanych przez policję. Ilu nie zostało zatrzymanych, bo im się udało? Zostawiam to pytanie otwarte, zostawiam znak zapytania, ale myślę, że każdy zdaje sobie sprawę, że takich osób było więcej. Tak że musimy z tą patologią skończyć. Musimy także ujarzmić piratów drogowych, spowodować, aby dopuszczalna prędkość zarówno w obszarze zabudowanym, jak i poza nim była przestrzegana. W tym przypadku szacunek dla prawa równa się szacunkowi dla życia. Mocniej chcemy karać tych, którzy za nic mają innych i w sposób celowy, bardzo często systematyczny, łamiąc przepisy prawa, zagrażają innym. Szanowni Państwo! Z niecierpliwością czekam na wystąpienia klubowe, z niecierpliwością czekam również na indywidualne oceny pań i panów posłów dotyczące tego projektu ustawy. Śledzę media, które opisują ten projekt ustawy w ostatnim czasie. Śledzę również wypowiedzi tych, którzy się tym tematem interesują. Jestem przekonany, że na i tej sali, i zapewne na posiedzeniu Komisji Infrastruktury dyskusja będzie bardzo energiczna, żywa, ale mam nadzieję, że będzie bez emocji, i mam nadzieję, że będzie merytoryczna. Chcę powiedzieć, że nie zamykam się na argumenty, nie zamykam się na propozycje. Być może ten projekt będzie jeszcze ulegał zmianom, zapewne będą składane do niego poprawki.

Natomiast mając doświadczenie zarówno z tej, jak i z poprzedniej kadencji, obawiam się że będą takie propozycje, które będą nawzajem się wykluczały. Jedna strona będzie chciała karać jeszcze bardziej, druga strona będzie chciała, aby kar w ogóle nie było albo aby były mnie dotkliwe.

Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1504. Rozpatrywany projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ma dwa zasadnicze cele: po pierwsze, wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, po drugie, poprawę bezpieczeństwa na drogach, w szczególności przez walkę z przestępstwami drogowymi. Aby wzmocnić funkcję prewencyjną i sprawiedliwościową prawa, zdecydowano się na wprowadzenie szeregu zmian, które pozwolą na skuteczniejszą walkę z niebezpiecznymi kierowcami na drodze. Proponowane regulacje wynikają zarówno z odpowiedzi na szeroki problem społeczny o wysokiej szkodliwości społecznej, jak i z potrzeby uspójnienia regulacji prawnych, w szczególności przez zerwanie z uprzywilejowaną pozycją sprawców przestępstw drogowych. W związku z tym w projekcie przewiduje się zaostrzenie kar dla sprawców wykroczeń drogowych. W projekcie zakłada się również oddziaływanie innymi środkami niż środki karne i proponuje się powiązanie wysokości opłat z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą uzyskanych punktów karnych i historią popełnionych wykroczeń. Proponuje się wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK oraz dostosowanie taryfikacji do historii i wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. Dostosowanie wysokości składek do historii wykroczeń kierowcy pozytywnie wpłynie na wysokość składki w przypadku kierowców, którzy jeżdżą zgodnie z przepisami. Będzie to niewątpliwie pozytywne wzmocnienie. Różnicowanie wysokości ubezpieczenia motywuje finansowo kierowców do bezpiecznej jazdy. Bezpieczna jazda jest premiowana brakiem konieczności poniesienia dodatkowych kosztów umowy ubezpieczenia. Za umowę ubezpieczenia płaci każdy kierowca, a za mandat płaci tylko ten, który dopuści się wykroczenia.

Daje to wskaźnik ok. 11 osób zabitych i 112 osób rannych na 100 wypadków. Wynika z tego, że w co dziesiątym wypadku zginął co najmniej jeden człowiek. Co istotne, zgodnie z danymi niemal 90% z nich wydarzyło się z winy kierujących. Zginęło w nich 216 osób, a rannych zostało 1847 osób. Wysoki Sejmie! Z dużą satysfakcją należy przyjąć, że w tym projekcie przewiduje się również uproszczenie postępowania w sprawie renty, która będzie wypłacana przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym osobom najbliższym ofiary wypadku drogowego mającej na swoim utrzymaniu osoby, które w efekcie straciły członka rodziny. Świadczenie to będzie zwolnione od podatku dochodowego i nie będzie wliczane jako dochód przy obliczaniu świadczeń rodzinnych. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość zamierza w toku dalszych prac parlamentarnych wspierać ten projekt. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Maciej Lasek, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ustawa zwiększająca wysokość kar za wykroczenia drogowe na pewno wzbudzi wiele emocji, ale niestety jest to przykra konieczność.

Jednocześnie w 2019 r. na drogach w Polsce zginęło prawie 3 tys. osób, a 34 tys. zostało rannych. Znajdujemy się pod tym względem w niechlubnej czołówce Europy razem z takimi państwami jak Bułgaria czy Rumunia. Ryzyko śmierci na drodze w wyniku wypadku jest w Polsce cztery razy większe niż w Norwegii czy Szwajcarii. Są nimi dobra infrastruktura, właściwy system szkoleń, przemyślane przepisy i nieuchronność kary. Raport o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym obejmujący okres do 2019 r. włącznie wskazuje, że większość trendów opisujących poprawę bezpieczeństwa uległo zahamowaniu.

Omawiana ustawa zdaje się kontynuować ten dobry kierunek zmian, jednak w aktualnej formie jest ona daleka od ideału i budzi wiele poważnych zastrzeżeń.

Zmiana ta jest całkowicie nieuzasadniona, na co wskazuje w obszernym stanowisku rzecznik praw obywatelskich. Obywatel musi z góry wiedzieć, czy jego czyn wypełnia znamiona wykroczenia i jakie za nie poniesie karę. Ta nowelizacja otwiera zaś drogę do karania nie tylko za poważne wykroczenia drogowe, z czym się wszyscy zgadzamy, ale również za czyny, które mają znacznie mniejszą społeczną szkodliwość. Takim przykładem może być proponowane w ustawie podwyższenie do 5 tys. zł kary za tamowanie ruchu. Czy obejmować to będzie również karanie przez policję wielotysięcznymi mandatami spontanicznie protestujących osób? Przecież to jest otwarta droga do naruszenia swobód obywatelskich. Myślę, że to powinniśmy w toku prac wyjaśnić. Według wnioskodawców drastyczne podwyższenie kar za wykroczenia ma budować prewencję i odstraszać. Ale to nie wysokość sankcji, tylko jej nieuchronność buduje prewencję. Ustalenie wysokości kar w całkowitym oderwaniu od średnich zarobków na głowę spowoduje, że będą one nieegzekwowalne. Według obecnych przepisów, gdy niemożliwa jest egzekucja, grzywnę można zamienić na ograniczenie wolności lub areszt do 30 dni. Może się okazać, że kary na poziomie 10, 15 czy 30 tys. zł będą nieściągalne, bo ukarani nie będą w stanie ich zapłacić, co będzie skutkowało ich zamianą na areszt. Jakie koszty poniesie w ten sposób budżet państwa, o kosztach społecznych nie wspominając? Kiedy rozmawiamy o zasadności wysokości mandatów, zastanówmy się też, jak to rzutuje na procedurę wystawiania mandatów. Wątpliwości zgłasza również rzecznik praw obywatelskich. Policjant w ciągu kilku minut bez żadnego głębszego rozeznania w możliwościach zarobkowych sprawcy i jego sytuacji osobistej może wystawić mandat nawet w wysokości 6 tys. zł. Ba, może go przyjąć w gotówce, co stwarza realne zagrożenie korupcją przy takiej dysproporcji w stosunku do zarobków. Według projektu wpływy z kar mają zasilić Krajowy Fundusz Drogowy z przeznaczeniem na budowę i remonty dróg krajowych oraz poprawę ich bezpieczeństwa. Ustawodawca jednak w żaden sposób nie definiuje, co rozumie przez poprawę bezpieczeństwa, i nie pochyla się też nad kwestią proporcji podziału tych środków. Wątpliwości budzi również to, że pieniądze mają iść tylko na drogi krajowe. Kompletnie pomija się drogi gminne, na których przecież w równym stopniu dochodzi do wykroczeń drogowych i które tak samo potrzebują środków na remonty i infrastrukturę bezpieczeństwa. W świetle postulatów wsparcia poszkodowanych w wyniku wypadków uzasadnionym jest postulowanie, aby część pieniędzy została przeznaczona na dedykowany ofiarom wypadkom fundusz, który mógłby zapewnić niezbędną im do życia i powrotu do zdrowia pomoc finansową, zwłaszcza że ofiary nieumyślnych przestępstw drogowych nie mają swojego funduszu pomocy.

Jednakże procedura dotyczy tylko przestępstw umyślnych, a w toku orzecznictwa i praktyki przyjęto, że wypadki drogowe to w większości przestępstwa nieumyślne. Dodatkowo, jeżeli mówimy o postępowaniu o przyznanie renty, to ma ono kilka mankamentów. Co w sytuacji, gdy ofiara wypadku jest w jego wyniku trwale niezdolna do pracy? Dziękuję bardzo. Dlaczego ci, którzy przeżyli, mają być skazani na udowadnianie swojej szkody i niezdolności do pracy w długotrwałych procesach cywilnych? Po drugie, to, co wydaje się być największą zaletą projektu, czyli wszczynanie postępowania wraz z odpisem prawomocnego wyroku, wydatnie może opóźnić jego rozpoczęcie. Przecież takie sprawy z apelacją mogą trwać nawet 2 lata. W rygorze zwykłym poszkodowani mogą zwracać się o wypłatę renty już na poziomie postępowania likwidacyjnego. Wierzę, że w toku rzetelnej i ponadpartyjnej pracy w komisjach, nie pomijając przy tym zdania instytucji prawniczych, organizacji społecznych i wysłuchania publicznego, stworzymy akt prawny oddający sprawiedliwość wszystkim poszkodowanym, który sprosta oczekiwaniom społecznym i pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pani poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Lewica. Wysoka Izbo! Powiedzmy sobie wprost: na polskich drogach i ulicach od lat trwa po prostu krwawa rzeź. W ich konsekwencji śmierć poniosło niemal 2,5 tys. osób, a ponad 26 tys. odniosło rany, nierzadko wymagające wieloletniej i kosztownej rehabilitacji. To są konkretne, dramatyczne liczby, ale przecież największych krzywd związanych z tragediami na polskich drogach nie da się zmierzyć. Nie policzy się bólu i cierpienia po stracie ukochanej babci, ojca, dziecka, brata czy siostry. Gdyby dowolny rząd, niezależnie od tego, która partia była u władzy, wcześniej pochylił się nad zmianami legislacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, szeregu tragedii udałoby się uniknąć. Wiele rodzin mogłoby się nadal cieszyć z obecności ukochanej osoby. Oprócz tej najcenniejszej wartości, jaką jest ludzkie życie i zdrowie, wypadki drogowe kosztują budżet państwa konkretne, ogromne pieniądze. W skali rocznej to ok. 56 mld zł. Poprawiając sytuację na drogach, możemy wiele jako społeczeństwo zaoszczędzić, a pozyskane w ten sposób pieniądze przeznaczyć np. na podwyżki dla przedstawicieli zawodów medycznych, nauczycieli, pracowników służby cywilnej, sądów czy prokuratur. Polki i Polacy mają dość bandyterki na drogach. 82% polskiego społeczeństwa popiera wprowadzenie surowszych kar za przekraczanie prędkości. Aktywiści i społecznicy słusznie zwracają uwagę, że maksymalna stawka mandatu, która wynosi niezmiennie od prawie 25 lat zaledwie 500 zł, przestała już kogokolwiek odstraszać. Przestępcy drogowi przestali mieć jakikolwiek respekt dla prawa i polskiego państwa. Dlatego jako Lewica aprobujemy główny kierunek zmian zaproponowany w projekcie ustawy, czyli zwiększenie kar dla łamiących przepisy na drogach, podniesienie wysokości kwoty mandatów, wprowadzenie renty dla bliskich zmarłego czy powiązanie stawek ubezpieczenia OC z bezpieczną jazdą. Ale projekt ten niestety budzi także nasze poważne wątpliwości. Bardzo niepokojąca jest chociażby kwestia podniesiona przez rzecznika praw obywatelskich. Radykalne zaostrzenie kar ma bowiem dotyczyć również art. 90 kodeksu wykroczeń, który dotyczy tamowania ruchu. Co to oznacza w praktyce? Czy rząd za pośrednictwem tej nowelizacji chce sobie zapewnić instrument do zniechęcania ludzi do korzystania ze swojego konstytucyjnego prawa do pokojowych zgromadzeń, narzędzie ograniczające prawo do strajku, spontanicznego protestu czy pikiety? Szczerze chciałabym wierzyć, że nie, że to jest po prostu błąd i niedopatrzenie, ale ponieważ prawa nie stanowi się na wiarę, dlatego Lewica złoży odpowiednie poprawki w tym zakresie. Projekt ustawy wprowadza także chaos w przypadku drogowej recydywy. Dobór wykroczeń, które będą skutkować surowszą sankcją w przypadku ponownego popełnienia czynu karalnego w przeciągu 2 lat wygląda jak loteria. Dla przykładu, jeśli wcześniej wystawiono komuś mandat za tamowanie ruchu, a następnie ta sama osoba zostanie przyłapana na niewłaściwym parkowaniu, zostanie ukarana grzywną o wartości minimum 3 tys. zł. Z drugiej strony zaś, jeśli dwukrotnie popełni wykroczenie w postaci prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu do 0,5 promila, za recydywistę uznana nie zostanie. W tym zakresie także zgłosimy poprawki, które uporządkują system karania w warunkach powrotu do wykroczenia. W projekcie nowelizacji zabrakło również wielu innych bardzo istotnych zmian. Wciąż czekamy na możliwość czasowego zatrzymania samochodu osobom jeżdżącym wbrew zakazowi. Nie wiadomo, czy Ministerstwo Sprawiedliwości spełni swoje obietnice dotyczące konfiskaty aut za najcięższe przestępstwa drogowe. Projekt ustawy nie zawiera także realizacji postulatu nieuchronności kary przez zmianę egzekucji mandatów na uproszczone postępowanie administracyjne. Cały czas czekamy także na zwiększenie liczby fotoradarów, przywrócenie możliwości ich stawiania przez samorządy, ustanowienie policji autostradowej, wprowadzenie odcinkowych pomiarów kontroli prędkości na autostradach i drogach szybkiego ruchu, na których dziś panuje po prostu wolna amerykanka. Jako Lewica będziemy popierać wszelkie zmiany zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, ale nie pozwolimy, żeby stały się one wytrychem do ograniczania konstytucyjnych praw obywateli. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Stefan Krajewski, Koalicja Polska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Oczywiście nie robicie tego. Drugi z przedstawionych celów projektu to jeden z najbardziej palących problemów społecznych w Polsce. Zgodnie z danymi statystycznymi przygotowanymi przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w 2020 r. zgłoszono 23 540 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub w strefach ruchu, w wyniku których 2491 osób poniosło śmierć, a ranne zostały 26 463 osoby, w tym ciężko ranne - 8805.

Nie mają gdzie zjechać, odpocząć, wypić kawy.

Wiele MOP-ów dzisiaj jest zamkniętych.

Wy oczywiście potraficie tylko karać.

Kierowca, który jeździ zawodowo za najniższe stawki, który zarabia najniższą krajową i będzie musiał zapłacić taki mandat, będzie płacił i będzie płakał. Was to nie interesuje.

Nikt się nie zastanawia nad, co dana poprawka wnosi, czy ona jest potrzebna, czy nie. Nie wierzę, że treść tej ustawy ulegnie zmianie, dlatego na ręce pani marszałek składam wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Dobromir Sośnierz, Konfederacja.

Pan minister powiedział, że powinno podejmować się w takich sprawach decyzje na chłodno i bez emocji, a tymczasem po raz kolejny uchwalamy ustawę po to, żeby skonsumować oburzenie społeczne po jakimś głośnym wypadku, prawda? Mediokracja w praktyce. Jak rząd potrzebuje jakiegoś sukcesu, to idzie na wojnę, oczywiście nie z jakimś tam potężnym, groźnym przeciwnikiem, bo w takich przypadkach nasz rząd zwykle dostaje lanie, ale na wojnę z własnymi kierowcami, bo to najłatwiej. Na kierowców od lat zrzuca się wszystkie winy, przypisuje się im skutki zaniedbań rządu, wychowuje się w ciągłym poczuciu winy i każe nawet wbrew prawom fizyki ustępować wszystkim i wszystkiemu, zwłaszcza rowerzystom wpadającym znienacka na przejście dla rowerów. To jest właśnie wojna na miarę waszych możliwości, w dodatku skazana na sukces, bo liczba wypadków od lat systematycznie spada, więc za rok powiecie, że tym razem to wasza zasługa, a jak akurat nie zmaleje, to odczekacie rok i ogłosicie sukces za 2 lata. Nie potraficie walczyć z kradzieżami, nie potraficie wyłapać imigrantów na granicy, nie potraficie obronić się przed Unią Europejską, więc będziecie po prostu kroić na kasę bezbronnych obywateli za karę, że jadą samochodem i nikogo nie krzywdzą, bo te drakońskie kary są przewidziane przede wszystkim za przestępstwa bez poszkodowanych, np. za to, że jakiś hipokryta za biurkiem uznał, że on wie lepiej, jak szybko można jechać w danym miejscu. I tylko dlatego, że ten idiota za biurkiem postawił jakiś głupi znak, którego i tak nikt nie przestrzega, karany będzie jakiś pechowy kierowca jadący zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Tylko ofiara losu jeździ po mieście pięćdziesiątką. Miliony ludzi jeżdżą normalnie i większość z nich nigdy nie powoduje żadnego wypadku. Po prostu jakiś nieszczęśnik od czasu do czasu zapłaci taki podatek od pecha, bo tym są właśnie te mandaty. To jest podatek od pecha, podatek od normalnej jazdy. A wy chcecie zasadzać się na normalnych ludzi jak zbóje przy moście i ściągać haracz, chociaż sami jeździcie przecież tak samo. Brzydzę się hipokrytami od lewa do prawa, którzy to popierają. Za kradzież poniżej 500 zł grozi w tym kraju łagodniejsza kara niż za przekroczenie prędkości albo jazdę bez świateł w dzień, bo państwo wolicie wysyłać policję do krojenia kierowców zamiast do uganiania się za prawdziwymi przestępcami. Ci sami ludzie, którzy wielokrotnie twierdzili, że kara śmierci nie działa, bo nie liczy się surowość, tylko nieuchronność i resocjalizacja, tutaj ścigają się na penalny populizm z rządem. Za nieostrożną jazdę grozi już teraz kara śmierci wymierzana na miejscu siłami natury. Jeśli kogoś, jakiegoś wariata ta kara śmierci nie odstrasza, to dlaczego miałyby go odstraszyć mandaty i grzywny. One po prostu spadną nie na piratów, tylko na normalnych ludzi jadących do pracy. Na jakiej więc podstawie stwierdzacie, że to nie działa? Jeśli chodzi o porównanie tempa przyrostu liczby pojazdów z tempem spadku liczby wypadków, to jesteśmy jednym z liderów w Europie, tylko zawsze wybieramy (Dzwonek) sobie wskaźnik, w którym wypadamy źle, i na tej podstawie chcemy niszczyć ludziom życie. Konfederacja składa wniosek o odrzucenie tego gówna w całości.

Panie Ministrze! By skutecznie chronić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, szczególnie tych najsłabszych, potrzebny jest cały system, nie tylko jednostkowe rozwiązania.

To działa. Kara powinna być jednak adekwatna, nieuchronna i jak najbardziej zbliżona w czasie do popełnianego czynu. Omawiany projekt nie zapewnia niestety żadnej z tych cech, ale zasadniczo jest dobry co do kierunku, bo limit mandatu nie zmienił się od 24 lat, choć przeciętna pensja wzrosła ośmiokrotnie. Gdyby rozsądnie powiązać wysokość kar ze średnim wynagrodzeniem, może dziś nie mielibyśmy kłopotu. To rozwiązanie będziemy zresztą postulować. Ale rząd proponuje wzrost tak absurdalny, że protestuje nawet rzecznik praw obywatelskich. Na grzywnę będzie stać zamożnych, a ubożsi zapełnią areszty. O skuteczności systemu decyduje nie tylko współmierność, ale też nieuchronność kary, a tu zamiast skutecznej egzekucji, z czym w Polsce jest wieczny problem, urządzacie ludziom swoistą grę w Monopoly, której reguły wyznacza rzut kostką przynoszący raz ruinę, a innym razem wysyłający do pola: więzienie.

Dodatkowo projekt jest pułapką dla uczestników ulicznych protestów i czujemy się nieco urażeni, panie ministrze, że myśleli państwo, że się w tym nie zorientujmy. Czy osoba, która podczas protestu zostanie zepchnięta przez tłum z chodnika na jezdnię, ma zapłacić 30 tys. zł kary tak jak pijany kierowca? Mówi pan, panie ministrze, o budzeniu respektu i odstraszaniu. I zgoda: zero tolerancji dla drogowych zabójców gnających 200 czy 300 km przez miasto po kilku głębszych. Natomiast kara musi mieć przede wszystkim wymiar wychowawczy, korygujący zachowanie. O tym zupełnie, wydaje się, zapomnieliście, bo kiedy nawet za najmniejszy błąd grozi niewspółmiernie wysoka kara, a w dodatku rzadko nakładana i egzekwowana, to taki przepis niestety pozostaje martwy. Jako Koło Parlamentarne Polska 2050 złożymy poprawki i deklarujemy chęć pracowania nad tym projektem w dobrym kierunku. Mamy nadzieję na rzeczywistą współpracę, tak by ten projekt naprawdę służył życiu i bezpieczeństwu. Decyzję oczywiście uzależnimy od ich przyjęcia. Dziękuję bardzo, pani poseł. Zamykam listę. Jako pierwsza pytanie zadaje pani poseł Iwona Maria Kozłowska, Koalicja Obywatelska.

Panie Ministrze! Poprawa bezpieczeństwa na drogach, a szczególnie walka z przestępcami drogowymi, to temat od lat analizowany i zawsze aktualny. Codziennie słyszymy o wypadkach i tragediach na drogach.

Wolicie więc karać niż przeciwdziałać. Ale mam pytanie odnośnie do tego projektu: Na jakiej podstawie i według jakiego algorytmu zostały ustalone stawki i kary? Czy nie warto zastanowić się jednak nad waloryzacją grzywien, np. co 3 lata lub 5 lat? Dałoby to większą szansę na to, aby przeanalizować, czy rzeczywiście wysokość nałożonych kar daje jakąkolwiek poprawę bezpieczeństwa pojazdów na drogach i osób korzystających z dróg publicznych? Bardzo proszę, pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Mam wrażenie, że w państwa podejściu do polityki karnej jedyne, co widzicie, to zasada represji. Coraz surowsze kary, coraz wyższe mandaty. To jest teoria odpłaty w pełnej krasie, jak 100 lat temu. O tym, że kara powinna mieć też walor wychowawczy, mam wrażenie, wszyscy państwo zapomnieli. A już Monteskiusz nie miał wątpliwości, że drakońskie zaostrzanie kar jest symptomatyczne dla państwa oddalającego się od wolności. No i w tym dokumencie to również widać. Sprawiedliwościową funkcję prawa karnego uzależniacie państwo od stopnia zamożności. Przecież to absurd. Pytam pana jak prawnik prawnika: Gdzie jest walor wychowawczy tych drakońskich kar? Tylko bez populizmu, bo wszyscy na tej sali wiemy, że szaleni kierowcy niosą śmierć, że pijani kierowcy są zbrodniarzami. Tylko co państwo robi obecnie, aby skutecznie egzekwować nakładane (Dzwonek) kary? Skąd przekonanie, że sprawniej pójdzie egzekwowanie wyższych kar, skoro dziś nie radzicie sobie z niższymi? I ostatnie, choć też dosyć istotne pytanie, panie ministrze: Kiedy pan widział uprzywilejowany pojazd wiozący ministra, sekretarza stanu, który jechałby zgodnie z przepisami? Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Jan Szopiński, Lewica.

Jest jednak taki moment, że kara przestaje odstraszać, a zaczyna budzić śmieszność. Panie Ministrze! Proszę nie patrzeć na średnią dochodów podbijaną przez wasze rodziny, krewnych, czy znajomych, tłuste koty ze spółek Skarbu Państwa. Proszę spojrzeć na zwykłego Polaka niepowiązanego z PiS-em. Większość z nich żyje za minimalne wynagrodzenie krajowe, a emeryci - często za połowę tej kwoty, natomiast mandaty po 3 tys., 5 tys. czy 6 tys. czy nawet po 30 tys., jak zwraca uwagę rzecznik praw obywatelskich, są śmieszne i niedorzeczne. A więc mam pytanie do pana: Kiedy pan chce dokonać konsultacji tego projektu i z kim? Z kim pan chce dokonać wysłuchania publicznego?

Polacy! Dziękuję bardzo. Pan poseł Ryszard Wilczyński, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Karać, karać - to potraficie, ale znajdować rozwiązania - nie. Trzy razy na tej mównicy mówiłem, jeszcze w poprzedniej kadencji: zrobić oznakowanie poziome na obszarach, gdzie często jest mgła. Mówiłem to jako człowiek, który widział na własne oczy śmierć dwóch ludzi we mgle. Minister Adamczyk mówił: oczywiście, zrobimy. Zrobiliście? Wiecie, jak wygląda oznakowanie poziome do jazdy we mgle na autostradach? Nie, bo może nie jeździcie za granicę. Wie pan, ile wynosi prędkość dopuszczalna w obszarze zabudowanym w Austrii na zmodernizowanej drodze landowej? No pewnie pan nie wie, bo pan nie jeździ.

A więc racjonalnie podnosić kary, ale też zmieniać przepisy, zmieniać oznakowania, dostosowywać to do realiów modernizacji. Ludzie przekraczają prędkość głównie dlatego, że nie są w stanie dojechać nigdzie w rozsądnym czasie.

Pan poseł Ryszard Galla, poseł niezrzeszony. Panie Ministrze! Na pewno naszym celem jest dbanie o to, aby wyeliminować pijanych kierowców, piratów drogowych, walczyć z wszelką patologią, która występuje na jezdni. Pytanie: Czy to wszystko osiągniemy właśnie polityką wzrostu cen mandatów? Tutaj już przedmówcy mówili o tym, że rzecznik praw obywatelskich bardzo mocno skrytykował poziom tych kwot, wskazując też, powiedziałbym, pewnego rodzaju patologię.

Pan poseł Lasek wymienił kilka elementów, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym: infrastruktura, kultura kierowców, ale też i prawo. Nie wiem, czy pan (Dzwonek) w ogóle śledzi korespondencję, ale wielokrotnie pisząc do państwa, wskazywałem na pewne niedociągnięcia, wręcz powiedziałbym: nielogiczne sytuacje, jeśli chodzi o polskie prawo w ruchu drogowym. Czy rzeczywiście podejmiecie też prace nad tym, żeby to prawo tak dostosować, aby ono naprawdę było bardzo, bardzo racjonalne? Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zacytuję informacje ze strony internetowej kancelarii adwokackiej, która pomaga odzyskać zatrzymane prawa jazdy: Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że postępowanie karne za jazdę po alkoholu może zakończyć się warunkowym umorzeniem. Warunkowe umorzenie postępowania jest korzystne, gdyż nie dochodzi wówczas do skazania.

Pytanie: Czy w przedłożonym projekcie ministerstwo wprowadziło stosowną regulację, która uniemożliwia wykorzystywanie przez pijanych kierowców, czy mówiąc inaczej: potencjalnych zabójców, luki w prawie? Pani poseł Daria Gosek-Popiołek, Lewica. Wysoka Izbo! Pamiętam dyskusję na sali sejmowej o pierwszeństwie pieszych na pasach. Po 3 miesiącach obowiązywania tych przepisów już wiemy, jak bardzo znaczącą zmianę one wprowadziły. Statystyki nie pozostawiają żadnych wątpliwości - 30% mniej zabitych na przejściach, 30% mniej ciężko rannych. Teraz pora na kolejny krok. Jeżeli chodzi o statystyki, to Polska jest na trzecim miejscu od końca pod względem śmiertelności na drogach. Popieramy ten kierunek, natomiast są wątpliwości, jeżeli chodzi o ten projekt, chociażby te podniesione przez rzecznika praw obywatelskich, dotyczące zaostrzenia kar z art. 90 Kodeksu wykroczeń. A więc moje pytanie jest takie: Czy ministerstwo weźmie te wątpliwości pod uwagę? Bo ta ustawa powinna ratować życie. Dziękuję. Bardzo proszę, pan poseł Dariusz Kurzawa, Koalicja Polska. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze!

Przecież nadal mamy wiele wakatów w Policji, nie mamy pracowników w służbach drogowych, mamy problemy, jeżeli chodzi o infrastrukturę. A kto to będzie egzekwował? Wobec tego postulowałbym, żeby znaleźć środki przede wszystkim na to, aby zatrudnić policjantów, aby podnieść im pensje, bo to prawo, które mamy. Dzięki temu byłoby mniej wypadków na drogach i mniej ofiar śmiertelnych.

Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Panie ministrze, to wszystko, co pan tutaj powiedział, byłoby o wiele bardziej wiarygodne, gdyby pan przyszedł i powiedział: Zaczynamy od siebie.

To by było rzeczywiste wyjście naprzeciw społecznym oczekiwaniom. Ale nie od tego zaczynacie. Zaczynacie od tego, że wprowadzacie 30 tys. zł grzywny za wykroczenia określone w rozdziale XI Kodeksu wykroczeń. Jakie to są wykroczenia? Jazda hulajnogą elektryczną z prędkością inną niż zbliżona do prędkości pieszego, pozostawienie pojazdu bez oświetlenia czy też tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej, czyli protesty. Panie Ministrze! Nikt nie dyskutuje z potrzebą wprowadzenia sprawiedliwych kar dla pijanych kierowców, dla tych, którzy rzeczywiście są jak przysłowiowe pociski na drodze.

Bardzo proszę, pani poseł Klaudia Jachira, Koalicja Obywatelska. Panie Przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Kaczyński! Wysoka Izbo! Znaczne podniesienie stawek mandatów i uzależnienie składek OC od bezpiecznej jazdy jest krokiem w dobrą stronę, tylko chciałabym zapytać, co z egzekwowaniem tych nowych przepisów. Kiedy skończy się przyzwolenie na przekraczanie prędkości? Niedawno wszedł przepis o zakazie jazdy na zderzak, ale każdy, kto jechał autostradą, wie, że ten przepis jest martwy. A więc czy planujecie zwiększyć liczbę kontroli na drogach? Mam prawo jazdy od 14 lat. Przez ten czas zaledwie dwa razy byłam kontrolowana przez Policję.

Nie powinno być półśrodków (Dzwonek) ani kompromisów, jeśli chodzi o ludzkie zdrowie i ludzkie życie. Bardzo o to proszę. Pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Ten projekt jest krytykowany przez rzecznika praw obywatelskich, ekspertów i samych kierowców. Forsując swoje propozycje, nie zauważacie niedawnego raportu Najwyższej Izby Kontroli i wytycznych w nim zawartych.

Trudno oczekiwać, że samo gwałtowne zwiększenie wysokości kar odniesie oczekiwany skutek w postaci poprawy bezpieczeństwa na drogach. Dlaczego nie wprowadzicie w Polsce modelu według wzoru z Finlandii, gdzie wysokość mandatu uzależniona jest od wysokości zarobków? Jak będą rozdysponowane pieniądze z kar? Jakie będą kryteria? Dlaczego tylko na drogi krajowe, a (Dzwonek) nie na drogi gminne i powiatowe? Czy chcecie przekazać te pieniądze, tak jak to było z funduszem inwestycji lokalnych? Tylko dla swoich oczywiście. Dziękuję, pani poseł. Nie ma pana posła. Pani poseł Karolina Pawliczak, Lewica.

Wysoka Izbo! Przedkładany projekt ustawy, choć określa dobry kierunek, to jednak w wielu aspektach budzi nasze wątpliwości, stąd Lewica będzie składać do niego liczne poprawki.

Otwarcie tej definicji to zaprzeczenie podstawowych zasad gwarantujących, gwarancyjnych, które nauka prawa karnego wypracowała przez ostatnie dwa stulecia. Granice i warunki tej odpowiedzialności wykroczeniowej muszą być precyzyjnie zdefiniowane i o to proszę, licząc na poprawienie tego projektu.

Chciałabym odnieść się do kwestii sankcji i karania kierowców. Szanowni państwo, ta ustawa doprowadzi do takiej sytuacji, że osoby majętne zapłacą karę, osoby mniej majętne bądź biedne po prostu pójdą siedzieć do więzienia. Panie ministrze, może warto byłoby zacząć od siebie i pokazać, jakie państwo chcecie podjąć działania, aby wzmocnić to bezpieczeństwo, np. poprzez zwiększenie środków na modernizację dróg. Ja tylko przypomnę. Ja panu nie przeszkadzałam, panie ministrze. Ja tylko przypomnę powszechnie znane dane, że za naszych czasów rządów koalicji PO-PSL wybudowano ponad 3,5 tys. dróg krajowych, autostrad i dróg ekspresowych. Druga sprawa. Może też warto zwrócić się do zarządców dróg o pewną weryfikację oznakowania. Myślę, że każdy z (Dzwonek) nas ma przykłady, gdzie mamy przejścia, chociażby kolejowe, gdzie jest znak STOP, a one nie działają od 30 lat. Proszę się wykazać najpierw swoim działaniem, a później szukać pieniędzy na łatanie budżetu. Dziękuję bardzo. Proszę, pani poseł Marta Wcisło, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pan minister Weber mówi nam o przestrzeganiu prawa w ruchu drogowym, o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, o bezpieczeństwie pieszych, o szacunku dla prawa. Brawo, panie ministrze! To jak to bezpieczeństwo w ruchu pieszym, w ruchu drogowym ma się do faktu i do mieszkańców Janowa Lubelskiego? Jak ten szacunek dla prawa ma się w odniesieniu do ich apeli, próśb, pism i braku konsultacji społecznych? Chcecie przenieść ruch pod ich okna, pod ich domy, ograniczając im bezpieczeństwo i wyjazdy. Jesteście silni wobec słabych i słabi wobec silnych.

Pani poseł Zofia Czernow, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Prawo o ruchu drogowym zmieniane jest kilka razy w roku. Bardzo często. Wielu kierowców często nie nadąża za tymi zmianami, ale ta zmiana jest tak represyjna, tak szokująca, że postawiła na nogi wszystkich kierowców. Ja się pytam: Dlaczego pan minister nie przeprowadził szerokich konsultacji z Polakami i nie potraktował ich podmiotowo, tylko nagle przed świętami jeszcze wprowadza tak drastyczne kary? Pytam się: Ile pieniędzy z tych represji wpłynie na fundusz drogowy, bo nie ma na ten temat nic w uzasadnieniu, a ilu ludzi będzie musiało pójść do aresztu, żeby to odpracować?

Brak płynności. Dziękuję bardzo.

Pan minister w czasie debaty nad poprzednią zmianą ustawy mówił, że jest świadomy tego problemu, że pracujecie nad tym.

Jeśli chcecie naprawdę coś zrobić dla bezpieczeństwa, to pozwólcie Polakom na to, żeby się szybciej bogacili. Pozwólcie im wymieniać te auta na nowsze, na lepsze, żeby dorównywali swoimi autami sąsiadom z Zachodu, z którymi lubicie ich porównywać, mówiąc że powodują oni rzekomo mniej wypadków. Albo chociaż zmieńcie ten kretyński system OC, w którym to właściciel, a nie sprawca (Dzwonek) ponosi konsekwencje finansowe, co nie zachęca do ostrożnej jazdy. Dziękuję. Pan poseł Paweł Rychlik, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Proponowany projekt ma przede wszystkim jeden cel, zmniejszenie ilości tragedii ludzkich, do których dochodzi niestety na naszych oczach codziennie w różnych częściach kraju. Pani poseł mówiła o programie radar+. Przypominam sobie taki program w Polsce za czasów Platformy Obywatelskiej, kiedy to przy drogach jak grzyby po deszczu rosły, wyrastały nowe fotoradary, a w projekcie budżetu państwa były zapisywane prognozowane przychody właśnie z kar z fotoradarów. Tak walczyliście nie z przestępcami VAT-owskimi, ale z kierowcami i szukaliście sposobów łatania dziur budżetowych. Panie ministrze, chciałem zapytać. Powiedział pan zresztą o tym, że oprócz nowych restrykcji ważna jest poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg. Chciałem zapytać, na jaką kwotę i na jakich warunkach on będzie działał. Dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Sprawiedliwe i sprawne państwo dba o życie i zdrowie swoich obywateli. Panie ministrze, to, co jest najważniejsze, to zapewnienie prawdziwej egzekucji przepisów. Egzekucja mandatów za wszystkie wykroczenia drogowe poprzez system Centrum Automatycznego Nadzoru Ruchu Drogowego przez Policję i inne uprawnione służby powinna być prowadzona w uproszczonym postępowaniu administracyjnym, a nie jak obecnie, w postępowaniu wykroczeniowym, które niestety nieuczciwi kierowcy często wykorzystują do tego, żeby unikać kary przez przeciąganie postępowania. Według danych Najwyższej Izby Kontroli mamy kilka miliardów niewyegzekwowanych mandatów. W jaki sposób zamierzają państwo rozwiązać ten problem? Pan poseł Dariusz Klimczak, Koalicja Polska. Wysoka Izbo! Wszystkim nam zależy na bezpieczeństwie ruchu drogowego. Natomiast myślę, że w tym projekcie rządowym nie chodzi o podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale podwyższenie dochodów budżetu państwa. Gdyby państwo wykazali się implementacją dobrych rozwiązań, które funkcjonują z powodzeniem na zachodzie Europy, gdybyśmy wiedzieli, że te obwodnice, które poobiecywaliście, są budowane, ludzie by inaczej do tego podeszli. Natomiast na tak horrendalne kary, tak wysokie kary my jako PSL nigdy się nie zgodzimy. Bo wy chcecie po prostu wydoić ludzi z pieniędzy, a nie zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pani poseł Anna Maria Siarkowska, Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma pani poseł. Pan poseł Radosław Lubczyk, Koalicja Polska. Pani Marszałek! Panie Ministrze!

Dziękuję bardzo. Pan poseł Stefan Krajewski, Koalicja Polska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam konkretne pytanie. Chcecie to powiązać z wysokością ubezpieczenia.

Bo nie podejrzewam was o to, że odniesiecie to tylko do tego samochodu, w którym zostało popełnione dane wykroczenie.

Bardzo proszę, pan poseł Franciszek Sterczewski, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Cieszę się, że po 25 latach wysokość mandatów zostanie podwyższona do aktualnych potrzeb. To krok w dobrym kierunku. Ale co z egzekucją? Według NIK suma niezapłaconych mandatów to kilka miliardów złotych. Wypadki drogowe kosztują nas jako społeczeństwo ponad 57 mld zł rocznie. Ale co z fotoradarami? Pan Alvin Gajadhur, generalny inspektor transportu drogowego, rozdaje odblaski i maskotki, zamiast rozpatrywać wnioski samorządów o instalowanie fotoradarów. Na kilka tysięcy wniosków rozpatrzonych jest zaledwie kilkadziesiąt. Skąd to ślimacze tempo? Panie ministrze, co skuteczniej ratuje życie: maskotki czy ograniczenie prędkości? Pieniądze z mandatów powinny być przekazywane na rzecz funduszu DRD, na rzecz ratowników medycznych, policjantów drogówki oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pokażcie, że za słowami idą również czyny. Chodzi o życie. Pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! 8 lipca br. pod Stalową Wolą był tragiczny wypadek. Wtedy premier zapowiedział przepisy dotyczące odpowiedzialności kierowców. Zgoda, o tym chcemy rozmawiać, o tym mówił pan poseł Maciej Lasek, ale chcielibyśmy po pierwsze, żeby nastąpiło wysłuchanie publiczne. Chcemy rozmawiać o nowym szkoleniu kierowców, którzy zdobywają prawo jazdy, ale w ogóle nie jeżdżą po autostradach.

Bardzo proszę, pan poseł Tomasz Zimoch, Polska 2050.

Panie Ministrze! W swoim wystąpieniu zachęcał pan do spokojnej rozmowy, do spokojnej debaty. Zwątpiłem, kiedy obserwowałem pana reakcje. Kiedy poseł Lasek przedstawiał swój pogląd, swoje stanowisko, pan łapał się za czoło. Kiedy mówiła jedna z posłanek, pan arogancko machał dłonią. Moje pytanie jest następujące: Czy zapoznał się pan z opinią rzecznika praw obywatelskich?

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury pana ministra Rafała Webera o odpowiedź na pytania.

Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Żaden moment nie jest dobry na to, żeby wprowadzać tego typu zmiany w przestrzeni prawnej albo, z drugiej strony, każdy dzień jest dobry, żeby to robić, bo każdego dnia na polskich drogach kilka osób traci życie, każdego dnia mamy do czynienia z dramatami ludzkimi.

Nie możemy tworzyć prawa pochopnie, nie możemy tworzyć prawa na szybko i na gorąco, tylko musimy dobierać takie rozwiązania, które przede wszystkim wpłyną korzystnie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a z drugiej strony nie będą, jak to się mówi, wylaniem dziecka z kąpielą. W mojej ocenie proponowane przez Ministerstwo Infrastruktury, przez rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego przepisy są stworzone właśnie w tym duchu. Dzisiaj odpowiem na część państwa pytań. Mam nadzieję, że rozwieję wątpliwości, chociaż samo przeczytanie tego projektu pozwoliłoby uniknąć wielu pytań, szczególnie związanych z tym, na co wpłyną zwiększone mandaty czy kary zwiększonych mandatów, bo to w tym projekcie, szanowni państwo z PSL-u, jest wprost napisane. Te mandaty wpłyną do Krajowego Funduszu Drogowego, a nie do budżetu państwa. Jest to wprost napisane, nie jest to zakamuflowane, tylko jest to napisane w sposób bezpośredni. Nie widzimy w nich jakiejś przyszłości związanej z podreperowaniem systemu finansów publicznych, nie liczymy na nie, dlatego nie jesteśmy w stanie ich wyszacować.

Natomiast jeżeli to się zdarzy, to chcemy, żeby te środki wpływały na inwestycje drogowe.

To jest fakt.

Tak że, drodzy państwo, warto o tym mówić.

Jeżeli chodzi o rzeczywisty stan inwestycji drogowych, to tak on wygląda, a dzięki naszym działaniom, naszym staraniom będzie wyglądał jeszcze lepiej.

Również kwestia związana... poruszana przez wielu z państwa w oparciu o pismo rzecznika praw obywatelskich. Naprawdę nie wpadłbym na pomysł, który wskazuje, że ten projekt ustawy otwiera jakieś nadmierne czy w ogóle jakiekolwiek karanie demonstrantów, którzy protestują na ulicach. Naprawdę koncentrujemy się tylko i wyłącznie na ruchu drogowym i w tym obszarze chcemy działać. Podobnie jak kwestie płatności mandatów na miejscu. Tego prawa też nie zmieniamy. Zapisujemy tylko to, że ci, którzy będą chcieli to zrobić na miejscu, będą mogli to zrobić kartą płatniczą, czyli nie gotówką, tylko kartą płatniczą, z 10-procentowym upustem właśnie po to, żeby nie tworzyć całej papierologii, która jest związana z wypisywaniem, opłatą i później przyjmowaniem przez dany urząd skarbowy danego mandatu. Tak że ci, którzy będą chcieli to robić, po to żeby uniknąć tej całej administracji, zrobią to na miejscu, ale nie gotówką, tylko za pomocą karty płatniczej. Otóż, szanowni państwo, nic bardziej mylnego. Przecież w tym projekcie ustawy nie obniżamy dopuszczalnych prędkości, z którymi można się poruszać, nieważne, czy to w obszarze zabudowanym, czy to w obszarze niezabudowanym. Nie obniżamy minimalnych prędkości, jeżeli chodzi również o drogi szybkiego ruchu.

Mówię: co do zasady, bo każdy zarządca drogi może te zasadnicze reguły dostosowywać do realnej, bieżącej sytuacji, np. wtedy, kiedy prowadzone są zadania remontowe, zadania inwestycyjne i są utrudnienia na drogach. W ogóle w ten obszar nie wchodzimy. Wymagamy, i chyba wszyscy powinniśmy wymagać, żeby ustalone przepisy prawa były przestrzegane. Tylko tyle i aż tyle. Natomiast tych, którzy ich nie będą przestrzegać i łamią je w sposób radykalny, chcemy karać surowiej. Zobaczcie państwo, nie dotykamy sfery przekroczenia prędkości o 10 km/h. Dlaczego? Bo takie wykroczenia mają niższą ciężkość.

Cel numer dwa to walka z pijanymi na drogach. Oczywiście w ramach tej ustawy zmieniamy tylko i wyłącznie Kodeks wykroczeń, natomiast Kodeks karny, tam gdzie mówimy już o przestępstwie, czyli mówimy już o ponad 0,5 promila alkoholu we krwi, to ta będzie sprawa regulowana łącznie z konfiskatą pojazdów przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości jest w tej chwili w trakcie uzgodnień międzyresortowych, a także konsultacji społecznych projektu, który będzie tę sferę regulował.

Szanowni Państwo! Liczę na naprawdę merytoryczną dyskusję, na naprawdę merytoryczne odniesienie się do tego projektu na posiedzeniach sejmowej Komisji Infrastruktury. Jeszcze raz chcę powtórzyć, że nie zamykam się na głosy, sugestie czy poprawki, które będą miały na celu uszczegółowienie, dopracowanie przepisów, które proponujemy. Jestem przekonany, że idziemy w dobrym kierunku, że idziemy w kierunku, w którym musimy iść. Zobaczcie państwo, mówiłem o tym, inwestycje drogowe prowadzone są na skalę jak nigdy dotąd. Kampanie związane z edukacją, ze wzmocnieniem świadomości społecznej wszystkich uczestników ruchu drogowego również prowadzone są od wielu lat i będą prowadzone w kolejnych latach. Od 1997 r. nie nastąpiła nawet korekta czy nie nastąpił wzrost kwot mandatów za jakiekolwiek wykroczenia drogowe, ale skupmy się tylko na tych najpoważniejszych. To trzeba zmienić. To chcemy zmienić, bo w tym upatrujemy szansy na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mam nadzieję, że państwo nam w tym pomożecie, a jeżeli nie, to proszę o to, abyście nie przeszkadzali.

Wszelkie procedury zostały przeprowadzone zgodnie z prawem. Pani poseł chyba wie lepiej niż ja, bo tym tematem bardzo żywo się interesuje. Zdecydowana większość mieszkańców Janowa Lubelskiego popiera budowę obwodnicy Janowa Lubelskiego. Mam nadzieję, że ta obwodnica w ciągu drogi nr 74 również powstanie. Zamykam dyskusję. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy w bloku głosowań.

Wznawiam obrady. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych, druk nr 1623. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku. Powracamy do rozpatrzenia punktu 16. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1605. Czy jesteśmy gotowi do głosowań, proszę państwa?

Proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nie wierzę, żeby pod egidą pana ministra Ziobro można było gospodarować Funduszem Sprawiedliwości w sposób urągający przepisom ustawy o finansach publicznych. Nie wierzę, że minister polskiego rządu mógł przyznawać granty na projekty, za które potem sam odpowiadał na uczelni. Nie wierzę, że z tegoż funduszu, który był przeznaczony dla ofiar przestępstw, remontowano toalety w raciborskiej szkole.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ja wierzę, że minister Ziobro nie dopilnował gospodarki finansami, Funduszu Sprawiedliwości. Ja wierzę tezom, które zostały zawarte w informacji Najwyższej Izby Kontroli, że środki z funduszu były wydawane w sposób niecelowy i niegospodarny, [[Oklaski]] a praktyki sprzyjały rozwojowi korupcjogennych zachowań. W tej sytuacji wnoszę o odroczenie obrad i przygotowanie informacji przez ministra sprawiedliwości dla Wysokiej Izby na temat funkcjonowania funduszu.

Ale, panie pośle, ten mikrofon bardzo dobrze zbiera. Naprawdę nie trzeba tak krzyczeć.

Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Kiedy państwo rządziliście, na ośrodki pomocy ofiarom wydawano 1200 tys. zł, w naszych czasach to 80 mln. Przeliczcie sobie: 70 razy więcej. Po drugie, szanowni państwo, chciałbym to bardzo wyraźnie powiedzieć. Nie, to ja się pytam, gdzie były pieniądze, kiedy wy rządziliście, gdzie były pieniądze. Zapytajcie się swoich kolegów, którzy wówczas rządzili, wy również.

Panie pośle, ostrzegam pana, proszę usiąść. Dziękuję, panie ministrze. 180 mln na straże pożarne, tak, proszę państwa, na ratowanie ludzi, ratowanie życia i zdrowia ludzi. Co wam strażacy zrobili? Odpowiedzcie sobie. 16 tys. jednostek ochotniczej straży pożarnej, a wy protestujecie. Wy tego nie zrobiliście. Gdzie wy byliście? Dlaczego nie dawaliście tych pieniędzy?

Chciałabym tylko powiedzieć, że ponieważ bardzo wyraźnie. Proszę państwa, to jest skandaliczne zachowanie. Bardzo państwa proszę o zachowanie powagi. Jesteśmy na sali plenarnej. Panie pośle, jak chce pan dyskutować ze mną, to zapraszam do mojego gabinetu po zakończeniu głosowań. Proszę bardzo, wniosek formalny. Przepraszam, padł wniosek o odroczenie posiedzenia. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Kogo pani nazwała złodziejem, pani poseł? Rozumiem, że państwo odnosicie to do siebie. Bardzo dobrze, dziękuję bardzo. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Bardzo proszę. Proszę państwa, nie chcecie, żeby ktoś recenzował wasze wystąpienia z mównicy, więc proszę nie recenzować wystąpienia pana posła Winnickiego, kiedy zmierza do mównicy. Wysoka Izbo! Wnoszę o zamknięcie obrad, o zamknięcie tego posiedzenia, dlatego że myślę, że po wczorajszej debacie na temat stanu wyjątkowego na tej sali posłowie Lewicy i Koalicji Obywatelskiej zaciągnęli bardzo wiele zobowiązań, mówiąc o tym, jak bardzo chcą przyjmować imigrantów do naszego kraju. Dlatego my wychodzimy z inicjatywą, żeby zadośćuczynili temu, i wydrukowaliśmy im pierwszą stronę zaproszenia.

Co więcej, zakreśliliśmy już dla was odpowiednią opcję, że zakwaterujecie tego cudzoziemca we własnym domu.

Panie pośle, tego wniosku nie poddam pod głosowanie, bo nie możemy przerwać posiedzenia, na którym są sprawy związane z podatkami. Powracamy do rozpatrzenia punktu 16. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1605. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1605, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosowało 451 posłów. Wszyscy byli za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Powracamy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1597-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Henryka Kowalczyka o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych. W czasie drugiego czytania zgłoszono 64 poprawki. Komisja rekomenduje 26 poprawek przyjąć, 38 poprawek odrzucić. Komisja przedstawia również wnioski mniejszości, a także w dodatkowym sprawozdaniu poprawki.

Komisja wnosi o odrzucenie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość poprawek 3. i 54. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął. Nad nimi głosować będziemy łącznie. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy byli za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Sejm poprawki przyjął.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 11. i 29., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił. Obecnie w pierwszej kolejności pod głosowanie poddam poprawkę 25., której przyjęcie lub odrzucenie rozstrzygnie o innych poprawkach. W 25. poprawce wnioskodawcy proponują zmiany w przepisach ustawy nowelizującej dotyczące vacatio legis. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 25. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Głosujemy.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął. W 13. poprawce wnioskodawcy proponują m.in. nie uchylać art. 27b. Nad nimi głosować będziemy łącznie. Przyjęcie tych poprawek spowoduje bezprzedmiotowość 2. wniosku mniejszości. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Nad nimi głosować będziemy łącznie. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 17. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 20. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Poprawki 28. i 29. zgłoszone zostały do art. 9 projektu ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek mniejszości odrzucił.

Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 47. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 48. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 59. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 60. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 64. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów jest za przyjęciem całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1597 wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 17. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1601-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę panią poseł Urszulę Rusecką o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Składam dodatkowe sprawozdanie z druku nr 1601-A Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, druk nr 1509. Sejm na 38. posiedzeniu skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1601 do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Komisja przedstawia jednocześnie wnioski mniejszości oraz poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Ich przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawek 13. i 16. oraz obu wniosków mniejszości. Głosujemy.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił. Ich przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawek 5. i 6. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 4. i 7., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 13. i 16., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

W 2. wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują skreślenie art. 55. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 31. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 32. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1601 wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Rolnictwa i Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1551-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Aleksandra Mrówczyńskiego o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dodatkowe sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Rolnictwa i Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, druk nr 1454.

Komisje przedstawiają w dodatkowym sprawozdaniu wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości oraz poprawki, nad którymi Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności. pod głosowanie poddam zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. Jego przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość pozostałych propozycji. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 11. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 12. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 13. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 14. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 16. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 17. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 20. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Komisje wnoszą o odrzucenie tych poprawek. Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 22. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 27. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 29. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisje wnoszą o przyjęcie tej poprawki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 30. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 33. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 34. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 37. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1551, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1430-A. Proszę pana posła Kazimierza Moskala o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Przedstawiam dodatkowe sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, druk nr 1398. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrzyła 30 września 2021 r. poprawki zgłoszone w drugim czytaniu.

Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości oraz poprawki. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddam wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. Komisja wnosi o odrzucenie tego wniosku. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1430, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1553-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę panią poseł Annę Paluch o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! W czasie drugiego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji została złożona jedna poprawka. Ta poprawka polega na tym, że górna granica kar za niewłaściwej jakości przekazywanie danych wraca do aktualnej wysokości 25 tys. zł. Trzeba podkreślić, że kara będzie mogła być proporcjonalna, bo będzie mogła być naliczana od 200 zł za każdy dzień do 25 tys., niemniej jednak połączone komisje rekomendują Wysokiej Izbie przyjęcie tej poprawki. Komisje przedstawiają również w dodatkowym sprawozdaniu poprawkę, nad którą Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności.

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1553, wraz z przyjętą poprawką, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Powracamy do rozpatrzenia punktu 10. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1603-A. Proszę pana posła Andrzeja Szlachtę o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Komisja Finansów Publicznych na wczorajszym posiedzeniu rozpatrzyła dwie poprawki złożone podczas drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1547. Komisja obie poprawki zaopiniowała negatywnie i rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie przedmiotowego projektu ustawy w całości. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1603. Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość 2. poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1603, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1592-A. Proszę pana posła Jerzego Małeckiego o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawiam dodatkowe sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Komisje rekomendują przyjęcie ww. ustawy w całości. Komisje przedstawiają również w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności. Obie poprawki zgłoszone zostały do art. 1 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 1451, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Powracamy do rozpatrzenia punktu 12. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw. Proszę pana Krzysztofa Janusza Kozika o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1503.

Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 30 września 2021 r. proponuje trzy poprawki odrzucić, jedną poprawkę przyjąć. Komisja przedstawia również dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1602, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 13. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1555-A. Proszę pana posła Daniela Milewskiego o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Komisja Ustawodawcza po rozpatrzeniu zgłoszonej poprawki rekomenduje jej przyjęcie, jak również wnosi o uchwalenie całości projektu ustawy. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1555. Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu poprawkę, nad którą Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności. W jedynej poprawce do art. 4 wnioskodawcy proponują wyrazy „dzielnicy miasta stołecznego Warszawy” zastąpić wyrazami „miasta stołecznego Warszawy” Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? A już teraz działa, bo u mnie też nie działało.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1555, wraz z przyjętą poprawką, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego. Powracamy do rozpatrzenia punktu 18. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1596-A. Proszę panią poseł Gabrielę Masłowską o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Podczas drugiego czytania rządowego projektu ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego, druk nr 1541, zgłoszono 11 poprawek. Sejm na 38. posiedzeniu skierował te poprawki ponownie do rozpatrzenia w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Finansów Publicznych.

Komisje w dodatkowym sprawozdaniu przedstawiają również poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Z poprawką tą łączą się poprawki od 7 do 11. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1596, wraz z przyjętą poprawką, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Powracamy do rozpatrzenia punktu 19. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Wsi o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1594-A. Proszę pana posła Jana Dudę o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawić dodatkowe sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, druk nr 1502. W trakcie drugiego czytania zostało zgłoszonych 12 poprawek do projektu ustawy. Komisje na wspólnym posiedzeniu rozpatrzyły zgłoszone poprawki i wnoszą o przyjęcie przez Wysoką Izbę poprawek 4., 8., 9. i odrzucenie pozostałych poprawek. Komisje przedstawiają również w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Głosujemy. Kto jest przeciw?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Pani poseł, u kogo nie działa?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Nie działa? Ja poczekam. Dobrze.

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest przyjęciem 4. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1594, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Powracamy do rozpatrzenia punktu 9. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1565-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Andrzeja Szlachtę o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Komisja Finansów Publicznych na wczorajszym posiedzeniu rozpatrzyła dwie poprawki złożone do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw z druku nr 1565. Obie poprawki komisja zaopiniowała pozytywnie i rekomenduję w imieniu komisji ich przyjęcie. Komisja rekomenduje również przyjęcie w całości przedmiotowego projektu ustawy. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1565. Komisja w dodatkowym sprawozdaniu przedstawia poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Obie poprawki zgłoszono do art. 1 projektu ustawy nowelizującej, zawierającego zmiany do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 20. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1604-A. Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki z dnia 1 października br. o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie, druki nr 1590, 1604 i 1604-A. Komisja rozpatrzyła trzy poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania i zaopiniowała, aby poprawki 1. i 3. odrzucić, poprawkę 2. przyjąć. Przy wielkiej aprobacie całej komisji wnosimy o przyjęcie w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1604. Komisja przedstawia jednocześnie wnioski mniejszości oraz poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przekrzykuję samą siebie, bo słyszę państwa, a nie słyszę siebie. Bardzo proszę, trochę spokojniej. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1604 wraz przyjętą poprawką, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o sporcie. Powracamy do rozpatrzenia punktu 25. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1616-A. Proszę pana posła Henryka Kowalczyka o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Do ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 w czasie drugiego czytania zgłoszono osiem poprawek. Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła poprawki i rekomenduje jedną poprawkę o charakterze legislacyjnym przyjąć, a pozostałe poprawki odrzucić. Komisja przedstawia również wniosek mniejszości oraz w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 200 mln zł. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 3 mld zł. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 3 mld zł. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto za pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

We wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują w części 39: Transport zmniejszyć wydatki o kwotę 10 mln zł. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne zmniejszyć wydatki o kwotę 16 mln zł. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. W 8. poprawce wnioskodawcy proponują zmianę w załączniku nr 6 zawierającym wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwotę tych dotacji w 2021 r. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1616 wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 26. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. Proszę pana posła Henryka Kowalczyka o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! W czasie drugiego czytania do ustawy okołobudżetowej zgłoszono dwie poprawki. Komisja przedstawia jednocześnie poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1615, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Powracamy do rozpatrzenia punktu 28. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Krystyny Malinowskiej reprezentowanej przez adwokat Aleksandrę Głogowską z dnia 23 października 2018 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Małgorzaty Gosiewskiej. Na podstawie art. 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zgodą Sejmu. Przypominam, że Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych na podstawie art. 7c ust. 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora proponuje, aby Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Małgorzaty Gosiewskiej. Na podstawie art. 7c ust. 6 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów. Głosować będziemy nad wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Małgorzaty Gosiewskiej. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku oskarżyciela prywatnego Krystyny Malinowskiej reprezentowanej przez adwokat Aleksandrę Głogowską z dnia 23 października 2018 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Małgorzaty Gosiewskiej za czyn określony w tym wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Za - 71, 308 - przeciw, wstrzymało się 33.

Powracamy do rozpatrzenia punktu 30. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, który poddam pod głosowanie. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 1515, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Na podstawie art. 87 ust. 2, w związku z art. 90 ust. 1 regulaminu Sejmu, kieruję ten projekt ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia. Powracamy do rozpatrzenia punktu 34. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, który poddam pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku oznaczać będzie, że Sejm zgodnie z propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu, skierował ten projekt ustawy do Komisji Infrastruktury w celu rozpatrzenia. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 1504, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował ten projekt ustawy do Komisji Infrastruktury w celu rozpatrzenia. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 35. porządku dziennego: Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2020 roku wraz z opinią Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (druki nr 1329 i 1501) - głosowanie. Na 37. posiedzeniu Sejm przeprowadził dyskusję nad sprawozdaniem z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2020 r. Pod głosowanie poddam propozycję przyjęcia sprawozdania. Odrzucenie tej propozycji oznaczać będzie, że Sejm sprawozdania nie przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2020 r. zawartego w druku nr 1329, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 36. porządku dziennego: Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1623) Prezydium Sejmu na podstawie art. 20 ust. 1 regulaminu Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 1623, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm podjął uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Na tym zakończyliśmy głosowania. Ogłaszam 5 minut przerwy.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 37. porządku dziennego: Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2021 r. (przewodnictwo Portugalii w Radzie Unii Europejskiej) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druki nr 1528 i 1572) Proszę ministra do spraw Unii Europejskiej pana Konrada Szymańskiego o przedstawienie informacji. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czas prezydencji portugalskiej to było kolejne 6 miesięcy, kiedy głównym wyznacznikiem, zasadniczym wyznacznikiem działania Unii były konsekwencje pandemii. Szczęśliwie już nie te najbardziej palące problemy bezpośrednio związane z zagadnieniami medycznymi, zdrowotnymi czy dostępnością szczepionek. Te problemy zostały rozwiązane, natomiast przede wszystkim chodziło o konsekwencje ekonomiczne. Najważniejszą z konkluzji, które po pandemii próbuje wyciągać Unia, to oczywiście jest ograniczenie zależności od krajów trzecich w obszarze polityki handlowej, polityki przemysłowej. Polska była jednym z promotorów takiego myślenia, uznając, że jeżeli doświadczenie pandemii ma przynieść coś ważnego w Unii, to przede wszystkim ograniczenie zależności nie tylko w kwestiach medycznych, ale chociażby w kwestiach cyfrowych. W obszarze budowania odporności, tak jak to nazwała prezydencja, na pewno należy postrzegać debatę dotyczącą migracji i azylu. Polska doprowadziła do przełomu, jeśli chodzi o myślenie europejskie w tym obszarze. Zaznaczaliśmy, że jakakolwiek polityka migracyjna jest zależna od tego, czy będziemy w stanie skutecznie chronić granicę zewnętrzną. Dzisiaj w bardzo dramatycznych okolicznościach przekonujemy się, że mieliśmy w tej sprawie rację. Kolejna sprawa to blok zagadnień klimatycznych. Na początku trzeba zaznaczyć, że Polska, podobnie jak wszystkie kraje Europy Środkowej, oczekuje przede wszystkim elastyczności dotyczącej tej polityki, tak aby tempo, scenariusz transformacji były dostosowane do naszych warunków społecznych i gospodarczych. To jest zagwarantowane przez fakt, że cele transformacji są ustalone na poziomie ogólnounijnym. To daje pole tej elastyczności.

Chodzi przede wszystkim o to, aby koszty, ciężary były rozłożone w sposób sprawiedliwy zarówno między kraje, jak i między branże, a także między grupy społeczne. Polityka klimatyczna, transformacja energetyczno-klimatyczna nie mogą wiązać się ze wzrostem ubóstwa energetycznego. Jednocześnie podkreślamy, że kraje Europy Środkowej, w tym Polska, we własnym interesie muszą prowadzić ambitną politykę w tym względzie, ponieważ opóźnianie transformacji energetycznej powoduje tylko i wyłącznie wzrost kosztów tego procesu. Po pierwsze, na rozporządzeniu rynkowym, którego zadaniem jest wymierzenie lepszych zasad gry, jeśli chodzi o relacje między dużymi platformami a resztą rynku.

W obszarze społecznym, który był bardzo ważny dla Portugalii, dla rządu portugalskiego, mieliśmy szczyt społeczny w Porto. Polska przy prowadzeniu niezwykle ambitnej polityki społecznej zwraca uwagę na to, że w tej sprawie kluczową rolę odgrywają kompetencje państw członkowskich i wszystkie te dokumenty, te deklaracje nie powinny sugerować nawet rozszerzenia kompetencji prawodawczych Unii Europejskiej w obszarze społecznym. Ostatni aspekt to kwestie globalne, międzynarodowe. Po pierwsze, negatywny rozwój wypadków na Białorusi, falę represji po wyborach. To spowodowało, że Polska z sukcesem zmobilizowała opinię europejską, by przyjąć czwarty pakiet sankcji wobec Białorusi, a także aby zaoferować demokratycznej Białorusi, przyszłej Białorusi, realne wsparcie, realną perspektywę współpracy z Europą. Ta odpowiedź złożona z dwóch komponentów: bardzo twardej opozycji wobec aktualnego reżimu i możliwie daleko idącej otwartości na przyszłość, jest, myślę, warunkiem koniecznym powodzenia tej polityki. To ściśle powiązane tematy.

Jednocześnie potwierdziliśmy przywiązanie do kluczowych zasad, które powinny rządzić polityką Unii Europejskiej wobec Rosji. Po pierwsze, jest to realizacja porozumień mińskich, poszanowanie integralności Ukrainy, wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego i utrzymywanie współpracy z Federacją Rosyjską tylko i wyłącznie na tym możliwie najniższym poziomie, gdzie obie strony mają wyraźną wspólnotę interesów. Ostatnim elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę, to bardzo niewielki, bardzo niezadawalający postęp, ale jednak postęp, w obszarze polityki rozszerzenia, w szczególności wobec Bałkanów Zachodnich. Przyjęliśmy nową metodologię rozszerzenia wobec Serbii i Czarnogóry. Udało się zwołać dwie konferencje międzyrządowe. Niestety tego samego nie udało się uczynić w stosunku do Albanii i Macedonii Północnej. To są elementy polityki Unii Europejskiej, które są niezgodne z europejskim interesem. W europejskim interesie jest prowadzenie aktywnej polityki rozszerzenia, aktywnej polityki w rejonie Bałkanów Zachodnich. Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że w obszarze międzynarodowym ta prezydencja była skoncentrowana, skupiona na bardzo ważnych zagadnieniach, w szczególności w stosunku do Białorusi i Rosji. To są zagadnienia kluczowe także z polskiego punktu widzenia. Jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, mieliśmy do czynienia przede wszystkim z pewnym postępem, jeżeli chodzi o europejską odpowiedź na gospodarcze konsekwencje pandemii, w szczególności w obszarze ograniczenia zależności od państw trzecich. Bardzo proszę o przyjęcie przez Wysoką Izbę szczegółowej, dużo bardziej szczegółowej niż moje wystąpienie, informacji na temat polityki polskiej w obszarze Unii Europejskiej w czasie prezydencji portugalskiej. Dziękuję bardzo. Proszę pana posła Andrzeja Grzyba o przedstawienie uzasadnienia projektu uchwały.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedkładam w imieniu Komisji do Spraw Unii Europejskiej projekt uchwały, w którym to komisja zwraca się do Wysokiego Sejmu o przyjęcie informacji przedłożonej przez rząd w sprawie polskiej aktywności w okresie przewodnictwa Portugalii w Radzie Unii Europejskiej. Taka jest konkluzja po debacie i takie było głosowanie w Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

Przez to też otwarła się pewna nowa możliwość, jeżeli chodzi o szczyt Unia - Stany Zjednoczone, który otwiera, wydaje się, drogę do pewnej nowej ery w relacjach pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Nie będę szerzej do tego wracał, ponieważ mówił o tym pan minister Szymański. Ale to, co było najważniejsze, co najbardziej oczywiście interesowało wszystkie państwa członkowskie i wszystkie instytucje unijne, to oczywiście kryzys pandemiczny czy postpandemiczny. To zajmowało najwięcej czasu. Oczywiście w tym otoczeniu też należy wspomnieć o tym, że kwestie presji migracyjnej nie zostały w żaden sposób, w szczególności ze strony kontynentu afrykańskiego, w jakiś sposób rozpatrzone. Nie znaleziono nowych instrumentów, które by w tych relacjach mogły cokolwiek pomóc, dlatego że ten szczyt Unia - Afryka po prostu się nie odbył w okresie prezydencji, a to było jedno z takich priorytetowych założeń, jeżeli chodzi o Europę globalną ze strony prezydencji. My oczywiście mamy pewne zastrzeżenia do umowy Unia - Mercosur. Jest to jeden z tych elementów. Europa odporna, cyfrowa, zielona, socjalna i globalna - takie były generalne zawołania, które prezydencja portugalska założyła sobie w trakcie swojego półrocznego przewodnictwa w Unii Europejskiej. 20 stycznia premier Portugalii António Costa przedstawił w Parlamencie program prezydencji. Szczepienia przeciw COVID-19, ale to jeszcze w tym kontekście pełnego zaopatrzenia wszystkich państw członkowskich w szczepionki. Wydaje mi się, że w tym mieściła się też kwestia pomocy dla krajów trzecich, bo przecież Unia Europejska jest jednym z najważniejszych donatorów finansujących akurat te szczepionki dla krajów trzecich. Bez rozwiązania tej kwestii w sensie globalnym, a w szczególności w sąsiedztwie Unii Europejskiej, trudno będzie mówić o jakimś istotnym otwarciu. I oczywiście transformacja cyfrowa i klimatyczna oraz wzmocnienie filaru praw socjalnych oraz relacji ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, Wielką Brytanią, która już jest poza Unią Europejską. Wzywał jednocześnie do współpracy w celu osiągnięcia tych celów. Wezwanie było adresowane nie tylko do Parlamentu Europejskiego i Komisji, ale też do wszystkich państw członkowskich.

Te cele były również prezentowane w Komisji do Spraw Unii Europejskiej przez ambasadora Portugalii. Jednym z najważniejszych wydarzeń prezydencji, co podkreślał też w swoim przedstawieniu w Wysokiej Izbie pan minister Szymański, był szczyt społeczny, który był głównym przedsięwzięciem w kwestiach społecznych ze strony prezydencji portugalskiej.

Dlatego podkreślam ten element działań prezydencji, ponieważ zawarte porozumienie de facto określa podstawowe reformy w ramach WPR, a to m.in. dotyczy wprowadzenia planów strategicznych wspólnotowej polityki rolnej.

W tej materii Polska jest jeszcze przed tą decyzją. Jak wyglądała aktywność Polski w obszarach priorytetowych?

Chcę wspomnieć dla porządku o tym - za każdym razem o tym mówimy - jakie były transfery finansowe.

Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję. Jako pierwszy pan poseł Sylwester Tułajew w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec informacji pana ministra, informacji rządu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach w Unii Europejskiej od stycznia do czerwca 2021 r., czyli podczas kolejnej już prezydencji, prezydencji portugalskiej.

To niezwykle obszerny dokument, bo warto zaznaczyć, że ten dokument to ponad 120 stron informacji o pracach w Unii Europejskiej, o naszym zaangażowaniu, o tym, w jaki sposób wyglądały te prace. To, na co warto zwrócić uwagę, to przede wszystkim to, że kolejna prezydencja cały czas musiała koncentrować się na kwestiach odbudowy po-COVID-owej. Chciałbym zwrócić uwagę na dwa - a właściwie już po pewnym czasie można mówić o trzech - pakiety legislacji w zakresie rynku wspólnotowego. Ten pierwszy odnosił się faktycznie do konstrukcji rynku, czyli przede wszystkim do wyważenia relacji między dużymi platformami internetowymi a całą resztą użytkowników, w szczególności pod kątem gospodarczym. Przede wszystkim chodzi tu o interoperacyjność, o dostęp do danych, lepszą regulację nieuczciwych praktyk konsumenckich.

To, na co chciałbym zwrócić uwagę w moim wystąpieniu, to przede wszystkim Europejska Unia Zdrowia. W tym obszarze oprócz pewnych zmian, oprócz wzmocnienia mandatu agencji medycznej, agencji ds. zapobiegania i kontroli chorób bardzo ważnym niewątpliwie zagadnieniem i elementem jest inicjatywa HERA.

No i oczywiście otwarta autonomia strategiczna, to przede wszystkim ścisłe strategiczne zagadnienia związane z relacjami Unii Europejskiej ze światem zewnętrznym. Bardzo ważne zagadnienie. Mam na myśli przede wszystkim Partnerstwo Wschodnie, Bałkany Zachodnie, Stany Zjednoczone, w szczególności po zwycięstwie prezydenta Joe Bidena, relacje z Wielką Brytanią, która jest krajem trzecim o bardzo specyficznym położeniu względem Unii Europejskiej, i oczywiście relacje z Rosją.

Myślę, że na uwagę zasługuje porozumienie i bardzo szybkie, efektywne wdrożenie cyfrowych zaświadczeń o szczepieniu, o przeprowadzonym teście bądź przebytej chorobie, czyli nabyciu odporności własnej. To ma znaczenie o tyle, że dokument, ta platforma cyfrowa zagwarantowała rzeczywiście daleko idące wzajemne uznawanie dokumentów, które są wystawiane przez poszczególne administracje narodowe. Panie Marszałku! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wnoszę o przyjęcie tej informacji i poparcie projektu uchwały, który przedstawiła Komisja do Spraw Unii Europejskiej. Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Bardzo szczegółowo i niezwykle precyzyjnie została przedstawiona ocena - zarówno prezydencji portugalskiej, jak i wkładu polskiego rządu w prace Unii Europejskiej w trakcie prezydencji portugalskiej - przez pana ministra Szymańskiego i w szczególności przez sprawozdawcę naszej Komisji do Spraw Unii Europejskiej pana posła Andrzeja Grzyba i nie wymaga ani rozszerzania, ani dodatkowego omawiania, bo jest to niezwykle precyzyjne i niezwykle jasne.

A zatem prezydencja portugalska nakreśliła najważniejsze kwestie dotyczące zwalczania skutków pandemii, a także przygotowywania wspólnie Unii Europejskiej na przyszłość, by podobne sytuacje nie były tak bardzo zaskakujące i byśmy potrafili sobie z nimi radzić łatwiej, skuteczniej czy szybciej.

Zaraz wyjaśnię, dlaczego do tego na chwilę wracam. Otóż w roku 2007 prezydencja portugalska - za to powinniśmy być jej zawsze ogromnie wdzięczni i warto o tym przypominać, bo zapominamy - doprowadziła do podjęcia niezwykle istotnej dla nas decyzji, a mianowicie rozszerzenia strefy Schengen.

Otóż, Wysoka Izbo, jest to możliwe wtedy, kiedy jest dobra współpraca, wzajemne zrozumienie i poszukiwanie wspólnych interesów, a nie szukanie tego, co nas różni, tego, co nas dzieli, czy tego, czym możemy się nawzajem obrazić. Na tym polega ogromny sukces, na tym polegał także sukces wielu naszych polskich działań we wspólnocie. Dzisiaj te trudne wyzwania, przed którymi stanęła prezydencja portugalska w Radzie Unii i przed którymi stanęliśmy wszyscy, wymagają od nas jeszcze większego wysiłku co do wspólnych działań, bowiem uwspólnotowienie rozwiązywania problemów pokazuje, że możemy to zrobić lepiej, szybciej i skuteczniej w przeróżnych obszarach, tych, co do których Unia oczywiście ma kompetencje. By mogło to mieć miejsce, musi być jasny i klarowny system działania krajów członkowskich w Unii Europejskiej. Bo czymże jest Unia Europejska? My także jesteśmy Unią Europejską. A zatem krytykując ją czy na nią narzekając, krytykujemy samych siebie. Do tego potrzebna jest także jasna i klarowna sytuacja co do zarządzania polityką unijną.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2021 r., tj. w czasie przewodnictwa Portugalii w Radzie Unii Europejskiej (druk nr 1528) Okres od stycznia do czerwca był okresem pełnym wyzwań, przed którymi stanęła Europa. Związane to było przede wszystkim z pandemią koronawirusa. W tym roku jednak byliśmy już bogatsi o doświadczenia roku ubiegłego, ale przede wszystkim bogatsi o opracowanie szczepionki przeciwko COVID-19. Jednak samo to opracowanie nie dało rozwiązania problemu szalejącej pandemii. Należało jeszcze bowiem w sposób sprawiedliwy i rozsądny rozdzielić dawki poszczególnym państwom i grupom społecznym. Nie było to łatwe zadanie. Łatwe nie było również zachęcanie znacznej części społeczeństwa do tego, aby w momencie, kiedy nie było już problemów z dostawami szczepionek, obywatele chcieli z nich skorzystać.

Po udanych porozumieniach zawartych rok wcześniej należało w końcu zaimplementować krajowe plany odbudowy w poszczególnych 27 państwach członkowskich. Niestety problemy polityczne w wielu krajach, w tym również w Polsce, przedłużyły ten proces, przez co Unia nie była w stanie uruchomić pierwszych transz finansowych na pomoc dla krajów.

Postawiono sobie ten główny cel, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., a do 2030 r. wspólne - warto podkreślić to słowo „wspólne” - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 55% w stosunku do roku 1990. Prezydencja portugalska poniosła pewne porażki, chociażby nie zrealizowano umowy Unia - Afryka ani nie było sukcesów w polityce rozszerzeniowej w stosunku do Macedonii Północnej i Albanii. O tym mówił pan minister Szymański. Przechodząc do roli, jaką nasz kraj odegrał w tym czasie w pracach Unii, należy stwierdzić, że nie wykorzystaliśmy tego czasu tak, jak mogliśmy. Prezydencja portugalska nie odpuściła w tym czasie tematu związanego z praworządnością. Unia w dalszym ciągu naciskała na nasz rząd w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, uznając jej funkcjonowanie za niezgodne z prawem. Należy również podkreślić, że w tym czasie mieliśmy sytuację związaną z kopalnią w Turowie. To, że pracujemy razem w ramach Grupy Wyszehradzkiej, nie uchroniło nas od tego elementu, można powiedzieć, konfliktu z Czechami.

Oceniając te wszystkie działania na szczeblu międzynarodowym, szczególnie w kontekście polskim, klub parlamentarny Lewicy negatywnie ocenia przedstawioną informację.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Po pierwsze, był to okres pracy nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy.

Myślę, że to nie jest dobry sposób wyłączania polskiego parlamentu z dyskusji nad takim projektem.

Tego zabrakło. Sądzę, że jest to doświadczenie na przyszłość. Trzeci element to reforma wspólnotowej polityki rolnej.

Obszary wiejskie mają korzystać z polityki spójności w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz programu operacyjnego na szczeblu krajowym. Czwarta sprawa to polityka klimatyczna.

Oczywiście spodziewałbym się, że skoro decyzja rządu była pozytywna, to również większość parlamentarna będzie w tej sprawie wypowiadała się wspierająco, jeżeli chodzi o te rozwiązania, a tu mamy wiele krytycznych ocen. Proszę państwa, chcę zwrócić uwagę na coś, co będzie bardzo istotne.

Do tego się trzeba przygotować, bo ktoś będzie musiał to wykonać, fizycznie wykonać, a wiemy, jakie są w chwili obecnej trudności, jeżeli chodzi o potencjał wykonawczy. Przepływy finansowe. Z jednej strony są te pozytywne, które tutaj wskazywałem i o których mówił również pan minister, a z drugiej strony widzieliśmy raport pana europosła Jakiego. Myślę, że w tej sprawie potrzebna jest jakaś generalna debata tutaj, w Wysokiej Izbie, aby nie powstawało takie wrażenie, że oto zupełnie inne mamy wyobrażenie, oceniając półroczne prezydencje, a zupełnie inny wymiar dotyczy tych ocen generalnych, łącznie z przepływami rynkowymi. Dziękuję bardzo. Pan poseł Krystian Kamiński, koło Konfederacji.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym omówić dwa tematy, które w tym czasie były najbardziej istotne z punktu widzenia polskiego interesu narodowego. Po pierwsze, działania klimatyczno-energetyczne, po drugie, Fundusz Odbudowy. Można powiedzieć, że te sprawy, patrząc od początku roku, z miesiąca na miesiąc dla Polski i Polaków przybierały coraz gorszy obrót. W związku z jednoznacznie niekorzystnym dla nas pakietem energetyczno-klimatycznym, z europejsko-germańskim zielonym ładem ceny prądu w Polsce rosną praktycznie najszybciej w Europie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydaje dodatkowo wyroki karzące nas milionami złotych dziennie za funkcjonowanie kompleksu energetycznego w Turowie, w momencie gdy tak po czeskiej, jak i po niemieckiej stronie kopalnie i elektrownie tego typu funkcjonują bez żadnych problemów. Mało tego, Niemcy, co ciekawe, w pierwszym półroczu zwiększyli zapotrzebowanie na energię o 4,3%. A z czego ona pochodziła? Pochodziła ona w dużym stopniu ze zwiększonego spalania węgla brunatnego - o 30% oraz kamiennego - o 23%. Najważniejszym składnikiem miksu energetycznego w Niemczech jest gaz ziemny - ponad 30%.

A spełnienie tych oczekiwań doprowadziłoby do katastrofy energetycznej w Polsce. Zdecydowanie nie powinniśmy się na to zgadzać. Drugi temat: Fundusz Odbudowy, który my słusznie i właściwie nazywamy funduszem zadłużenia. Miliardy, które mieliśmy dostać i które były odmieniane przez wszystkie przypadki, a nawet widzieliśmy już na billboardach, jak je wydajemy, nie wzięły się z nieba.

Chociaż kwestia ich wydawania też robi się coraz bardziej dyskusyjna. Wiemy, że temat praworządności czy kwestie związane ze środowiskami tęczowymi powodują, że części tych pieniędzy możemy już nie dostać, o czym jest coraz głośniej i co coraz bardziej widać. Jest to kolejny szantaż, którego Polska staje się ofiarą. Ostrzegaliśmy przed tym rząd, aby nie dawać Unii Europejskiej do ręki takiego lewara, dzięki któremu ten szantaż mógłby zaistnieć, ale rząd zawsze wie lepiej, a potem ze zdziwieniem odpowiada: a kto mógł wiedzieć. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mottem tej prezydencji była taka oto sentencja: Czas na zapewnienie uczciwej, zielonej, cyfrowej odbudowy. Biorąc pod uwagę te słowa, a z drugiej strony politykę Prawa i Sprawiedliwości, chcę powiedzieć, że to musiał być dla tego rządu niezwykle trudny czas, bo przecież ani uczciwie, ani cyfrowo, ani tym bardziej na zielono ten rząd Polski nie buduje. Priorytety prezydencji można przyporządkować do pięciu obszarów, jak Europa: odporna, zielona, cyfrowa, socjalna i wreszcie globalna. Prezydencja Portugalii szczególną wagę przykładała także do promowania podstawowych wartości i zasad Unii Europejskiej, takich jak praworządność czy prawa człowieka.

Nie mam dobrych informacji. Pomimo że przyjęcie krajowych planów odbudowy było jednym z priorytetów tej prezydencji, to rząd robił naprawdę wszystko, co tylko można było, aby te środki nie trafiły do Polski. Nie lepiej rząd wyglądał w kwestiach polityki klimatycznej. Większość rządów w Europie chciała chronić życie obywateli, za wyjątkiem rządu Prawa i Sprawiedliwości, który uparcie robił wszystko w czasie tego półrocza, aby truć Polskę i nadal niszczyć klimat. To działanie wprost na szkodę naszego państwa i kolejnych pokoleń młodych Polek i Polaków. W informacji znajdujemy także takie kwiatki, jak ten, że Polska popierała inicjatywy w zakresie praworządności. W tej informacji czytamy także, że promocja praw człowieka należy do priorytetów polskiej polityki zagranicznej i że to się odbywało w trakcie tej prezydencji, a głównymi obszarami tematycznymi, jeśli chodzi o zaangażowanie Polski, była promocja demokracji oraz dobrego rządzenia, ochrona praw najsłabszych grup, w tym także dzieci. I to, że w tej informacji znalazły się takie zdania, to jest absolutny skandal. Politycy tego rządu wydają rozkazy, aby małe dzieci wypychać poza granicę. To jest łamanie nie tylko praw człowieka, ale także brak jakiejkolwiek przyzwoitości. Panie ministrze, ten rząd promuje agresję i arogancję, a nie troskę. Szanowni Państwo! W imieniu Koła Parlamentarnego Polska 2050 wnoszę o odrzucenie tej informacji. Ona absolutnie odbiega od tego, co (Dzwonek) na co dzień widzimy. Dziękuję bardzo. Do pytań zgłosili się. Nie ma takiej możliwości, panie pośle.

Pan poseł Andrzej Szejna, Lewica. Wysoka Izbo! Ja panu ministrowi trochę współczuję jako ministrowi do spraw europejskich, że musi pracować w rządzie antyeuropejskim. Kontynuując znakomite wystąpienie pana posła Jacka Czerniaka, chciałem zadać kilka pytań.

Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałem zapytać o ten udział w pracach i te najważniejsze priorytety Polski w trakcie prac w Unii Europejskiej. O części już mówiłem, takich jak promocja praw człowieka i promocja ochrony praw najsłabszych grup, w tym praw dzieci. W jaki sposób, jakie to są wartości, skoro rząd postępuje tak, jak to widzimy, z małymi ludźmi, z dziećmi, wypycha je przez granicę? Jakie to są wartości, jakie Polska promuje w Unii Europejskiej, skoro rząd w Polsce zachowuje się zupełnie inaczej? W tej informacji, którą państwo przedstawili, jest takie zdanie, że Polska wskazywała, iż należy podjąć duży wysiłek na rzecz zwalczania szkodliwych treści, w tym dezinformacji. Pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W dokumencie czytamy peany pochwalne dla prezydencji Portugalii przy jednoczesnym w polskim życiu publicznym podważaniu autorytetu unijnych organów, nieuznawaniu wyroków TSUE czy wreszcie wobec wniosku premiera do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie wyższości prawa polskiego nad unijnym. Z jednej strony Polska wnioskuje o przyznanie możliwie wysokich środków z unijnego budżetu, a z drugiej stara się przekonać unijnych komisarzy, że one wcale nie są nam potrzebne, a minister sprawiedliwości wręcz zachęca samorządy do podtrzymywania uchwał, które z automatu wykreślają je z listy beneficjentów określonych środków.

Panie Marszałku! Panie ministrze, trochę samotnie się pan chyba czuje w tej Unii Europejskiej, bowiem przystępuje pan z pozycji kraju, który jednak jest eurosceptyczny. Opinia o Polsce, praworządność, wolność słowa. Jak to wpływa na skuteczność negocjacji? Chciałbym zapytać pana, jak wyglądać będzie u nas analiza na poziomie naszego kraju i czy my budujemy jakąś większość, która będzie mogła zabezpieczyć nasze interesy, interesy obywateli w związku z czymś, co jest dużym zagrożeniem transformacyjnym związanym z tym pakietem, mianowicie ubóstwo energetyczne? Czy będzie i czy wpisujemy w swoje negocjacje walkę o środki europejskie, które zabezpieczą nas przed negatywnymi wpływami tego pakietu? Druga sprawa to taksonomia i gaz, i atom.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Pod przewodnictwem Portugalii kontynuowano m.in. prace nad projektem dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. To na pewno dobra propozycja, szczególnie dla obywateli nowych państw członkowskich, w tym Polski. Do tej pory nie wypracowano jednak wspólnego porozumienia ze względu na różne uwarunkowania możliwości finansowych państw członkowskich. Dlatego chciałbym zapytać: Jakie stanowisko w tej kwestii zaprezentował i prezentuje polski rząd oraz na jaką propozycję wysokości płacy minimalnej byłby skłonny się zgodzić? Pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050. Panie Ministrze! Podczas dyskusji Polska podkreślała zwłaszcza potrzebę zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych teleinformatycznych. W tym samym czasie w kwietniu z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wyciekło 20 tys. rekordów polskich funkcjonariuszy służb: imiona, nazwiska, adresy. W tym samym czasie Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgubił kilka, jeśli nie kilkanaście tysięcy e-maili polskich przedsiębiorców, nie wspominając o tym, że mniej więcej w tym samym czasie w tzw. aferze mailowej pana ministra Dworczyka okazało się, że ministrowie polskiego rządu w korespondencji pomiędzy sobą korzystają z darmowych i niezabezpieczonych narzędzi teleinformatycznych. Czy zamierzacie państwo wreszcie podejść poważnie do wyzwań XXI w., do bezpieczeństwa teleinformatycznego, do tego, jak bardzo w dzisiejszym świecie jest to istotne? Pan poseł Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Na początku tej kadencji w swoim exposé premier mówił, że idziemy zmieniać Europę. No i chciałem zapytać: Jak nam idzie? Co już zmieniliśmy w Europie?

I jak od tej pory udało się nam Europę zmienić od środka?

Dopóki w Polsce nie będzie poważnie leżała na stole opcja wyjścia z Unii Europejskiej, to nasza pozycja negocjacyjna będzie tam żadna.

Bardzo dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo! Rząd nie jest antyunijny, ale propolski, dlatego bardzo dziwią mnie wypowiedzi państwa, jeżeli chodzi o jakieś antyunijne doniesienia, jakoby polski rząd w jakiś sposób negatywnie odnosił się do polityki Unii Europejskiej. Natomiast nikt nie mówi o polexicie. Faktem jest np. koszt emisji i ceny gazu i wpływ tych czynników na galopujące ceny nawozów azotowych. Tak więc to, że z jednej strony państwo chwalicie Unię Europejską i na każdym kroku chcecie być państwem przedmiotowym, nie zwalnia państwa z odpowiedzialności, aby mądrze negocjować w tej Unii Europejskiej. Nie wmawiajcie więc państwo rządowi jakichś antyunijnej polityki. Jedni z państwa na słabych warunkach do tej Unii wchodzili, a drudzy z państwa bardzo słabo negocjowali ceny gazu. Pan poseł Czesław Siekierski, Koalicja Polska. Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Prace nad zasobami własnymi trwają permanentnie od dłuższego czasu. Czy w okresie prezydencji portugalskiej one w jakiś sposób się posunęły dalej?

Prezydencja portugalska przypadła po prezydencji niemieckiej, po objęciu funkcji przez prezydenta Bidena, prezydencja niemiecka w ostatnim momencie szybko podpisywała porozumienie z Chinami. Czy jest świadomość porwania łańcucha dostaw i nowego spojrzenia na globalizację? Wreszcie problem Zielonego Ładu Europejskiego i wspólnej polityki rolnej.

Panie Przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Kaczyński! Wysoka Izbo! Zacytuję kilka fragmentów z dokumentu informującego o udziale polskich pracach w Unii: Polska brała udział w wypracowaniu stanowiska Unii w odniesieniu do kwestii udziału kobiet w życiu publicznym, wzmocnienia ich roli społecznej w sferze życia publicznego, wpływu kobiet na podejmowanie decyzji oraz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Drugi cytat: Promocja praw człowieka należy do priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Trzeci cytat: Głównymi obszarami tematycznymi zaangażowania Polski były - uwaga - promocja demokracji oraz dobrego rządzenia, ochrona, promocja praw najsłabszych grup, w tym praw dzieci, osób z niepełnosprawnościami oraz osób należących do mniejszości religijnych. Naprawdę, panie ministrze? Pani poseł Urszula Zielińska, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W kontekście polityki klimatycznej starania Polski były skierowane na uzyskanie odpowiedniej ilości środków na przeprowadzenie niezbędnej transformacji. Zapotrzebowanie na środki w Polsce jest ogromne, bo rząd zaplanował, iż polska energetyka będzie oparta w przyszłości na najdroższych źródłach energii, na gazie z importu, którego ceny na giełdzie osiągnęły właśnie rekord 20-lecia, i na energii jądrowej, również jednym z najdroższych źródeł energii, również na importowanej technologii. Tymczasem środki na transformację w Krajowym Planie Odbudowy są wstrzymane, bo Polska łamie podstawowe prawa Wspólnoty Europejskiej. Idzie zima, ceny energii rosną, kary za Turów rosną. Smog truł i truje nas tak, jak truł, pieniędzy na transformację jak nie było, tak nie ma.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Filozof, socjolog Zygmunt Bauman mówił o tym, że Europa to jest niedokończona przygoda. Unia Europejska jest też formą otwartą, o czym warto pamiętać, i jest to ogromna zdobycz: to, czym dzisiaj możemy się dzielić ze społeczeństwami poszczególnych krajów, które współuczestniczą w tworzeniu Unii Europejskiej. Ale my tutaj w Polsce mamy ogromny problem, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości nie chce obecności w Unii, chce z tej Unii jak najszybciej wyjść. Pan marszałek zresztą jest również jednym z tych, którzy taką opinię wyrażali. Ale dla mnie ciągle najbardziej skandaliczna pozostaje wypowiedź prezydenta Dudy, który mówił o wyimaginowanej wspólnocie, która nam niczego właściwie nie daje. Jest ona ciągle kompromitująca.

Teraz głos ma minister do spraw Unii Europejskiej pan Konrad Szymański. Panie Marszałku! Postaram się odnieść do wielu wątków, które tutaj zostały poruszone. Podkreślamy, że polityka społeczna jest rzeczywiście kompetencją praw państw członkowskich. Mówimy o tym często, natomiast to nie zmienia faktu, że Polska w ostatnich latach prowadzi niezwykle aktywną i ambitną politykę społeczną, że poprawiły się wszystkie wskaźniki solidaryzmu społecznego. Na forum unijnym zwracamy uwagę na to, że nie jest to konsekwencja tak lub inaczej skrojonych kompetencji unijnych, ale jest to konsekwencja bogacenia się kraju. Nie ma innej ścieżki wzrostu standardów społecznych jak po prostu bogacenie się kraju. To bogacenie jest ściśle powiązane po prostu z integracją handlową i z tym, co daje wspólny rynek. Dlatego w debacie społecznej, unijnej podkreślamy rolę przede wszystkim wspólnego rynku, co na pierwszy rzut oka pewnie dla niektórych z państwa może wydawać się zaskakujące. Wiele pytań dotyczyło polityki klimatycznej. Rama prawa klimatycznego to jest dopiero początek. Najbardziej poważne pytania stoją przed nami. Zabezpieczyliśmy w tej sprawie oczywiście rolę Rady Europejskiej, bez której nic w zakresie pakietu Fit for 55 się nie może odbyć, ponieważ są to decyzje, które mogą wpływać daleko, bardzo daleko, jeżeli chodzi o rozłożenie kosztów. Te koszty, podkreślamy, muszą być sprawiedliwe, dlatego odpowiadając na pytanie o koszty, o ochronę, o środki na transformację, mogę powiedzieć przynajmniej kilka rzeczy. Po pierwsze, Polska będzie najważniejszym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Po drugie, gdyby nie Polska, dzisiaj nie byłoby żadnego powodu, abyście państwo na tej sali mówili o szansach, które się wiążą z funduszem społeczno-klimatycznym. Ale aby był przyjęty, musimy mieć gwarancję, że z tym funduszem nie będą się wiązały obciążenia dla polskich obywateli, dla polskich gospodarstw domowych, które będą przekraczały skalę tego funduszu, a o to jest bardzo łatwo. Dlatego Polska pozostaje aktywna w tej debacie i z całą pewnością nie da się zredukować do kogoś, kto powie po prostu: nie albo po prostu: tak, bo ta sprawa jest zbyt skomplikowana, żeby upraszczać odpowiedzi do poziomu, który by się spodobał przynajmniej niektórym z państwa. Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na to, że informacja dotyczy również bilansu korzyści polskiego członkostwa w Unii. To dotyczy nie tylko transferów, ale również korzyści rozproszonych dużo bardziej, za to dużo poważniejszych - korzyści płynących ze wspólnego rynku. Dwa razy do roku informujemy Sejm o tym aspekcie polskiego członkostwa i myślę, że warto, aby to wybrzmiało. Po pierwsze - uczciwość. Padły mocne słowa, oczywiście łatwo tutaj używać mocnych słów, więc każdemu to przychodzi z dużą łatwością, ale chętnie to skomentuję. Jeżeli chodzi o uczciwość i ten rząd, to proszę zobaczyć ostatnie sprawozdanie OLAF-u, unijnej służby walki z korupcją. Zobaczycie tam państwo, że Polska należy do tych państw, które radzą sobie z problemami korupcji lepiej niż średnia unijna. Jesteśmy w gronie państw, które o uczciwość w życiu publicznym, w szczególności oczywiście, jeżeli chodzi o uczciwość wydawania pieniędzy publicznych, walczy najbardziej efektywnie. I to nie jest moja opinia, to jest opinia instytucji, do których państwo mają zwykle znacznie większe zaufanie i lubią się państwo powoływać na ich autorytet. Więc proszę zajrzeć, ostatni raport roczny OLAF-u. O Polsce jest tam dużo, dużo dobrego. Cyfrowość. Nie spodziewałem się, że można akurat temu rządowi postawić tego typu zarzuty, ponieważ pandemia pokazała, w jakim realnym stanie, nie na papierze, ale w realnym stanie cyfryzacji są poszczególne państwa. Wiele zaskakujących wniosków. Państwa, które mają wizerunek państw niezwykle efektywnych, niezwykle dobrze zorganizowanych, w tracie pandemii pokazały swoje olbrzymie słabości. Niedawno wybrzmiało to w kampanii wyborczej naszego zachodniego sąsiada z bardzo dużą siłą. Polska w tym czasie pokazała, że stopień cyfryzacji państwa, usług publicznych jest na tyle duży, że mogliśmy z łatwością użyć tych instrumentów również do tego, by pomóc ludziom w bardzo trudnych miesiącach, najgorszych miesiącach pandemii. O klimacie, o transformacji już mówiłem. Prawda jest taka, że dynamika transformacji klimatyczno-energetycznej w ostatnich 5 latach jest najwyższa przez ostatnie 20 lat. Tylko my nigdy tego nie zrobimy w sposób, który byłby nieodpowiedzialny. Będziemy to robili według własnego tempa, według własnych reguł. I tak, uznajemy, że rola gazu i rola energii jądrowej jest kluczowa dla sprawiedliwej transformacji, dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Padło generalne pytanie o skuteczność negocjacji. Zwykle trudno się odpowiada na takie pytania, ale dziś, myślę, że wciąż jest stosunkowo łatwo odpowiedzieć. Jeżeli państwo spytają w stolicach europejskich o to, to myślę, że łatwo znajdą państwo potwierdzenie tej tezy. W przypadku negocjacji budżetu wieloletniego i Funduszu Odbudowy to można zrobić, bo chodzi tylko o liczby. Te liczby są bardzo jednoznaczne. Polska jest jedynym dużym krajem Unii Europejskiej, który jednocześnie jest bardzo dużym beneficjentem budżetu wieloletniego i Funduszu Odbudowy. Myślę, że to jest miara skuteczności negocjacji. Czy te negocjacje są łatwe? Nie. Wynika to ze zmian politycznych, które dokonują się we wszystkich stolicach państw członkowskich Unii Europejskiej.

Również te państwa dzisiaj przechodzą na kurs, który, powiedzmy, nazwałbym ograniczonym zaufaniem do procesu europejskiego. To stąd biorą się problemy z procesem rozszerzania Unii Europejskiej. To stąd biorą się problemy związane z protekcjonizmem na wspólnym rynku. To stąd w końcu biorą się problemy z tym, że państwa, które zarabiają na integracji najwięcej, nie chcą płacić na wspólny budżet.

Bez Polski, bez rządu Beaty Szydło, bez rządu Mateusza Morawieckiego nie byłoby kolosalnej zmiany w zakresie polityki migracyjnej Unii Europejskiej.

To jest zmiana w bardzo ważnej dziedzinie.

Bez Polski nie byłoby rynkowych ograniczeń dla dyktatu rosyjskiego eksportu gazu na rynek europejski.

Na to miał wpływ nasz zachodni sąsiad.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

To jest bardzo dobre.

Wtedy będziemy wiedzieli tak naprawdę, ile te dobra publiczne kosztują.

To jest kwestia do dyskusji. Proszę przeczytać, jak wielu teoretyków, laureatów Nagrody Nobla w zakresie ekonomii wycenia dobra publiczne, ile one kosztują. To nie jest tak, że to jest bezpłatne. Nam się wydaje, że to jest bezpłatne, bo jest w zasięgu ręki. Tam nie ma kasjera. Tam nie ma bankomatu.

One rosną również ze względu na politykę europejską, ale nie tylko. Przecież pokłady węgla mamy coraz niżej. W związku z tym musimy mieć tę refleksję, że musimy zastępować. Każda wymiana tego bloku to jest koszt.

Dobrze, że ten proces idzie w kierunku odnawialnych źródeł energii, ale też w kierunku technologii, które być może powinny być rozwijane, chociażby takich technologii jak small modular reactor, czyli małych reaktorów jądrowych, które są dużo mniej kosztowne, mniej obciążające środowisko. Może tu znajdziemy jakiś kompromis?

To jest niezmiernie ważne pytanie. Proszę państwa, koszty ETS. Dlatego że podjęto, uważam, błędną decyzję, że one są poddane obrotowi giełdowemu na rynkach finansowych. Następuje niestety spekulacja tymi uprawnieniami. Nie wiem, czy to jest możliwe w chwili obecnej, żeby wycofać właśnie te uprawnienia. To zdecydowano się na to, że można nimi również obracać na rynkach finansowych.

Przykładem jest francuski sprawozdawca z Renew Europe, który w Parlamencie Europejskim o tym powiedział. Jeżeli takie mają być koszty społeczne, to jest to nieakceptowalne społecznie, to nie będzie do zaakceptowania.

Czyli udało się. Mimo że zaostrzone zostały kryteria związane z przyznawaniem tych uprawnień i wycofywaniem ich z rynku, udało się 30% dla polskiego sektora ciepłowniczego przyznać. Wszyscy stwierdzili, że sektor ciepłowniczy, że zorganizowane źródła ciepła sprzyjają klimatowi, w szczególności zaś kogeneracja sprzyja klimatowi. Nie.

Zawsze jest to pytanie, która narracja jest prawdziwa, to pytanie tutaj też padało, czy ta w Polsce, czy ta na poziomie europejskim. Myślę, że to jest naturalne, że w polityce, jak komunikujemy się z wyborcami, to używamy innych określeń, innych kwantyfikatorów niż te, których używamy w gremium międzynarodowym.

Nikt nie musi informować gremiów międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej, jakie są nasze poglądy. Przecież codziennie jesteśmy słuchani, codziennie jesteśmy obserwowani, również obrady tego parlamentu są obserwowane. I codziennie idą clarisy informujące o tym, jakie są rzeczywiste poglądy poszczególnych frakcji politycznych w naszym parlamencie i nasze jako polityków.

Z jednej strony zbudowaliśmy gazoport, z drugiej strony budujemy w tej chwili Baltic Pipe.

Myślę, że to byłoby bardzo ważne. W pełni zgadzam się z tym, co powiedział pan minister Szymański, że kwestia OLAF-u i tego, co wynegocjowaliśmy jako Polska, występując przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, to jest przykład korzystnych decyzji dla Polski.

Wysoka Izbo! One są takie, że powinniśmy liczyć na skrócone łańcuchy dostaw, w szczególności jeżeli chodzi o kwestię komponentów, np. do produkcji leków. Europa wyzbyła się tych komponentów. One w większości były produkowane na rynku chińskim czy indyjskim.

A więc to, co jest strategiczne z punktu widzenia europejskiego przemysłu, również polskiego przemysłu, polskiego konsumenta i odbiorcy, w dużej mierze powinno być dostępne i produkowane w Europie. Nie wszystko możemy oprzeć na usługach.

Jeżeli ten procent jest niższy, to istnieje ogromne zagrożenie dla funkcjonalności i funkcjonowania gospodarki.

To decyduje o nowoczesnych technologiach. Dziękuję bardzo za możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie. Marszałek Sejmu proponuje, aby Sejm bezzwłocznie przystąpił do drugiego czytania projektu uchwały. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Czy ktoś z pań i panów posłów chciałby zabrać głos w drugim czytaniu?

Wystarczy, panie marszałku. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Panie ministrze, odniosę się do dwóch rzeczy, o których mówił pan podczas odpowiedzi na pytania z pierwszej części debaty. Po pierwsze, kwestia polityki klimatycznej. To nie jest kwestia tego, w jakim świecie żyjemy dzisiaj. To jest kwestia tego, czy kolejne pokolenia Polek i Polaków będą mogły żyć w naszym państwie. Dzisiaj nie możemy działać na alibi. Musimy działać w taki sposób, żeby ich życie tutaj było możliwe, bo inaczej cały nasz trud w innych obszarach jest na nic. Dzisiaj po stronie rządu tej determinacji nie widzimy. Wręcz przeciwnie, cały czas widzimy działanie na rzecz niszczenia klimatu, na rzecz takich rozwiązań, które ten nasz świat czynią niezdatnym do życia. Jeżeli przedstawiacie państwo sprawozdanie, to ono powinno odzwierciedlać to, co rzeczywiście się w Polsce dzieje, jakie decyzje są podejmowane. Niestety tak się nie stało, dlatego składam poprawkę (Dzwonek), w ramach której zmieniamy projekt tej uchwały na odrzucający przedstawione sprawozdanie.

Sprzeciwu nie słyszę. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szklany Piotrków. Wjeżdżając do Piotrkowa Trybunalskiego dawną linią Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej od strony Koluszek, uważny podróżny zauważy potężną nadal zabudowę przemysłową. To pozostałości dużego kompleksu przemysłowych hut szkła o dość egzotycznych nazwach: „Kara” i „Hortensja” Ta pierwsza od zawsze produkowała asortyment ewidentnie przemysłowy: szkło okienne, które z czasem stało się jej głównym produktem, ale również butelki różnego rodzaju, cylindry oświetleniowe i wiele innych. Dopiero wtedy uruchomiono pierwszą maszynę do ciągnięcia tafli szkła. Będąca w obcych rękach „Kara” bardzo często była areną strajków robotniczych. W czasie II wojny światowej teren „Kary” był obozem pracy dla Żydów z piotrkowskiego getta.

Artystyczne wyroby z piotrkowskiej huty zachwycały i nadal zachwycają zwykłych ludzi i kolekcjonerów. Bardzo często na różnych aukcjach w Polsce i za granicą osiągają wysokie ceny. Z zakładem wiązały się całe rodziny przez wiele dziesięcioleci. Znane są w Piotrkowie dynastie hutników, którzy pracowali w niej przez cały okres jej istnienia. W roku 1989 ukazała się książka o historii huty „Hortensja” Huta ta przetrwała tylko kilka lat dłużej. Po co dziś mówię o tych zakładach? To od nich rozpoczął się prawdziwy przemysłowy rozwój Piotrkowa Trybunalskiego, który wtedy był co prawda stolicą guberni, ale praktycznie nie było tam żadnego przemysłu. Dziś hut już nie ma, ale mieszkańcy miasta nadal pamiętają o piotrkowskich hutach. Na ich gruzach powstało kilka małych firm. Pani poseł Teresa Hałas. Pan poseł Jan Szopiński. Też nie ma?

Może na piśmie pan złoży, do protokołu?

Wysoka Izbo! Ich celem była przede wszystkim budowa mieszkań na wynajem dla osób, których dochody były na tyle wysokie, że nie mogły skorzystać z pomocy mieszkaniowej samorządu, a jednocześnie były zbyt niskie, aby mogły one wziąć kredyt na własne mieszkanie. TBS-y otrzymywały wsparcie finansowe ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, jednakże okazuje się, że kontrola TBS-ów jest ograniczona, ponieważ Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować tylko te TBS-y, których wspólnikami są jednostki samorządu terytorialnego, i to tylko i wyłącznie w zakresie tzw. dyscypliny finansów publicznych. Oznacza to, że kwestia rozporządzania przez TBS-y środkami finansowymi pochodzącymi od najemców, czyli właściwie partycypantów, pozostaje poza wszelką kontrolą organów niezwiązanych z funkcjonowaniem towarzystwa budownictwa społecznego. Kolejnym zagadnieniem jest kwestia dysponowania przez TBS-y partycypacjami płaconymi przez osoby zainteresowane najmem w zasobach towarzystwa.

Pomimo bowiem wpłacenia od ok. 25% do 30% kosztów budowy danego lokalu mieszkalnego partycypant uzyskał w zamian jedynie uprawnienie do wskazania najemcy tegoż lokalu, które to prawo w przeważającej liczbie przypadków po upływie pewnego czasu określonego w umowie partycypacyjnej po prostu wygasa. Na skutek tak przyjętego rozwiązania ustawowego niektóre TBS-y pozbawiły partycypantów prawa do uzyskania zwrotu wpłaconej partycypacji w przypadku rozwiązania tej umowy. TBS-y często swobodnie dysponują wpłaconymi partycypacjami, nie informując partycypanta ani o ich przeznaczeniu, ani o postępach w spłacie kredytu. Tymczasem TBS ma obowiązek tak skalkulować czynsz, aby jego wysokość wystarczyła w danym miesiącu jedynie na spłatę raty zaciągniętego kredytu, koszty eksploatacji budynku oraz koszty remontów. Jeśli TBS pobierze od lokatorów środki na spłatę kredytu, a następnie ich nie przekaże do banku, defraudując je w istocie, to okres spłaty wydłuża się o kilka lat, a na dany lokal będzie w dalszym ciągu przypadała kwota do spłaty. TBS nie ma prawa obciążać lokatorów kilkukrotnie spłatą tego samego kredytu. Czynsz po spłacie kredytu powinien się zmniejszyć o wysokość raty. Niestety TBS-y nie są chętne, aby udzielać lokatorom jakichkolwiek informacji na ten temat. Najemcy nie wiedzą często ani na jaki okres dany TBS zaciągnął kredyt i kiedy powinna się zakończyć planowo spłata, a tym samym zmniejszyć czynsz, ani czy TBS wydłużył okres spłaty z powodu notorycznego zalegania z zapłatą. Niestety przez wiele lat funkcjonowania TBS-ów w niektórych z nich doszło do różnego rodzaju patologii i nadużyć, takich jak finansowanie z pieniędzy wpłacanych przez partycypantów koncertów muzycznych. Skoro państwo udziela takim podmiotom jak TBS-y kredytów ze środków publicznych na preferencyjnych warunkach, to powinno mieć kontrolę nad tym, jak umowy z partycypantami są skonstruowane. Z punktu widzenia prawnego partycypacja jest prawem majątkowym i podlega dziedziczeniu. Pozostałą kwotę wartości lokalu najemca spłaca w czynszu. Fakt ten ma doniosłe znaczenie, oznacza bowiem, że spłata kredytu zaciągniętego przez TBS obciąża de facto w całości nie kredytobiorcę, lecz najemcę, czyli partycypanta. Oznacza to, że najemca jest obciążony pełnym kosztem spłaty budowy mieszkania, a nigdy nie zostanie jego właścicielem. Innymi słowy, pewna grupa społeczna ze względu na dochody niewystarczające do zakupu mieszkania na własność zmuszona była wybrać TBS, aby mieć gdzie mieszkać ze swoimi rodzinami. Tymczasem ustawodawca tak niefortunnie sformułował przepisy, że ta grupa społeczna o ograniczonych dochodach zmuszona jest do fundowania gminie lub podmiotowi prywatnemu jako właścicielowi TBS-ów lokali na wynajem. Ustawa dotycząca TBS-ów musi zostać zmieniona, a zmiany winny iść w kierunku większej transparentności oraz ułatwień w uwłaszczaniu partycypantów. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Skażenie środowiska na terenach po byłych Zakładach Chemicznych Zachem w Bydgoszczy jest od wielu lat ogromnym problemem mieszkańców. Bulwersujące są w tej sprawie zaniechania i nieskuteczność działań kolejnych rządów, w tym także obu rządów Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski. Dziękuję bardzo z tego miejsca dziennikarzom „Expressu Bydgoskiego” za monitoring tego tematu i wspieranie mieszkańców Łęgnowa, walczących o czystą wodę i czyste powietrze. Przypomnę, że w bydgoskim Łęgnowie i w okolicach naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej odkryli całą listę niebezpiecznych substancji rakotwórczych. W wodach gruntowych w otoczeniu państwowego Nitro-Chemu wykryto także trotyl. Dopiero w połowie września br. regionalna dyrekcja ochrony środowiska rozpoczęła tzw. remediację, czyli oczyszczanie Łęgnowa ze szkodliwych związków chemicznych. Tyle że instalacja powinna pracować już dawno temu, a działania podjęte w związku ze skażeniem tego terenu o wartości 100 mln zł budzą liczne wątpliwości specjalistów i samorządowców. Według nich błędem jest to, że przed wybraniem terenu remediacji nie przeprowadzono kompleksowych badań środowiska gruntowo-wodnego i nie opracowano kompleksowego planu zarządzania terenem zanieczyszczonym, a projekt obejmuje zaledwie fragment strumienia zanieczyszczonych wód podziemnych. Projekt nie obejmuje także rekultywacji ogniska zanieczyszczeń, czego powodem jest brak możliwości interwencji na terenach prywatnych.

I tu, wraz z mieszkańcami Bydgoszczy, zwracam uwagę rządowi oraz Ministerstwu Klimatu i Środowiska na konieczność dokonania zmian prawnych takich, by dać regionalnej dyrekcji ochrony środowiska możliwość działania także na terenach prywatnych w szeroko pojętym interesie publicznym i w interesie mieszkańców. W tej sprawie należałoby rozważyć nawet uchwalenie specustawy. Postulujemy też, by środki przyznane Polsce na realizację Polskiego Ładu przeznaczyć na kompleksowe badania, monitoring i pełną remediację terenów poprzemysłowych, uwzględniając w tym oczywiście tereny pozachemowskie. W powyższych sprawach składam interpelację, kolejną zresztą, do ministra klimatu i środowiska i razem z samorządowcami i

Wysoka Izbo! Czarnca to miejscowość w gminie Włoszczowa, miejsce urodzenia i pochówku wielkiego hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego, który w tradycji narodowej jest wzorem niezłomnego żołnierza. Postrzegany przez potomnych jako wzór patrioty, został wymieniony w naszym hymnie narodowym. W tradycji ziemi włoszczowskiej zajmuje miejsce poczesne - jest patronem szkoły podstawowej w Czarncy, zespołu szkół nr 2 we Włoszczowie oraz największego w powiecie klubu sportowego Hetman Włoszczowa. Istotną rolę w popularyzowaniu wiedzy o tym bohaterze narodowym pełni Towarzystwo Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Czarncy. Wieloletnim prezesem towarzystwa był śp. Zygmunt Fatyga, który za działalność na rzecz krzewienia pamięci o hetmanie został uhonorowany przez prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi. Doceniono go za aktywną działalność na rzecz popularyzacji postaci hetmana, pielęgnowanie i rozwijanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczanie i odnawianie pamiątek po hetmanie, a także organizację uroczystości ogólnokrajowych. Obecnie funkcję prezesa pełni pani Wiesława Krawczyk. Od 1992 r. towarzystwo utrwala pamięć o hetmanie Stefanie Czarnieckim jako bohaterze narodowym, eksponuje jego patriotyzm i zasługi dla ojczyzny oraz związki łączące go z Czarncą i ziemią włoszczowską. Towarzystwo podejmuje wiele działań ukierunkowanych na popularyzację wiedzy i pamięci o wielki bohaterze. Odnowiło wiele pamiątek znajdujących się w miejscowym kościele, otoczyło opieką park arboretum, doprowadziło do usytuowania pomnika przed szkołą, odsłoniło tablicę pamiątkową oraz posadziło dąb przyjaźni. Wszystkie te działania miały na celu kultywowanie pamięci o wielkim człowieku, który jest naszym bohaterem narodowym. Organizacja turniejów oraz uroczystości hetmańskich powoduje, że do Czarncy zjeżdżają tłumy pasjonatów historii. Działania te znajdują odzwierciedlenie w zwiększeniu atrakcyjności turystycznej ziemi włoszczowskiej. Serdecznie dziękuję towarzystwu za kultywowanie pamięci o wybitnym Polaku - wielkim hetmanie polnym koronnym Stefanie Czarnieckim. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W Polsce zostało przyjęte, że osoba starsza to osoba w wieku 60 lat i więcej. Systematycznie rośnie liczba osób starszych. Na koniec 2019 r. liczba osób w wieku 60 lat i więcej przekroczyła 9 mln i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 2,1%.

W 2019 r. przeciętna emerytura miesięczna i renta brutto wypłacana z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych ukształtowała się na poziomie 2327 zł brutto. Z emerytury potrącane są podatek i składka zdrowotna, która będzie zwiększona w najbliższym czasie i wchłonie proponowaną ulgę podatkową. Zdecydowanie niższa była przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych, która w 2019 r. osiągnęła wielkość zaledwie 1292 zł.

Proces starzenia się społeczeństwa wywiera wpływ przede wszystkim na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia - starsi ludzie częściej chodzą do lekarza, korzystają z opieki społecznej. I tutaj, proszę państwa, zaczyna się jeszcze większy problem. Jeszcze kilkanaście lat temu, szczególnie na obszarach wiejskich, mieliśmy rodziny wielopokoleniowe: dziadkowie, dzieci i wnuki. Było to uwarunkowane m.in. brakiem mieszkań na rynku. Obecnie poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym, dostęp do kredytów pozwalają młodym ludziom na szybkiej usamodzielnienie się i zamieszkanie na swoim. Dziadkowie, starsi rodzice pozostają sami w swoich domach czy mieszkaniach. Dopóki są sprawni i samowystarczalni, jest dobrze, ale problem zaczyna się w momencie zachorowania czy późnej starości. Potrzebna jest 24-godzinna pomoc na dobę. Opieka nad osobami starszymi w Polsce skoncentrowana jest na domach pomocy społecznej, które są częścią systemu publicznego. Opieka tam jest na bardzo różnym poziomie, pokoje są wieloosobowe i bardziej kojarzone jest to z hospicjum niż domem opieki dla seniorów. Niewystarczająca ilość personelu, brak przestrzeni, za mało zajęć rehabilitacyjnych. Domy pomocy społecznej, jednostki państwowe stanowią 43% całkowitej liczby placówek długoterminowego pobytu osób starszych i znajduje się w nim ponad 60% łóżek. Oznacza to, że są to przeważnie duże placówki. Wielkość w tym przypadku nie zawsze idzie w parze z jakością usług. Liczba placówek, w których pacjenci muszą płacić za pobyt z własnej kieszeni, a nie za pośrednictwem Narodowego Funduszu czy emerytury, rośnie dynamicznie w ostatnich latach. Jest duże zapotrzebowanie na prywatne domy opieki dla seniorów. Dzięki temu uzyskują m.in. mniejszy pokój czy liczne udogodnienia i usługi, np. strefy relaksu i urody, apartamenty małżeńskie urządzone w formie mieszkania. Dynamiczny wzrost placówek prywatnych w ostatnich latach dotyczy głównie tzw. placówek opieki całodobowej, które stanowią większość prawie 700 prywatnych placówek działających obecnie w Polsce. Warto też zaznaczyć, że duża część osób przebywających w DPS-ie nie stanie się nigdy klientami prywatnych placówek ze względu na ograniczone środki finansowe, jakimi dysponują.

Czasami składa się na to cała rodzina, ale co w przypadku, gdy rodzina jest mała albo jej brak? Polscy seniorzy nie chcą sprawiać rodzinie kłopotu. Emerytura jest zbyt mała, by pokryć koszt pobytu, i w mieszkaniach jest mnóstwo starszych osób zamkniętych jak więźniowie. Emerytura wystarcza tylko na pokrycie kosztów mieszkania. Pan poseł Jacek Kurzępa, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Środowisko Polskiej Nauki! Braci Studencka! „Gaudeamus Igitur” rozbrzmiewa w wielu polskich miastach, wszędzie tam, gdzie istnieją szkoły wyższe, uczelnie, których powinnością jest kształcenie przyszłych elit naszej ojczyzny. Po ubiegłorocznym doświadczeniu pandemicznego nauczania wracamy do tego, co wydaje się najpiękniejszym doświadczeniem społecznym, kulturowym, poznawczym - realne spotkania ze swoimi mistrzami w wybranych dziedzinach i podążania za nimi. Żywię nadzieję, że takie emocje i takie postrzeganie relacyjności pomiędzy naukowcem, badaczem, nauczycielem akademickim a jego studentami jeszcze jest obecne, tym bardziej odczuwalne, im skuteczniej ograniczone przez reżim sanitarny i konieczny dystans. Wracamy do naszych uczelni, almae matris, co oznacza w łacinie matkę karmicielkę, której rolą jest nasycić adeptów nauki na całe ich przyszłe życie i kariery zawodowe rzetelną, obiektywną i jak najbardziej aktualną wiedzą, która spowoduje, że absolwenci będą mogli nie tylko czuć się przydatni dla społeczeństwa, ale także realnie i ich potencjał przez to społeczeństwo zostanie spożytkowane. Matka karmicielka. Któż dziś jest sfokusowany na takie postrzeganie uczelni? Oby wielu z was, nawet jeśli to pojęcie zamknięte w dyskretnym łacińskim pierwowzorze, niedostępne wielu, którzy ponownie lub po raz pierwszy wejdą w rozwarte ramiona, wrota waszych uczelni, kojarzyło się ono ze źródłem mądrości, źródłem, z którego czerpać możecie dzięki szczodrości mistrzów i ich przekonania, że domeną tego, który wie więcej, jest ponoszenie większej odpowiedzialności. Ta odpowiedzialność w murach uczelni wyższej odnosi się do trzech perspektyw: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Przeszłość, gdy jeszcze z głębi wielowiekowego dorobku naszych poprzedników, możemy, ba, musimy czerpać, korzystając z zakotwiczenia w dorobku przeszłości. Lżej nam rozumieć współczesność, mając dzięki nim sposobność wystrzegania się błędów, przed którymi ustrzegli nas swoją dociekliwością poprzednicy. Możemy zatem sięgać wyżej, śmielej, głębiej, intensywniej skupić się na współczesności, jednakże ona nas nie zadawala. Idziemy dalej tym gorliwiej, im mocniej rozumiemy, że oni, nasi uczniowie, studenci, będą funkcjonować w przyszłości. Zatem dla nich i wraz z nimi chcemy ją kształtować, do niej się przygotować. Wchodząc w przestrzeń akademii, wchodzisz w stały intelektualny flirt z czasem ci zadanym dziś, z czasem minionym, który wyznacza ci wysokie standardy uprawiania zawodu, a jednocześnie wychylony jesteś ku przyszłości, której wyobrażenie starasz się urealnić, opisać, kreować. Nie jesteś tu sam, otacza cię gęsty dorobek innych, to sukno z mądrości wieków wyścieła twoją marszrutę i poniekąd wyznacza kierunek eksploracji. Jeśli personifikujemy uczelnię jako matkę karmicielkę, to wiedz, że ofiaruje ci, studentowi, najlepsze warunki dla rozwoju. Zechciej to docenić i adekwatnie do jej szczodrości postępuj i ty. To znaczy jak? Jak dziecko kochające swoją matkę, dla której najpiękniejszym dowodem twojej miłości jest przekonanie, że syn, córka wyszli na ludzi. Mierz wysoko, nie gaś swoich aspiracji, wzmocnij je pracowitością, korzystaj z czasu ci danego, rozsmakuj się w poczuciu zadowolenia z samego siebie, w pozytywnym egoizmie maksymalnego czerpania z krynicy mądrości. Bądź dzielny, twórczy i pracowity. Gaudeamus igitur! Cieszmy się wszyscy, bo wracamy do naszych uczelni. Pan poseł Tomasz Olichwer, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Premierze! Zwracam się do pana z tego miejsca w imieniu swoim oraz innych posłów mojego okręgu wyborczego z wnioskiem o pomoc w rozwiązaniu problemu odoru, który od wielu już lat mocno utrudnia normalne funkcjonowanie mieszkańcom Zabrza. Pod koniec ubiegłego roku zakończono modernizację instalacji przetwarzania odpadów w regionalnej instalacji odpadów komunalnych firmy FCC przy ul. Cmentarnej w Zabrzu. Warta ponad 15 mln zł inwestycja obejmująca przede wszystkim hermetyzację, miała na celu wyeliminowanie smrodu w centrum miasta. Temat ten stał się na przestrzeni ostatnich lat jednym z głównych problemów społecznych. Dzieci, które uczęszczają do szkół w centrum miasta, na boiskach wdychają to cuchnące powietrze. Nie wspomnę o ludziach, którzy mieszkają lub pracują w pobliżu. To tak na powitanie. Mówię to niestety z lekką ironią. To bardzo przykry wizerunek mojego rodzinnego miasta. Problem ten poruszano wielokrotnie na sesjach rady miasta, w prasie lokalnej i regionalnej, w mediach społecznościowych również. Był on także przyczyną wielu protestów i blokad zorganizowanych na drodze dojazdowej do firmy czy przed urzędem miasta przez zabrzańskich społeczników. Niestety, przeprowadzona za aż 15 mln zł inwestycja mająca na celu wyeliminowanie przykrego zapachu nie spełniła do tej pory oczekiwanych rezultatów. Na ostatniej sesji Rady Miasta w Zabrzu prezydent miasta poinformowała, że zwróciła się do wojewody śląskiego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w Katowicach o przeprowadzenie kontroli, czy hermetyzacja została przeprowadzona w firmie FCC prawidłowo. Poprosiła również lokalnych posłów o wsparcie w tej sprawie, gdyż, jak zaznaczyła, jej kompetencje do rozwiązania tego problemu są niewystarczające ze względu na uregulowania natury prawnej. Szanowny Panie Premierze! Nie możemy pozwolić na to, żeby ta sytuacja ciągnęła się w nieskończoność. Dlatego zwracamy się do pana premiera o pomoc w rozwiązaniu tego bardzo uciążliwego dla mieszkańców problemu. Prosimy pana również o osobiste wsparcie oraz zaangażowanie odpowiednich służb w celu przeprowadzenia kontroli, czy inwestycja w firmie FCC została przeprowadzona prawidłowo, gdyż nie przyniosła do tej pory mieszkańcom Zabrza oczekiwanych efektów. Wniosek składamy też na piśmie, pod którym oprócz mnie podpisali się posłowie: Tomasz Głogowski, Krystyna Szumilas, Wanda Nowicka i Marta Golbik. Dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Podczas mojego wystąpienia chciałbym się odnieść do wczorajszego posiedzenia Sejmu, do debaty o stanie wyjątkowym. Naprawdę jest to przykre, że w sytuacji, gdzie, jako cała Izba powinniśmy się skupić na interesie narodowym, na obronie polskich granic, na współpracy. Byliśmy jako parlamentarzyści na posiedzeniach Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, również na tajnych posiedzeniach, doskonale zdawaliśmy sobie sprawę jako cała Izba z tej wielkiej odpowiedzialności, jaka na nas ciąży.

Powiem tak: Jeżeli chodzi o te głosy przeciw, to ufałem, że po tej refleksji totalnej opozycji, która chciała w pewien sposób kierować się do centrum, czyli odbudowywać elektorat i głosy utracone. Widziałem konwencję pana Donalda Tuska w Płońsku i wręcz o mało nie założyłem się z jednym z redaktorów podczas programu telewizyjnego. Uważałem, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska zagłosuje za przedłużeniem stanu wyjątkowego, bo uznałem, że to będzie taki gest, takie: sprawdzam, że 60 dni rząd Zjednoczonej Prawicy dostanie tego zaufania właśnie od totalnej opozycji. Że to będzie konkretny gest, nie, że z jednej strony jest atak na katolików, pójście w stronę skrajnej lewicy, później odbudowywanie tego elektoratu, później całowanie chleba, mówienie o wartościach. Czekałem na konkret, natomiast konkretu nie było. Było głosowanie przeciw, tylko dlatego, żeby pokazać tani populizm, czyli populizm ważniejszy niż interes państwa. Lewica zrobiła podobnie, chociaż wielu parlamentarzystów mówiło, że zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, natomiast interes polityczny wygrał z interesem państwa. 22 osoby się wstrzymały, była to Koalicja Polska. No nie da się wstrzymać w sytuacji, gdy bronimy granic. Nie wiemy, jaki głos ma ten parlamentarzysta, czy on chce być za i bronić polskich granic czy on chce być przeciw i buduje interes polityczny. Tak naprawdę jest to bardzo niebezpieczny głos, bo to jest głos, który nie wie i waży interes Polski. To jest bardzo niebezpieczne i przykre z punktu widzenia interesu państwa polskiego. Mam nadzieję, że przy podobnych głosowaniach w przyszłości Wysoka Izba w całości stanie na wysokości zadania. Nie może być podobnych sytuacji i mówienia, że ministrowie Kamiński czy Błaszczak w żaden sposób nie poinformowali parlamentarzystów. To nie jest przedszkole, że my musimy mieć wszystko napisane, narysowane i spakowany plecak. Każdy z państwa reprezentuje swoich wyborców, został wybrany, powinien być poważny i poważnie traktować ten mandat. I wydaje mi się, że w sytuacji, w której. Może te informacje nie były 100-procentowe, bo w żaden sposób nie mogły być. Żaden z posłów Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski też nie miał 100-procentowej informacji.

Niestety nie było całości ku uciesze Łukaszenki, ku uciesze reżimów, które będą na pewno wykorzystywać ten fakt i wykorzystywać poprzez swoją propagandę również krzywdę dzieci. Mam nadzieję, że w przyszłości Wysoka Izba stanie na wysokości zadania w całości. Pani poseł Magdalena Łośko, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej proponują wprowadzenie 70-procentowych podwyżek tzw. opłat nawigacyjnych dla linii lotniczych w 2022 r. Już przed pandemią stawki opłat nawigacyjnych były na polskich lotniskach niekonkurencyjne w porównaniu ze stawkami w całej Unii Europejskiej. W 2019 r. średnia opłata na europejskich lotniskach wynosiła średnio 166 euro. Z kolei w Polsce - średnia 181 euro. Proponowana podwyżka w wysokości 70% sprawi, że polskie lotniska staną się jeszcze bardziej niekonkurencyjne zarówno na rynku europejskim, jak i polskim. W pierwszej strefie, w której znajduje się lotnisko Chopina w Warszawie, w 2022 r. stawki mogą wynosić ponad 524 zł. W przypadku wszystkich pozostałych portów, które należą do drugiej strefy, opłaty będą wynosić 1347 zł. Wprowadzenie tak drastycznych podwyżek opłat nawigacyjnych może doprowadzić do załamania się rynku lotniczego w Polsce. W pierwszej kolejności w sposób znaczący zdrożeją bilety lotnicze, następnie likwidacji ulegną niektóre połączenia, a część linii całkowicie wycofa swoją ofertę z połączeń z Polski, przenosząc je na inne europejskie lotniska. Stanowi to bardzo poważne zagrożenie dla funkcjonowania polskich regionalnych portów lotniczych. Dotyczy to również dla Portu Lotniczego Bydgoszcz funkcjonującego w moim regionie. Port Lotniczy Bydgoszcz zapewnia realizację połączeń lotniczych mieszkańcom całego regionu kujawsko-pomorskiego, ale również inwestorom i turystom z zagranicy. Port stanowi bardzo ważny element rozwoju miasta i naszego regionu. Jest naszym oknem na świat. Z tego miejsca apeluję do rządu, Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o wycofanie się z 70-procentowych podwyżek opłat nawigacyjnych, które stanowią bardzo poważne zagrożenie dla funkcjonowania polskich regionalnych portów lotniczych.

Dziękuję. Pani poseł Teresa Glenc, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Do misji szkolnictwa wyższego należy nade wszystko kształcenie studentów na jak najwyższym poziomie, współtworzenie kultury narodowej w duchu wierności 1050-letniego dziedzictwa Polski. To od młodzieży zależy przyszłość Polski. Bardzo ważny elementem dla środowiska akademickiego jest opowiedzenie się za wartościami, jakimi są umiłowanie prawdy, honor i wzajemny szacunek. W szkołach oraz na uniwersytetach potrzeba pedagogów, którzy z poświęceniem, pasją i oddaniem będą przekazywać wiedzę oraz kształcić młodzież w duchu poszanowania ojczyzny oraz wartości chrześcijańskich, którzy będą dla nich punktem odniesienia na etapie wchodzenia w dorosłe życie. Powinni być autorytetami w każdej dziedzinie. Uczniom minął już pierwszy miesiąc nauki w szkołach podstawowych i średnich. Premier Mateusz Morawiecki razem z rządem dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczny powrót dzieci i młodzieży do szkół.